Wysoka Izbo! Dla 100, może 200 tys. polskich rodzin nadchodzące święta będą bardzo smutne. Będzie żal, będą łzy, będą wspomnienia o tych, których niestety zabraknie przy wigilijnym stole. Do dziś bowiem z powodu pandemii zmarło ponad 88 tys. Polaków, a w tym samym czasie odnotowano ok. 140 tys. nadmiarowych zgonów. Zmarli może i mieli poglądy polityczne, ale nie umierali jako zwolennicy tej czy innej partii. Umierali Polacy, obywatele, umierali ojcowie i matki, bracia i siostry, żony i mężowie, córki i synowie. Nie przywrócimy im życia, nie zmniejszymy żalu, którego źródłem jest ich nieobecność, ale możemy wykonać gest szacunku wobec zmarłych i okazać serdeczność ich zrozpaczonym krewnym. Gesty, także te gesty symboliczne, są ważne dla poszczególnych ludzi i dla całej naszej narodowej wspólnoty. Ważne są zawsze, ale w tym przedświątecznym czasie są zarówno potrzebne, jak i niezbędne. Musimy się pokłonić przed zmarłymi i objąć myślami naszych zasmuconych rodaków. Stać nas na to. Prawdę mówiąc, to nasz moralny i po prostu ludzki obowiązek. Mam głębokie przekonanie, że wszyscy tu to rozumiemy i czujemy. Pani Marszałek! Proszę, byśmy nisko się pochylili przed zmarłymi i przed tymi, którzy ich opłakują. Otoczmy ich szczerą modlitwą czy też serdeczną myślą.

Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, z wnioskiem formalnym pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wiemy, że inflacja i drożyzna są wam na rękę, bo wtedy puchną portfele rządu, a tracą polskie rodziny. Wzywam pana, panie premierze. Wiem, że był pan bankierem, ale wzywam pana, niech pan pochyli się nad tymi, którzy odliczają grosz do grosza.

To jest wasza odpowiedzialność. Tarcza nie działa. Dziękuję bardzo. Ponieważ padł wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Proszę. Wysoka Izbo!

Jest z nami Mejza czy go nie ma? Bo na urlopie od nicnierobienia już jest, to wiemy. Panie Premierze! Proszę o wyjaśnienie sprawy korupcji politycznej, bo oferowanie stanowisk rządowych w zamian za głosowanie nad budżetem czy kagańcem Czarnka, to jest absolutny skandal.

Dziękuję, pani poseł. Pani poseł. Nie pani jest od tego, żeby mówić, które jest poprawnie złożone, a które nie. Od tego są Komisja Etyki Poselskiej i CBA.

Wtedy, kiedy rozpatrywany jest budżet, nie można zamknąć posiedzenia Sejmu.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To jest dobra okoliczność, żeby pani marszałek wyjęła z szuflady i poddała pod głosowanie wniosek Konfederacji o to, żeby z funkcji wicemarszałka Sejmu odwołać PZPR-owskiego funkcjonariusza, gloryfikatora armii sowieckiej, a jednocześnie człowieka, który zhańbił Wysoką Izbę podczas debaty parlamentarnej. wywieszając nowy symbol lewicy, tęczowej lewicy, w miejscu, gdzie pani marszałek w tym momencie siedzi i prowadzi obrady. Jest to dobry moment, szanowni państwo, żeby poddać pod głosowanie wniosek Konfederacji o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Proszę. Bardzo dziękuję. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Te działania, które podejmują rząd i większość, są niewystarczające, zbyt płytkie i niczego nie zmienią. Specjaliści mówią, że to, co zaproponowaliście, nie jest warte... nie jest tym, czego potrzebują Polacy, a Polacy dziś potrzebują realnego wsparcia. Specjaliści mówią, że inflacja zostanie z nami na dłużej. Powiedzcie prawdę: Jak długo drożyzna zostanie z Polakami, ta drożyzna, która dzisiaj demoluje portfele Polaków? Ale chcę zapytać też o to, co z naszym projektem dotyczącym zawieszenia poboru opłaty emisyjnej, tej opłaty, którą wprowadził rząd PiS i która oznacza niestety wyższe ceny paliwa. Wy podczas posiedzenia komisji odrzuciliście ten projekt. Dziękuję, panie pośle. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Proszę.

Wysoka Izbo! Przecież kilka dni temu głosowaliście przeciwko walce polskiego rządu. o niskie ceny energii i ciepła, a teraz mówicie o drożyźnie. Drożyzna w Unii Europejskiej ma twarz Donalda Tuska i Europejskiej Partii Ludowej. To wy odpowiadacie za wysokie ceny energii i ciepła. I te obrazki pokażcie Donaldowi Tuskowi. A skoro mowa o Donaldzie Tusku, to, szanowni państwo, przeczytajcie sobie fragment mojej książki o Donaldzie Tusku. o waszej prorosyjskiej polityce. bo to wy w 2010 r. przestawialiście Polskę na wschód, to wy w 2010 r. chcieliście zabetonować rosyjskim gazem do 2037 r. Polskę.

To Donald Tusk jest najbardziej proputinowskim premierem III RP. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 (druki nr 1624 i 1819)

Szanowna Pani Marszałek! Panowie Premierzy! Wysoki Sejmie! Projekt ustawy budżetowej na rok 2022. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w dniu 14 października br. Proszę państwa, mamy bardzo ważną debatę budżetową, dlatego proszę wszystkich posłów, którzy mają inne zajęcia, o to, żeby w miarę sprawnie opuścili salę plenarną, tak żeby pan poseł mógł przedstawić sprawozdanie. Bardzo proszę.

Bardzo proszę państwa posłów o sprawne opuszczanie sali, bo to jest ważna debata. Pozwólmy panu posłowi przedstawić sprawozdanie. Proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w dniu 14 października br. 30 września rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Sejmowi projekt ustawy, po czym, zgodnie z art. 106 ust. 1 regulaminu Sejmu, został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych celem przedstawienia sprawozdania do dnia 3 grudnia br. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła projekt, kierując się przyjętym przez Prezydium Sejmu harmonogramem prac, a efektem tychże prac jest prezentowane sprawozdanie zawarte w druku sejmowym nr 1819. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 został przygotowany w warunkach niepewności i istnienia ryzyka niepomyślnego przebiegu zjawisk gospodarczych w perspektywie najbliższych kilku lat.

W projekcie rząd założył wzrost o 4,6. To jednak, jak ostatecznie ukształtuje się wzrost gospodarczy w roku przyszłym, jest jeszcze niewiadome, bowiem trudno przewidzieć nie tylko rozwój pandemii, ale także reakcje na nią rządów oraz przedsiębiorców z różnych państw, w tym zwłaszcza u naszych głównych partnerów handlowych. Trudno też przewidzieć rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

Rząd zakłada także dług sektora rządowego i samorządowego na poziomie 56,6% PKB, a ostatnia prognoza Komisji wskazuje na wielkość niższą, wynoszącą 51% PKB. Można zatem uznać, iż polskie finanse publiczne odpowiadają właściwie na obecną trudną sytuację po pandemii COVID-19 i nie powinny być zagrożeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego w dłuższym okresie.

Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych dotyczące w szczególności zastosowania skorygowanej okresowo stabilizującej reguły wydatkowej. Kwota wydatków na rok 2022 została powiększona o 1/3 prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrecjonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymywanie skutków epidemii w 2020 r. i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nimi podmiotów. Ponadto w kwocie wydatków na rok 2022 uwzględniono aktualizacje dotychczas wprowadzonych i skutki nowych działań dyskrecjonalnych w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy mogę prosić państwa posłów o wyciszenie rozmów? Dziękuję bardzo, panie marszałku.

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zapewniono środki m.in.: na finansowanie programu „Rodzina 500+”; na realizację zobowiązania rządu do zwiększenia w roku 2022 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB; na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem państwowej waloryzacji na poziomie 104,89%; na finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego oraz na realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia przyszłego roku; na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2% PKB; na finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej; na realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej; na realizację inwestycji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na odbudowę Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla; na finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, dopłaty do paliwa rolniczego. Projekt budżetu na rok 2022 opracowano przy zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetów rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej. Chciałbym przybliżyć szczegółowe prace Komisji Finansów Publicznych, jakie odbyły się w ramach pierwszego czytania i doprowadziły do przygotowania sprawozdania z prac tejże komisji. Komisja Finansów Publicznych na swoich posiedzeniach rozpatrywała własne części budżetowe.

Posłowie przedstawiali najważniejsze informacje z dyskusji na posiedzeniach innych komisji. Szczególne zainteresowanie posłów budziły m.in. kwestie dotyczące założeń makroekonomicznych budżetu, w tym w odniesieniu do inflacji, deficytu i długu publicznego, oraz kwestie dotyczące zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w różnych jednostkach. Jeśli chodzi o prace innych komisji, do których skierowany był do rozpatrzenia projekt ustawy budżetowej, to należy wskazać, iż komisje sejmowe przedłożyły Komisji Finansów Publicznych łącznie 25 opinii. Były to opinie pozytywne. Jedynie w dwóch opiniach komisji zawarto poprawki. Do części opinii komisji dołączono zdania odrębne, było ich łącznie 32. Scharakteryzuję krótko poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok przyszły. Zgłoszonych zostało łącznie 599 poprawek. 132 poprawki dotyczyły dochodów budżetu państwa, zawartych w załączniku nr 1, i wskazywały na potrzebę podniesienia dochodów podatkowych, z podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, po to aby możliwe było sfinansowanie określonych wydatków. 456 poprawek dotyczyło wydatków budżetu państwa. W poprawkach tych odwoływano się do pomniejszenia wydatków m.in. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Funduszu Kościelnego, a także wydatków przewidzianych na obronę narodową, na obsługę długu Skarbu Państwa oraz na rezerwy celowe.

Komisja nie przyjęła 544 poprawek, z których zdecydowana większość została ponownie zgłoszona jako wnioski mniejszości - jest ich 498, załączono je do sprawozdania komisji. Komisja nie zaakceptowała wszystkich tych poprawek, co do których opinię negatywną wyraził przedstawiciel rządu. Należy wskazać, iż poprawki te nie miały istotnego wpływu na wielkości ogólne budżetu państwa, bowiem ogólna kwota dochodów i wydatków budżetu państwa nie uległa zmianom. Ta opinia dotyczy tych poprawek, które zostały przyjęte, a nie wszystkich poprawek, które zostały złożone. Zauważyć można, iż zmniejszone zostały wydatki niektórych jednostek mających autonomię budżetową, w tym: Kancelarii Senatu - o 7%, co wiąże się głównie z tym, że o 10 mln zł zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadań w zakresie sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, ponieważ wydatki na ten cel ujęto w innej części budżetu; Sądu Najwyższego - o 5%; Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego - o 4%; Państwowej Inspekcji Pracy - o 3%; Instytutu Pamięci Narodowej, rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka - o 1%. Zmniejszeniu uległy także wydatki sądów powszechnych i wydatki ujęte w rezerwach celowych - o 3%. Szanowni Państwo!

Chciałem podziękować wszystkim paniom i panom posłom, którzy uczestniczyli w pracach komisji tematycznych i w pracach Komisji Finansów Publicznych. Chciałem podziękować posłom referentom, koreferentom za dobre przygotowanie. Dziękuję za atmosferę tej pracy. Przede wszystkim zgodnie z wolą pani marszałek Sejmu byliśmy w stanie dostarczyć sprawozdanie z naszych prac we właściwym czasie, respektując harmonogram prac. Dziękuję też wszystkim przedstawicielom instytucji rządowych, instytucji konstytucyjnych za ich przygotowanie i merytoryczny wkład w debatę. Dziękuję tym wszystkim, którzy w tej debacie brali czynny udział. Cóż, pozostaje mi stwierdzić, że Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022, wraz ze stanowiskami przekazanymi przez właściwe komisje, wnosi o uchwalenie załączonego projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Bardzo dziękuję. Sejm ustalił w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego podział czasu pomiędzy kluby i koła, w zależności od ich wielkości, w granicach od 49 do 4 minut, tj. debatę krótką. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Wiesław Janczyk, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! Co można powiedzieć o budżecie, o którym już tyle powiedziano? To dokument, który jak co roku jest drogowskazem dla biznesu, dla ludzi, dla administracji, dla wszystkich grup społecznych i zawodowych, dla grup branżowych.

Dzisiaj ludzi w Polsce najbardziej interesuje kilka tematów. Według badań opinii społecznej jest to kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też bezpieczeństwa granic.

Kolejnym tematem, który w związku z pandemią COVID bardzo zajmuje naszych obywateli, jest kwestia zdrowia.

Realizujemy ten budżet nie bez przeszkód, bo COVID spowodował wzrost czynników zewnętrznych, które przekładają się na wzrost inflacji.

Będziemy działać odważnie i reagować elastycznie na potrzeby naszego społeczeństwa, zwłaszcza ludzi mniej zamożnych, którym będziemy starali się dać podstawę do funkcjonowania. Nie zapominajmy też o tym, że obniżając w tym pakiecie antyinflacyjnym akcyzę, opłatę paliwową, VAT, doprowadzamy do tego, że wszyscy, którzy dzisiaj pracują w przemyśle transportowym, ale także właściciele firm, wszyscy, będą beneficjentami tej pomocy państwa. Szanowni Państwo! Budżet ma być realizowany w warunkach niepewnych dostaw i drastycznego wzrostu cen światowych nośników energii, surowców, prądu, gazu, ropy naftowej, frachtu. Jaką odpowiedź niesie ten budżet dla tych, którzy chcą optymizmu, którzy troszczą się o przyszłość? Nie hamujemy wzrostu, nie hamujemy wzrostu płac, rosną emerytury, rosną renty. Proszę państwa, skonstruowaliśmy ten budżet, domykając go z niewielkim deficytem i nie wyprzedajemy polskich sreber rodowych, nie wyprzedajemy polskich firm, a nasi poprzednicy robili to prawie za każdym razem. Szanowni Państwo! Nie hamujemy inwestycji. Polski Ład to kwota ponad 100 mld zł, która zasila dzisiaj kasy jednostek samorządu terytorialnego - tam są przeznaczane potężne nakłady na infrastrukturę komunalną według uznania samorządów, według priorytetów, jakie one same ustalają. Utrzymujemy wydatki społeczne, utrzymujemy program 500+, program „Dobry start”, program „Maluch+”, utrzymujemy świadczenia dla pań, które urodziły czwórkę i więcej dzieci. O wydatkach na armię wspomniałem, na zbrojenia. Jeśli chodzi o zdrowie, realizujemy umowy społeczne - kwota przeznaczona na wydatki na zdrowie to 5,75% PKB. Chronimy miejsca pracy. Wiecie państwo, ile przeznaczyliśmy w roku COVID-owym na ochronę tychże miejsc pracy? Wiemy, że trudniej jest odtworzyć miejsca pracy, niż je utrzymać. Chcemy obniżać bezrobocie i to bezrobocie obniżyliśmy w porównaniu z naszymi poprzednikami o milion osób. Utrzymujemy zerowy PIT dla młodych ludzi do 26. roku życia, wielu z nich z tego powodu nie wyjeżdża za granicę, bo mają chociażby na to, żeby opłacić mieszkanie tam, gdzie dostają pracę.

O innych częściach budżetowych szczegółowo powiedzą moi koledzy w ramach przeznaczonego w debacie czasu dla klubu Prawo i Sprawiedliwość, nie chcę wchodzić w ich rolę.

Proszę państwa, chcę powiedzieć, że doprowadziliśmy do tego, że udział walut w naszych zobowiązaniach kredytowych spadł poniżej 25% i to zadłużenie jest uwolnione od tego czynnika ryzyka różnic kursowych, które było zmorą przez dziesięciolecia przy finansowaniu długu publicznego. Dług sektora general government wyniesie 56,6% PKB, chociaż jak czytałem w sprawozdaniu komisji dane Komisji Europejskiej, możemy być nastawieni optymistycznie, że będzie on trochę mniejszy.

Już nie będę przypominał, ile ona wynosiła jeszcze nie tak dawno. Te elementy, które pozwoliły na konstrukcję budżetu zrównoważonego, który przynieśliśmy w 2020 r., owocują dzisiaj. Owocuje reforma Krajowej Administracji Skarbowej, uszczelnienie celne granicy, wprowadzenie systemu SENT 1, SENT 2, SENT 3, odważne wprowadzenie regulacji zawartych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich, wprowadzenie komitetów audytu, rozdzielenie możliwości świadczenia usług doradczych i audytorskich przez te same wielkie podmioty. Bez kontroli, bez udziału kontrolerów Krajowej Administracji Skarbowej możemy liczyć na większe dochody do budżetu państwa. Z dumą chcę powiedzieć jedno: wspieram rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Chcę powiedzieć to z dumą i myślę, że nikt nie potrafi znaleźć argumentów, żeby temu zaprzeczyć. Ale jest tam jeszcze jeden element, który my przeoraliśmy i zmieniliśmy w sposób drastyczny: świadczenia dla rodziny bez dochodu. Myślę, że ci, którzy tę tablicę wtedy tworzyli, nawet nie myśleli o tym, że takie preferencje będą skierowane ze strony państwa do każdego obywatela. Przychodzimy z budżetem, który będzie wspierał wzrost gospodarczy i daje realną szansę na godne życie dla każdego Polaka. Proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Szlachtę. Pani poseł Izabela Leszczyna.

Dziękuję, panie marszałku. Tak, to równanie pokazuje cały ten wasz przyszłoroczny budżet - budżet proinflacyjny, budżet rozpasany i wreszcie budżet fasadowy. Wczoraj w wolnym, demokratycznym Senacie odbyła się debata o przejrzystości finansów publicznych, debata, która nie mogłaby się odbyć w Sejmie zarządzanym przez panią marszałek Witek. Wszyscy są głęboko zaniepokojeni wyprowadzaniem wydatków poza budżet i brakiem kontroli nad publicznymi pieniędzmi, brakiem kontroli Sejmu i brakiem kontroli opinii publicznej. W kontekście braku przejrzystości, w kontekście fasadowości tego budżetu potwierdzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli zasadne wydaje się pytanie, czy w ogóle warto rozmawiać o tej szczątkowej części finansów publicznych. Bo w gruncie rzeczy wprowadzamy tylko opinię publiczną w błąd. Dlaczego budżet jest fasadowy, rozpasany i proinflacyjny? Bo wskaźniki makroekonomiczne w tym projekcie są wzięte z sufitu, są jak rzut kulą w płot.

My będziemy przyjmować sprawozdanie z wykonania budżetu w czasie, kiedy rozpasanie rządowej konsumpcji będzie trwało w najlepsze. Budżet jest fasadowy, bo z limitu wydatków, stabilizującej reguły wydatkowej wyjęliście fundusz COVID-owy i to wszystko, co jest w BGK. To właściwie po co nam taka reguła? To o czym my tu rozmawiamy? Po co? Wam to jest potrzebne, ja rozumiem. Ale my nie będziemy w tym uczestniczyć. Do reguły finansów minister włożył jakieś lewe dowody, żeby jeszcze bardziej poszerzyć sobie przestrzeń wydawania publicznego grosza. Dług poza kontrolą parlamentu, poza budżetem - w przyszłym roku to będzie 350 mld zł. Jak pan przewodniczący może w ogóle mówić o niskim deficycie? 350 mld zł poza kontrolą budżetu, a deficyt, jaki musieliście zaraportować do Komisji Europejskiej, to przecież 143 mld. Dlaczego o tym nie mówicie tu, z mównicy sejmowej? Nadal rozdajecie obligacje, rozdajecie je telewizji Kurskiego. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że przyszły demokratyczny rząd będzie płacił za propagandę Kurskiego, za estetyczne bezguście tej telewizji i za etyczny upadek telewizji propagandowej, PiS-owskiej.

Rozpasanie państwa w czasie pandemii jest po prostu niemoralne. Uwaga, warto to pamiętać. Kłamią, że przeznaczają 5,75% PKB na zdrowie. Tak naprawdę w relacji do przyszłorocznego PKB, ale wyliczonego na podstawie prawdziwych wskaźników makroekonomicznych, a nie tych wymyślonych przez specjalistów z NBP i Ministerstwa Finansów, na zdrowie przeznaczą 4,89% PKB w drugim roku pandemii. 4,89%, z czego, uwaga, wszystko to są właściwie składki, które wpłacacie państwo do Narodowego Funduszu Zdrowia, a z budżetu idzie tylko 0,8%.

Dlatego że PiS zdradził Polaków. I zdradził Polskę. Mieli do wyboru ponad 20 mld zł zaliczki już w tym roku i kolejne transze z Krajowego Planu Odbudowy w przyszłym roku, żeby zapewnić środki na inwestycje i na prawdziwy dobrobyt obywateli. Wybrali partyjne sądy, zemstę na odważnych, niezawisłych sędziach i likwidację autonomii samorządów. Że klub Koalicji Obywatelskiej miał rację, kiedy przy głosowaniu nad Funduszem Odbudowy chciał wpisać obecność samorządów w komitecie monitorującym. Bo dzisiaj to jest jeden z warunków Komisji Europejskiej, żebyśmy w ogóle te pieniądze dostali. Ponieważ nie możemy na te pieniądze liczyć, ten budżet musi stać się bardziej inwestycyjny, a mniej rozpasany. Jeśli minister finansów uzna, że poprawki przedstawione przez panią Zofię Czernow dostaną pozytywną rekomendację i będą przyjęte, to być może wycofamy wniosek o odrzucenie tego budżetu w drugim czytaniu, który za chwilę na ręce pana marszałka złożę. To jest wasz budżet. Bardzo dziękuję, pani poseł. Teraz głos zabierze w imieniu klubu Lewicy pan poseł Dariusz

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście przedstawiony projekt budżetu jest projektem, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To swego rodzaju bajki z mchu i paproci, które rząd Prawa i Sprawiedliwości pisze nam w kolejnych budżetach od 2015 r.

Rzecz kolejna. Planujecie 86 mld środków z Unii Europejskiej. Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście środki z Unii Europejskiej się pojawią, bo przecież doskonale wiemy, że raczej w tym roku nie ma żadnych szans na to, ażeby środki z Unii Europejskiej się pojawiły. Aby była jasność, możecie zaklinać rzeczywistość, ale to jest tylko wasza wina, że dzisiaj wszyscy jako Polacy cierpimy z tego powodu, że tych środków nie otrzymujemy.

I żeby była jasność: wszyscy na tym cierpimy. Przyrost zadłużenia planujecie na poziomie 140 mld zł. 140 mld zł. Przypomnę, że jeżeli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli i o kontrolę, która była w tym roku prowadzona, to Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że ok. 290 mld zł jest wydatkowane poza budżetem.

Z czego to wynika?

Natomiast zdziwieni jesteśmy, że planuje się zmniejszenie dochodów, jeżeli chodzi o akcyzę, bo przecież na tej sali debatujemy nad ustawą, która podnosi podatek akcyzowy, w związku z czym konia z rzędem temu, kto jest w stanie wyjaśnić, jakim cudem mają się zmniejszyć wpływy z akcyzy w roku 2022. Zmniejszają się wpływy z CIT-u, zmniejszają się wpływy z PIT-u.

Kluczową sprawą są inwestycje. Co do tego nie ma wątpliwości, że mamy dzisiaj najniższy wzrost inwestycji w stosunku do PKB właściwie od początku transformacji, to jest poziom 16%.

To jest zdecydowanie za mało. Kwestie wydatków majątkowych na drogi, kwestie subwencji dla samorządów.

Prawie 40 mld zostawiliście sobie na rezerwy celowe. Ano mamy np. rezerwę na zwiększenie środków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych. Czyli znowu będziecie odwoływać po to, żeby dać komuś zarobić.

Mamy rezerwę na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania - 3 mld zł.

W tej sytuacji klub Lewicy przedstawia swoje poprawki. W przypadku ich nieprzyjęcia będziemy głosowali przeciwko przyjęciu ustawy budżetowej. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Czesława Siekierskiego, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Szanowni Państwo!

Podobna sytuacja jest w przypadku założeń odnośnie do deficytu budżetowego. Znaczna część wydatków jest wyprowadzona poza budżet.

Obligacje polskiego rządu tracą na wartości najszybciej od kilku lat. Przechodzę do Polskiego Ładu. Polski Ład to przede wszystkim duża niepewność, chaos, komplikacja systemu podatkowego, znaczny wzrost podatków dla firm oraz trwałe obniżenie dochodów samorządów. A więc - firmy i samorządy.

Polski Ład wpłynie nie tylko na podwyższenie kosztów wytwarzania w procesie produkcji, ale także na wzrost kosztów administracyjnych, księgowych i innych, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Wzrost kosztów wytwarzania, głównie ze względu na wzrost kosztów paliw, energii, przełoży się na wzrost cen towarów i usług. Mówią, że zatowarowanie firmy to wzrost kosztów o 100%. Taka jest sytuacja, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. W podobnej sytuacji są rolnicy.

O drożyźnie była tu mowa. Pakiet antyinflacyjny, osłonowy. Wspomniane przez pana przewodniczącego 10 mld to dużo, dużo za mało. Wreszcie trzeba się zastanowić, jak można było nie sięgnąć, nie skorzystać z pieniędzy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, które leżały na stole, były dostępne. Budżet to nie tylko liczby. Pomyślmy o tych najbiedniejszych. Po drugie, wczoraj jeden z wyborców w czasie rozmowy mówi: panie pośle, nie ma za co żyć. Ja to pytanie w imieniu tego wyborcy, a myślę, że też w imieniu milionów wyborców, kieruję do pana premiera: Za co żyć? Trudno, aby w takiej sytuacji popierać taki budżet. Dlatego proponujemy jako Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe poprawki.

Wiemy, jaka sytuacja jest w szpitalach, szczególnie w tych powiatowych, ale nie tylko. Samorządy ponoszą ogromne koszty finansowania edukacji, szczególnie jeśli chodzi o płace dla nauczycieli. To nie pozwala im realizować innych inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Po trzecie, mamy trzy poprawki sfinansowane z różnych źródeł, jeśli chodzi o utworzenie rezerwy celowej na fundusz klęskowy dla rolników. O trudnej sytuacji rolników mówiłem. Wymagają oni wsparcia, bo to jest problem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich. Kolejna poprawka dotyczy utworzenia rezerwy na „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”

Wreszcie także środki na program antysmogowy.

Proszę teraz pana posła Jakuba Kuleszę o to, aby przedstawił stanowisko koła Konfederacja. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zdradzę państwu sekret: perpetuum mobile nie działa, nie istnieje ani w fizyce klasycznej, ani tym bardziej w ekonomii. Dobrobyt nie bierze się z dotacji publicznych, dobrobyt bierze się z ciężkiej pracy obywateli, a od przelewania publicznych pieniędzy z konta na konto, z funduszu na fundusz, z budżetu do funduszy pozabudżetowych i na odwrót ten dobrobyt po prostu nie powstanie. Obywatele na tym całym mechanizmie mogą jedynie stracić, ponieważ państwa system jest dziurawy i po prostu przecieka, tak jak każdy publiczny system finansów. Szanowni Państwo! Ustawa, nad którą debatujemy, to najważniejsza ustawa w całym roku. To jest ustawa budżetowa, a państwo - mówię o większości sejmowej - ustalili, by nad tą ustawą przeprowadzić debatę krótką, czyli żeby np. kołu Konfederacji przypadło tylko 5 minut.

Naprawdę za dużo, za dużo. Jakie są państwa założenia? Sprawdźmy.

Na początku 2020 r. prezes Glapiński powiedział, że PKB urośnie o 2%. Na koniec roku okazało się, że PKB skurczyło się o 2,7%. Żeby pomylić się o 4,7% we wzroście PKB, to naprawdę nie trzeba być ekonomistą. W kwietniu 2020 r. prezes NBP straszył nas deflacją, że ceny będą spadać, że nie grozi nam drożyzna. Jak było, wszyscy widzieliśmy. W styczniu 2021 r. usłyszeliśmy, że inflacja, czyli drożyzna, będzie spadać i dalej grozi nam deflacja.

Już w czerwcu osiągnęła 4,5% i wtedy usłyszeliśmy od prezesa NBP, że to jest absolutny szczyt, a dzisiaj inflacja rok do roku wynosi 7,7%. Tyle wychodzi z państwa planów. I to nie jest tak, że państwo się pomylili. To wynika z tego, jak państwo próbują temu zapobiegać. Otóż państwo postanowili w zeszłym roku, że na 3 miesiące zamkną gospodarkę, a obywatele tego nie odczują, bo państwo stworzą dotacje publiczne.

Pieniądze się wpompuje i jakoś to będzie. I za państwa działanie, za zamknięcie gospodarki - ten dobrobyt nie bierze się z powietrza - zapłacą wszyscy obywatele. Rzeczywiście wszyscy za to płacimy ogromną drożyzną, inflacją na poziomie 7,7%. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że rząd, który myli się tak często w tak ważnych sprawach. Dziękuję bardzo. Stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 przedstawi pani poseł Paulina Hennig-Kloska. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Po wielu tygodniach pracy w Komisji Finansów Publicznych ten budżet można podsumować w zasadzie jednym zdaniem: zamiast przeznaczyć pieniądze na ratowanie zdrowia i życia Polek i Polaków, wolicie je przeznaczyć na telewizję Kurskiego i ministerstwo sportu, dla Mejzy. Czeka nas rok inflacji, a drożyzna będzie wywoływać u Polaków bezsenność. Tarcza nie zadziała - to już wiadomo. Inflacja dalej będzie utrzymywać się na poziomie blisko 7% w ujęciu rocznym. Ceny będą rosnąć przynajmniej do wiosny, jeśli nie dłużej. Przyjmuje się, że nawet w 2023 r. ceny będą rosnąć na poziomie nieakceptowalnym, trudnym dla portfeli Polek i Polaków. To są najnowsze prognozy. Jak reaguje rząd na te prognozy? Co to takiego? Nieudolna próba obniżenia rachunków za energię czy ogrzewanie mieszkania.

Do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły już wnioski o zmianę taryf dla gospodarstw domowych. Skala wnioskowanych podwyżek to 40%. Szacuje się, że skończymy na 20-procentowej podwyżce z początkiem roku.

By rozwiązać problem rosnących cen prądu, musimy przede wszystkim zacząć inwestować w energetykę, w rozwój odnawialnych źródeł energii, w rozwój sieci energetycznych, budowę magazynów energii.

Wy te pieniądze po prostu przepalacie w piecu na węgiel. Nie potraficie też zadbać o interesy Polek i Polaków w Brukseli. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, jak można było w tak trudnych czasach, przy tak rozchwianej gospodarce rynkowej doprowadzić do tego, że ta zaliczka do końca roku nie wpłynie na nasz rachunek.

Będziemy musieli na te inwestycje uruchamiać prefinansowanie, a więc finansowanie z kredytu, co dalej będzie pobudzało inflację, a warunkiem opanowania drastycznego wzrostu cen jest opanowanie wzrostu długu. Dalej nas zadłużacie poza budżetem i poza kontrolą parlamentu, a więc również poza regułami gry. Obchodzicie reguły gry, obchodzicie regułę wydatkową, obchodzicie kontrolę parlamentu. Dobrze wiecie, że naginacie prawo, bo ustawa okołobudżetowa jest pełna różnych wydatków, które będą finansowane z pieniędzy pozabudżetowych, z obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób po prostu wprowadzacie obywateli w błąd. Fundusz Medyczny miał dać miliardy złotych na zdrowie.

W tym roku mieliście wydać ponad 4 mld zł, z budżetu przeznaczyliście do funduszu niecałe 2 mld zł, a wydano, uwaga, 171 mln zł. Tak naprawdę utrudniliście dostęp do świadczeń medycznych, przesuwając zadania do Funduszu Medycznego i nie uruchamiając żadnych pieniędzy i żadnych konkursów.

Jaki jest efekt dla obywateli? Np. chorzy na mukowiscydozę mogliby przyjąć dostępne na świecie leki, które hamują rozwój tej choroby, ale lek ten jest dla nich zbyt drogi, a państwo go po prostu nie refunduje. Mimo że obiecywaliście refundację od 1 stycznia, to już wiemy, że jej nie będzie. Ten lek jest refundowany praktycznie w całej Europie Zachodniej: w Niemczech, we Francji, w Austrii, we Włoszech, również w Czechach i na Słowacji, ale nie w Polsce. A dlaczego?

To nie jest budżet dla ludzi. Będziemy wnioskować o odrzucenie tego budżetu w drugim czytaniu. Dziękuję bardzo. Teraz pani poseł Agnieszka Ścigaj przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Nie wiemy, jak one są wydawane, ponieważ są poza ustawą budżetową. Nie wiemy również, jak wydawane było 100 mld zł.

To ukrywanie, kreatywna księgowość i wspomniane zniesienie reguły wydatkowej na inwestycje. Brak jest reform poszczególnych instytucji.

Kolejne pokolenia nie będą mieścić się w systemie opartym na zastępowalności, nie będą mieć dobrych emerytur.

Mówiono nam, że nie możemy zarabiać tyle, ile zarabiają nasi rówieśnicy na Zachodzie, dlatego że spłacamy długi po komunie. Przecież tak właśnie będzie.

Zajmijmy się pracą nad polskimi wydatkami, nad polskim budżetem, żeby on był przejrzysty, klarowny, zadaniowy. To jest rozwiązanie.

Zacznijmy patrzeć na budżet państwa jak na budżet własnego gospodarstwa domowego.

Proszę teraz pana posła Andrzeja Szlachtę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!

Była ona większa o 40% do podobnej subwencji z roku 2015. Ta wysoka subwencja i duże środki finansowe kierowane były z budżetu państwa na inwestycje samorządowe.

To świadczy o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dobrze troszczy się o polskie samorządy.

Dla gmin popegeerowskich, o których zapomnieli wszyscy rządzący poprzednio, przeznaczono ponad 340 mln zł. Świadczy to o trosce rządu o polskie samorządy.

W pierwszym roku rządów koalicji PO-PSL subwencja oświatowa wynosiła niewiele ponad 30 mld zł.

Zadania w obszarze oświaty i wychowania realizowane są przez osiem ministerstw, wojewodów i fundusz pomocy kultury.

Ważnym zadaniem rządu jest również realizacja celu długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także kształcenie na poziomie wyższym. Skonsolidowana kwota wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi w budżecie na 2022 r. 32 850 mln zł, z czego na szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczono ponad 27 mld zł, a na badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom - blisko 6 mld zł. Największą pozycję w dziale 730: Szkolnictwo wyższe i nauka stanowią wydatki na działalność dydaktyczną i badawczą, tj. kwota 17 mld zł.

Tak dużych nakładów budżetowych na obiekty szkolnictwa wyższego i szpitale kliniczne nie było nigdy dotąd, chodzi o ostatnie kilkanaście lat. Bardzo dziękuję panu posłowi.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dziś odbywa się bardzo ważna debata o finansach państwa, o bezpieczeństwie finansów publicznych, o pieniądzach Polaków. Gdzie jest konstytucyjny minister finansów? Brak tych osób jest wymowny, proszę państwa. Rozmawiamy o tym, jak zostaną wykorzystane pieniądze Polaków. Chodzi o sprostanie wysokiej rangi wyzwaniom społecznym i gospodarczym, jak pandemia, która zbiera obfite żniwo śmierci, inflacja i związana z tym drożyzna, a także brak skuteczności w zwalczaniu smogu. Niestety problemy te nie są skutecznie rozwiązywane. Dlatego klub Koalicja Obywatelska zgłasza poprawki do projektu budżetu. Po pierwsze, żądamy, podkreślam: żądamy zwiększenia wydatków na zdrowie o 20 mld zł, [[Oklaski]] aby zapobiec katastrofie w ochronie zdrowia.

Jest to jeden z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników. Źródłem finansowania będzie tu podatek inflacyjny wyjęty z kieszeni Polaków. Polacy żądają zwrotu swoich pieniędzy, bo chcą się leczyć, leczyć swoich bliski i żyć, po prostu żyć. Na transformację energetyczną proponujemy 10 mld zł, [[Oklaski]] gdyż jest ona nie tylko nakazem chwili powstałym z powodu obniżania się mocy przestarzałych elektrowni, lecz jednocześnie jest to też ważne i skuteczne działanie antyinflacyjne. W przeciwnym razie czeka nas dalszy gwałtowny wzrost cen energii i konieczność kupowania jej na zewnętrznych rynkach.

Potrzebna jest zdecydowana walka ze smogiem, a dotychczasowe programy są niestety dziurawe, jak choćby ten dotyczący wsparcia wymiany ogrzewania w budynkach wielomieszkaniowych.

Już najwyższy czas, aby nauczyciele mieli godne wynagrodzenie.

Źródłem finansowania będą pieniądze, które są w budżecie, ale ukryte w różnych rezerwach.

Wynagrodzenia sfery budżetowej w ostatnim czasie uległy znacznemu rozwarstwieniu. Aby choć częściowo to zniwelować, konieczne jest - i o to wnioskujemy - zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych sądów i prokuratur o 390 mln zł, wzrost płac dla pracowników cywilnych w Policji i Straży Granicznej. Czas najwyższy się upomnieć o tych pracowników. Rząd nie reaguje, Wysoko Izbo, na lawinowo narastające problemy na wsi, w tym szczególnie kilkakrotny wzrost cen nawozów, który bezpośrednio przekłada się na rosnące ceny żywności i drożyznę. Rolnicy muszą otrzymać pomoc, aby ograniczyć inflację. Proponujemy 800 mln zł na dopłaty dla rolników do zakupu nawozów [[Oklaski]] oraz zwiększenie kwoty o 200 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Te pieniądze w budżecie już były, ale PiS na ostatnim posiedzeniu komisji finansów to zabrał. Niestety taka jest prawda. Jest wiele problemów społecznych, które można rozwiązać przy stosunkowo niskich nakładach.

To naprawdę słabo działa, [[Oklaski]] a młodzież popełnia samobójstwa. Jak długo to będzie trwało? Na co czekamy, Wysoka Izbo? Bardzo ważna poprawka, która jest nie tylko potrzebnym wsparciem, ale także wyrazem solidarności z gminami objętymi strefą stanu wyjątkowego. Proponujemy na ten cel 280 mln zł, po 10 dla każdej gminy. Te gminy tych pieniędzy potrzebują. Kończąc, zachęcam wszystkich posłów do poparcia tych ważnych i słusznych poprawek, które będzie świadczyło o tym, że szanujemy pieniądze Polaków i liczymy się z ich pilnymi potrzebami i oczekiwaniami. Składamy również dwie poprawki do części tekstowej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem zapytać, czy wynika to może z przeoczenia, czy faktycznie w proponowanych poprawkach do budżetu brakuje poprawki posłów PiS-u, którzy złożyli przecież uchwałę w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 i podjęcia działań na rzecz reformy poprzez likwidację praw do obrotu uprawnieniami. Rozumiem, że wszyscy posłowie PiS-u podpisani pod tamtą uchwałą zawnioskują o odrzucenie projektu budżetu, gdyż w przeciwnym razie będzie to przyznanie się, że ma ona charakter wybitnie propagandowy. Jej celem nie jest, tak jak napisano w uzasadnieniu, ochrona polskich interesów, a przeciwnie – będzie to wyrażenie zgody na spekulacyjne operacje finansowe rządu, powodujące drenaż polskiego podatnika. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Paszyka o kontynuowanie wystąpienia w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska.

Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiaj to powoduje, że pieniędzy, na które wyłączny wpływ mają samorządy, jest bardzo niewiele. Oczywiście próbujecie to maskować wsparciem, które jest dedykowane tym inwestycjom, które uzna wojewoda lub inny namiestnik władzy, natomiast nie o to chodzi w samorządzie.

Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska wnoszę kolejne poprawki regionalne, wychodzące naprzeciw właśnie rzeczywistym potrzebom samorządowym, które niestety w wyniku złej polityki regionalnej państwa nie mogą być spełnione. Uważamy, że właśnie w tym kontekście budżet państwa jest niestety niewystarczający, jeśli chodzi o realizowanie dobrej polityki regionalnej przez polskie samorządy. Bardzo dziękuję panu posłowi. Teraz głos zabierze pan poseł Robert Winnicki w imieniu Konfederacji. Wysoka Izbo! Ten budżet się nie zepnie. Ten budżet się nie zepnie w 2022 r., o ile Polska nie przystąpi do radykalnej walki z inflacją, z drożyzną, z procesami gospodarczymi wykańczającymi nasz przemysł, wykańczającymi również nasze gospodarstwa domowe; jeśli Polska nie wypowie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej; nie zatrzyma szalonego wzrostu cen prądu; nie zatrzyma szalonego wzrostu cen gazu i wszelkich innych nośników energetycznych poprzez radykalną obniżkę podatków. Tego nie ma w tym budżecie. To jest budżet przetrwania, a nie budżet rozwoju. Domagamy się radykalnych kroków, które zmniejszą koszty życia, ale też dadzą rozwój naszej gospodarce. To jest postulat Konfederacji i należy wreszcie (Dzwonek) na forum Unii Europejskiej zacząć walczyć o nasze interesy. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Ryszard Galla, poseł niezrzeszony. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powiedziałbym, wyjątkowej procedury. Właśnie doświadczam pewnych działań ukierunkowanych na, powiedziałbym, antyniemieckość. Już w pierwszym czytaniu mieliśmy kilka poprawek złożonych do budżetu, które miały na celu ograniczenie środków na funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Na szczęście, szanowni państwo, te poprawki zostały odrzucone w komisjach merytorycznych, a przede wszystkim w Komisji Finansów Publicznych, za co chciałbym moim koleżankom i kolegom z komisji serdecznie podziękować. Natomiast wczoraj dowiedziałem się, że to nie koniec, że jest złożona poprawka, która ma akceptację ministerstwa edukacji, panie ministrze, o kwotę 39 800 tys. zł obniżająca część oświatową subwencji ogólnej dla samorządów. Bo system państwo znacie, wiecie, jaki jest - nie ma pieniędzy przeznaczonych na poszczególne mniejszości, nie ma takiej możliwości.

Nie mam nic przeciwko temu, aby dokładać pieniądze na naukę języka polskiego w Niemczech.

Szanowni państwo, w mojej ocenie jest to rzecz nie do wykonania. Samorządy przeznaczają te środki na realizację zadań w szkole, czyli dostają je dyrektorzy szkół, pokrywają koszty, chociażby nawet związane z zatrudnieniem nauczycieli. A więc tak naprawdę krzywdzimy dzieci. W środowisku mniejszości niemieckiej jest ponad 48 tys., prawie 50 tys. dzieci, obywateli polskich, dzieci, które mają prawo, zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych czy też zgodnie z ustawą o oświacie, uczyć się tego języka. I dzisiaj ktoś proponuje zabrać te środki. Szanowni Państwo! Powiem tak. W ostatnim czasie dużo słyszymy na temat właśnie stosowania symetrii. Nikt, kto jest zainteresowany funkcjonowaniem mniejszości, środowiska mniejszości nie uznają takich zasad. A tutaj, żeby rozmawiać dyplomatycznie ze stroną niemiecką, stosuje się pewnego rodzaju zakładnictwo, bo, przepraszam bardzo, ale ja i moje środowisko czujemy się zakładnikami. My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, lojalni patrioci zamieszkujący ziemie na terenie Polski, stajemy się zakładnikami Polaków mieszkających w Niemczech.

A wiecie, że jest trudna sytuacja, pan szczególnie wie o tym, jak jest w samorządach. Dlatego też chciałbym tutaj i do pana, i do pana ministra Murdzka zaapelować o to, aby ta poprawka została zaopiniowana negatywnie.

O to proszę i za to dziękuję. Chciałbym także, wykorzystując jeszcze te parę minut, podziękować przedstawicielom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo, myślę, to jest jedyny ośrodek, który rozumie sprawy mniejszości narodowych i etnicznych i dba o to, aby jednak zadania, które są nałożone w ustawach (Dzwonek), były przez państwo polskie jak najlepiej realizowane. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Andrzeja Kosztowniaka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Szanowni Państwo!

Słyszymy z ust opozycji na wszelkie możliwe sposoby odmieniane informacje dotyczące wzrostu długu Skarbu Państwa, wzrostu wydatków w różnych obszarach, co do których państwo uważacie, że nie są tymi właściwymi, choć my będziemy uważali, że wsparcie dla przedsiębiorców, wsparcie dla rodzin, wsparcie dla służby zdrowia i wsparcie w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy - myślę o polskim wojsku, polskich służbach - jest niezbędne, a nie tylko potrzebne. I tym bez wątpienia, szanowni państwo, będziemy się różnić.

Myślę, że 2022 r. bez wątpienia też taki będzie.

Daleko nam jeszcze, szanowni państwo, do progów ostrożnościowych.

Chodziło o zabranie pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych po to, żeby nie przekroczyć określonego długu, maksymalnego długu określonego w naszej konstytucji. Szanowni Państwo! Jeżeli mówimy o długu Skarbu Państwa, on jest cały czas pod kontrolą i jest tym długiem, który jest jednym z niższych, ewentualnie środkowych stanów w Unii Europejskiej. Pokazujecie te wasze tablice: PiS równa się drożyzna. Jeżeli byśmy popatrzyli na drożyznę i na inflację w Europie, na świecie, to trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, że świat to drożyzna, a nie jedna czy druga partia polityczna, która jest przedstawicielem w naszym parlamencie.

To są, szanowni państwo, państwa, które od kilkudziesięciu lat nie notowały tak wysokiego poziomu inflacji. Pragnę powiedzieć, że w tych państwach, które wskazałem, w większości rządzą koalicje socjaldemokratyczne i lewicowe. I mówienie o tym, że my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadziliśmy państwo polskie i polską gospodarkę na jakiś grunt inflacyjny, jest nieprawdziwe.

To wszystko powoduje, szanowni państwo, że wystąpiły pewne przyczyny, które budują poziom inflacji nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. To przede wszystkim największy szok cenowy od lat 90. wynikający z nośników energii, przede wszystkim ropy naftowej, gazu, a w przypadku Europy i w przypadku państwa polskiego gaz będzie miał wielkie znaczenie. Niestety część przedstawicieli polskiej sceny politycznej, reprezentując nasze interesy na poziomie Unii Europejskiej, często o tym zapomina. Inflację trzeba czytać, proszę państwa, z kilkoma współczynnikami i czynnikami ekonomicznymi. PKB w Unii Europejskiej na poziomie 2%, my - ponad 5%. To jest coś, co nas cieszy i daje nam wielką nadzieję, pokazuje nam, że ta gospodarka polska jest prowadzona w sposób właściwy. Zbliżamy się do naturalnej stopy bezrobocia, która nigdy, przepraszam, przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Polsce nie była naszym udziałem. To wszystko pokazuje, szanowni państwo, jedną rzecz: polskie finanse publiczne nie są może w znakomitej formie, tak jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, również my ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale są zdecydowanie w lepszej sytuacji i kondycji niż finanse publiczne wielu państw Unii Europejskiej czy też wielu państw na świecie.

Proszę państwa, to dobry budżet. Gorąco państwa prosimy, abyście te wszystkie uwagi, które kierujecie, rozważyli. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Cichonia, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Białe jest białe, a czarne - czarne. To PiS jest odpowiedzialny za drożyznę w Polsce i nikt Polakom i Polkom nie wmówi, że jest inaczej. PiS to drożyzna, a drożyzna to wy właśnie. Inflacja jest jak przysłowiowa koza, mówiłem o tym w komisji finansów i na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Jeszcze wczoraj premier i minister finansów zacierali ręce, bo dzięki niej rosły wpływy budżetowe. Można było nowelizować kolejne budżety, opowiadając, że rząd zabiera mafiom, że skutecznie uszczelnia system podatkowy. Ale to nieprawda, ten wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z rosnących cen produktów i usług. To polskie gospodarstwa domowe z roku na rok, z miesiąca na miesiąc muszą wydawać coraz więcej, żeby normalnie żyć. Dochody z VAT rosną, ale co mają z tego polskie rodziny? Miały mieć pieniądze na godne życie, dzisiaj mają ledwo na przeżycie. Ale to nie wszystko, bo inflacja podbija nominalne PKB. Dzięki inflacji produkt krajowy brutto jest coraz wyższy, imponujący w tym nominalnym wymiarze, a dzięki temu spada też relatywnie zadłużenie. Inflacja pozwala wam na zadłużanie państwa na nienotowaną dotąd skalę zupełnie bez kontroli. Rozdajecie pieniądze dla swoich w formule, którą wielokrotnie już przytaczałem: komu na, komu nie. To w gruncie rzeczy komuna w czystej postaci. Opieracie wzrost gospodarczy na konsumpcji finansowanej długiem, spada stopa inwestycji, spada stopa oszczędności. Do tego wygląda na to, że ten rok to będzie pierwszy rok, w którym spadają oszczędności gospodarstw domowych. To jest karmienie tej kozy i tworzenie jej znakomitych warunków. A historia tej choroby to jest listek za listeczkiem, ponad 40 nowych podatków i opłat oraz podwyższanie istniejących. Za każdym razem mówiliśmy, że to jest napędzanie inflacji, że to kolejne impulsy inflacyjne, bo rosnące koszty podatkowe w działalności gospodarczej przerzucane są na klientów i ceny produktów i usług, i ceny produktów i usług rosną. Ile warte jest jeszcze słowo prezesa, który mówił, że nie będziecie podnosić podatków? Tu też mamy do czynienia z inflacją. Nic nie jadłam, nic nie piłam” A wy dalej tę kozę karmicie.

A do tego dochodzi jeszcze gospodarowanie majątkiem. Wielokrotnie o tym mówiłem, przytaczałem: Turów, Nowe Jaworzno, Bełchatów, Ostrołęka.

Parę lat temu ropa na rynkach światowych kosztowała 128 dolarów za baryłkę, dzisiaj - 75. Cen na stacjach nie będę przytaczał, bo każdy je widzi i klnie na czym świat stoi - drożyzna+, to ten PiS, tak mówią ludzie płacąc rachunki. To zapytam, kto w państwie polskim, kto w państwie PiS tak naprawdę odpowiada za siłę polskiej złotówki. Mam przypominać skrajnie nieodpowiedzialne interwencje na rynku walutowym, po to by przynieść rządowi parę miliardów w prezencie? To całkowicie niezależny - ale chyba od zdrowego rozsądku - prezes Narodowego Banku Polskiego. Nakręcacie spiralę inflacyjną. Tarcza inflacyjna, która ma, jak mówi premier, częściowo złagodzić skutki, będzie tę inflację tylko nakręcać, a potrzebna jest eliminacja przyczyn. Mówiłem to wielokrotnie: przestańcie doić państwo i obywateli, wstrzymajcie Nowy Ład w części dotyczącej przedsiębiorców, zmieńcie prezesa NBP, tak na dobry początek, i przedstawcie nowy budżet oparty na realnych założeniach, bo ten jest w gruncie rzeczy nie do zaakceptowania.

Dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze pan poseł Zdzisław Sipiera, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku miałem rozpocząć od swojej części, o której miałem mówić, ale dwa słowa odniesienia do mojego przedmówcy. Proszę państwa, wydaje mi się, że to jest dziwna sytuacja, że były minister mówi takie słowa: że czysta komuna w czystym wydaniu, że nikt nie czuwa nad długiem, skończcie rozdawnictwo pieniędzy, może powrót pana Balcerowicza, może pana Rostowskiego. Panie ministrze, dopóki nie macie władzy, starajcie się jednak nie przeszkadzać, lecz posłuchać, jaką mamy propozycję dla naszych obywateli. Przede wszystkim w tej dziedzinie, która jest istotna, dotyczącej bezpieczeństwa, co obywatele zawsze uważają za bardzo ważne, ale nie zawsze to było w przeszłości użytkowane w praktyce.

Dlatego, że to jest to, czego obywatele bezpośrednio oczekują.

To jest sfera ogromnych zagrożeń.

Podtrzymujemy to i wydajemy te środki finansowe. Przypomnę, jakie są cele wydatkowania tych pieniędzy: modernizacja techniczna Wojska Polskiego, wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostek operacyjnych dyslokowanych na wschodzie kraju - chyba nie muszę wszystkim tłumaczyć, dlaczego ma to być w tej części Polski - zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP, tworzenie warunków dla zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, formowanie struktur oraz budowa zdolności operacyjnych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, formowanie struktur i budowa zdolności operacyjnych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, realizacja procesu szkolenia Sił Zbrojnych, w szczególności w ramach krajowych i międzynarodowych ćwiczeń i treningów, zwiększenie zdolności wojskowej służby zdrowia do przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń epidemiologicznych.

Moi przedmówcy z klubu Prawa i Sprawiedliwości o tym mówili. Mówicie o rozdawnictwie pieniędzy, pan poseł mówił o rozdawnictwie pieniędzy. 77 wniosków zmniejszających wydatki Instytutu Pamięci Narodowej, 74 wnioski zmniejszające wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 21 wniosków zmniejszających wydatki Kancelarii Prezydenta i 16 wniosków zmniejszających wydatki na obronę narodową. Dlatego że to wszystko ma jeden cel. Mówicie państwo o drożyźnie, mówicie państwo o tym, że PiS to drożyzna.

Polacy chcą i oczekują realizacji zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zabezpieczenie granic państwa.

O tym nie mówiłem, ale jest cały komplet zagadnień związanych z KPRM.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu panią poseł Krystynę Skowrońską, Koalicja Obywatelska.

To PiS każdemu obywatelowi wyciąga każdego dnia z kieszeni pieniądze. Nie macie swoich pieniędzy. Rząd nie daje. Jak daje? Byle jak.

Zapowiadany był szumnie przez prezydenta Dudę.

A czekają np. dzieciaki chore na choroby rzadkie, mukowiscydozę. Mówię hasłowo, dlatego że czasu mamy mało.

A każdego roku przez ostatnie 6 lat - po 2 mld zł na telewizję Kurskiego. Czy wam nie wstyd? Przez ostatnie 6 lat drożyzna PiS. Zwiększają się długi szpitali. I manipulacja, czysta manipulacja na Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wynikiem tego są długi szpitali, kolejki do lekarza, bo one się nie zmniejszyły, i tragedie, które mogą czekać szpitale w przyszłości. Drogi prąd, drogie nośniki - zero osłony. Mówicie o dobrym budżecie? Jakby było tak dobrze w ochronie zdrowia i wszędzie, to nie strajkowaliby pielęgniarki, ratownicy medyczni, nie umierałoby tyle osób. Na państwa sumieniu ciąży 80 tys. zgonów COVID-owych - nie poradziliście sobie w ochronie zdrowia - i 140 tys. zgonów ponadwymiarowych. To brak działania. I nie mówcie, że ważniejsza jest obrona narodowa. Najważniejsze dla każdego Polaka, dla nas wszystkich jest życie Polaków i ratowanie. Wyciągacie każdego dnia z naszych kieszeni pieniądze. PiS - to drożyzna, PiS - to nadmiarowe zgony, PiS - to długi szpitali, PiS - to strajki pracowników ochrony zdrowia, PiS - to niewykorzystany Fundusz Medyczny. To wasze sumienie. Za to kiedyś odpowiecie. Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość.

Dziękuję, panie marszałku. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje politykę wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i jednocześnie wdraża jej reformę. Budżet ochrony zdrowia na rok 2022 jest kolejnym potwierdzeniem tego, że potrafimy dotrzymywać obietnic i realizować ambitne projekty.

Ustawowe gwarancje 7% PKB i konsekwentna ich realizacja rok po roku przez rząd PiS oznaczają, że do średniej krajów Unii Europejskiej dojdziemy już w 2027 r. W świetle powyższych liczb w osłupienie wprawia demagogia lub brak wiedzy - a pewnie jedno i drugie - byłego premiera, który przybył z Brukseli, podobno naprawiać Polskę, a który 24 listopada zarzucał rządowi, że, cytuję: dzisiaj Polska - co ludziom się chyba w głowie nie mieści - jest jedynym krajem w Europie, który w czasie pandemii obniżył ilość środków na ochronę zdrowia. Od 2009 r., gdy był premierem, wydatki na ochronę zdrowia w relacji do PKB zaczęły spadać, by w 2014 r. osiągnąć najniższy poziom 4,57% PKB. W 2015 r. nakłady według planu wynosiły 74 mld zł, to był ostatni rok waszych rządów.

Jak wspomniałam, są to jeszcze dodatkowe środki, które trafiają również na potrzeby w zakresie ochrony zdrowia.

I oczywiście dodajecie, że jest to wina PiS. Tusk nie chce pamiętać, państwo również, że kiedy rządziliście i kiedy nie było pandemii, nie było ochrony gospodarki, ochrony firm, które otrzymały ok. 200 mld zł w ramach pomocy, nie było wzrostu cen surowców energetycznych.

Wysoka Izbo, co wtedy państwo robiliście, jakie były wasze działania związane z przeciwdziałaniem inflacji? Przerzucaliście wszystkie ciężary na najuboższych, na społeczeństwo. Ano co robiliście? Co pani poseł robiła? Za czym pani poseł głosowała? powodując zadłużenie osób, które zaciągnęły kredyty, i bankructwa wielu kredytobiorców.

Sami koledzy klubowi przeszkadzają pani poseł w wystąpieniu.

To była wasza tarcza antyinflacyjna i to jest ta alternatywa, jaką macie dla Polski wobec polityki obecnego rządu Zjednoczonej Prawicy. Mówiłam o ogólnych wydatkach. 133 mld, czyli blisko 80% więcej, niż wy dawaliście na ochronę zdrowia.

No, jeśli jest to mniej, niż było przedtem, to jest to albo amnezja, albo próba nie naprawy państwa, tylko robienia zadymy, chaosu, po prostu żerowania na niskich uczuciach Polaków.

Podpuszczacie ratowników medycznych. Zwiększyliśmy o 24% środki na ratownictwo medyczne, o prawie 600 mln zł, do poziomu 2800 mln zł, na zwiększenie stawki za dobokaretkę oraz dodatki wyjazdowe. Gdzie to było za waszych czasów?

Sprzedawaliście w obce ręce, bo Niemcy potrafią lepiej robić badania diagnostyczne w polskich laboratoriach, w polskich szpitalach niż polscy diagności. Taka była wasza polityka. 4 mld zł na Fundusz Medyczny. Była tu mowa o Funduszu Medycznym. Pani poseł, dokładnie pan minister wyjaśniał kwestię Funduszu Medycznego zarówno w Komisji Zdrowia, jak i w komisji finansów. To są duże pieniądze, do dyspozycji m.in. na pediatrię. Choroba COVID spowodowała, że zapotrzebowanie na ten cel ze strony szpitali psychiatrycznych nie było tak duże, jak oczekiwaliśmy. I te pieniądze nie przepadają, one są. A to są duże pieniądze i trzeba dokładnie przygotować procedury ich wykorzystania. Jak widzimy, nie wierzą wam. Mamy także oczywiście dodatkowe środki na psychiatrię, która jest wielkim problemem w Polsce.

Proszę państwa, to wszystko, co będzie w roku 2022, będzie stanowiło kontynuację zadań i podejmowanie nowych zadań, bo od wielu lat walczymy z zaniedbaniami naszych oponentów, naszych przeciwników politycznych. Co zrobiliśmy? Co zrobiliśmy?

Tu mnie koledzy oczywiście mobilizują, że trzeba kończyć. Proszę państwa, myślę, że z czystym sumieniem można głosować za projektem budżetu na 2022 r. dla dobra Polaków, ponieważ dla nas stawką jest życie i zdrowie Polaków. Będziemy konsekwentnie to realizować. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Moja przedmówczyni nie zauważyła faktu, że od ponad 6 lat w Polsce niepodzielnie rządzi PiS, że inflację mamy największą od 20 lat i że PiS równa się drożyzna. System ochrony zdrowia jest nadwyrężony pandemią, tak samo jak przemęczeni walką o zdrowie i życie Polaków są medycy i pracownicy niemedyczni. To oni od wielu miesięcy walczą na pierwszej linii frontu walki z pandemią, która przez bezczynność i nieodpowiedzialność rządu zbiera tragiczne żniwo, jeśli chodzi o zgony i wykryte zakażenia. Rząd zapewnia, że w przyszłym roku nakłady na zdrowie będą wyższe. Nie wiem, skąd ten optymizm, bo w żadnej mierze nie jest to realny wzrost. Zdrowie zawsze powinno być najważniejsze, a w czasie pandemii potraktowane w sposób szczególny, nie tylko poprzez niewielkie zwiększenie środków, bo tych jest zdecydowanie za mało. Tę nadwyżkę przecież zje inflacja, a potem pożre ona jeszcze więcej.

Pandemia i niezdiagnozowani, zaniedbani pacjenci z chorobami onkologicznymi, kardiologicznymi, diabetologicznymi, z chorobami przewlekłymi zaciągają olbrzymi dług zdrowotny. Kiedy brakuje pieniędzy na świadczenia medyczne, kiedy publiczna służba zdrowia ciągle się zadłuża, a powiatowe szpitale stoją na skraju finansowego bankructwa, co robi rząd? Rząd uruchamia Fundusz Medyczny, fundusz, który ma funkcjonować w ramach tych samych środków z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, słysząc kilka dni temu takie wystąpienie, kolejną propagandę premiera Morawieckiego, który powiedział: Fundusz Medyczny to specjalnie skonstruowany wehikuł medyczno-finansowy, który ma zasilać cały system zdrowia, w jego najbardziej newralgicznych miejscach, w finansowanie. Jedynie 171 mln. No tak, ale wszyscy pamiętamy, że Fundusz Medyczny miał inne podłoże niż troska władzy o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Ciągle o nim słyszymy, nikt go nie widział, taki pic na wodę, fotomontaż. Ale kiedy się o nim opowiada, jest sprawdzonym lekiem na spadające słupki PiS-u. Tak nie uzdrowicie systemu ochrony zdrowia, dlatego żądamy realnego finansowego zastrzyku dla zdrowia.

Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoki Sejmie! Cóż, bardzo mało czasu, a chciałoby się tyle powiedzieć. Cała moja koncepcja wystąpienia została zdemolowana przez szanownych kolegów i koleżanki z Platformy, którzy wystąpili z tak prostym, chciałoby się powiedzieć: populistycznym, prymitywnym chwytem, z tym właśnie napisem. To jest problem demokracji.

To prawda. Ale partia, główna partia opozycyjna, która mieni się, aspiruje do wzięcia odpowiedzialności za ciężar rządów w kraju, powinna prezentować wyższy poziom i nie wciskać tego aż tak mocno, bo obrażacie inteligencję swoich wyborców, jak również innych myślących. Każdy Polak jest już na tyle wyedukowany, że dobrze to wie. Mamy swoją odpowiedzialność, ale przede wszystkim obiektywne, zewnętrzne, niezależne czynniki są główną tego przyczyną, w tym polityka klimatyczna. Nie mogę rozwinąć skrzydeł, skrótowo tylko mówię, [[Oklaski]] teraz 5 minut, a 3 minuty dla przewodniczącego. Proszę państwa, więc jeżeli tak - trudny wybór, kusa rada. Trzeba dokonać wyboru, za kilka miesięcy albo za 2 lata. Jeżeli PiS to drożyzna, to oddalę się trochę i powiem: a co to jest Platforma? A o Platformie mogę powiedzieć tak na gorąco, że gdybym dzisiaj rano te plakaty robił, to Platforma równa się dobrobyt, oczywiście ironicznie. Albo też ja bym osobiście powiedział: pogoda dla bogaczy. To lepiej. Ale można by też powiedzieć, z czym się kojarzy Platforma. Panie marszałku, króciutko ich. Przepraszam. To nieważne. Jeszcze mam ponad minutę. A więc Platforma to godziwa płaca minimalna, 5 zł za godzinę. Platforma to godziwa emerytura, przyjrzyjmy się, jak to było. Platforma - wakacje dla każdej rodziny. To najpiękniejszy symbol naszych rządów. To wam teraz odpowiem. Pomoc dla niepełnosprawnych, ta sprawa w Sejmie. A fakty, konkrety? 2015 r., sprawdźcie to, ci, którzy nas słuchają. 15 mld łącznie.

Obiecano? Obiecano. A więc słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Musimy to zrobić, naprawić ten błąd, przy 30 tys. kwoty wolnej. Kwota wolna od podatku, nie będę się już na was tutaj. I mieszkanie, gniazdo, to ciepło rodzinne. Idzie Wigilia. Tym, którzy wyjechali za granicę? Kończąc i przekazując pałeczkę przewodniczącemu, powiem tylko jeszcze jedną rzecz. To jest program pożyczkowy, bądźmy uczciwi i oddajmy sprawiedliwość. Skąd brać pieniądze? I Marek Balicki jak przysłowiowy prawdziwy lewicowiec powiedział: Podnieść podatki dla najbogatszych. To nic nie daje, bo w ministerstwie to analizowaliśmy, to tylko miliard. Jaka była odpowiedź? Pani redaktor, musimy każdą złotówkę oglądać, ale nie w tych kieszeniach, gdzie jest dużo pieniędzy, tylko w tych, gdzie jest ich mało.

Panie Marszałku! Drogo, drożej, ciemno - taką transformację energetyczną proponuje rząd PiS. Spółki Skarbu Państwa, zamiast inwestować w OZE, topią pieniądze w Ostrołękach, w kupowaniu gazet, a rosnące koszty przerzucają na odbiorców energii, powodując szalejącą drożyznę. Z drogich uprawnień tak naprawdę rząd się cieszy, bo z ich sprzedaży, tych bezpłatnych, które otrzymał, tylko w tym roku do budżetu wpłynie niemal 30 mld, prawie trzy razy więcej, niż zaplanował i... ślad po nich ginie w tym budżecie. 10 mld na swoisty fundusz odporności polskich rodzin na wasze wzrosty cen energii i zdrowe ciepło, czyli na bezpieczeństwo dostaw energii dla polskich rodzin i uniezależnienie się od drożyzny w postaci własnych źródeł energii odnawialnej, magazynów energii; na efektywność energetyczną, by oszczędzić zużycie, unikając strat energii w domach.

Przypomnę, że proponujemy także 1 mld na ekologiczne ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych. One są także źródłem smogu, mieszka tam najwięcej niezamożnych rodaków, tymczasem rząd bezpośrednio wspiera tylko właścicieli domów jednorodzinnych. Dziękuję bardzo. Pozostały czas przeznaczony dla klubu wykorzysta pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niestety mimo płomiennych apeli państwa posłów z Prawa i Sprawiedliwości będziemy głosować za odrzuceniem projektu budżetu. Z trzech powodów. Przecież wszyscy wiemy, że będzie wyższa. A może to nie jest błąd, może to celowa działalność. Po drugie, przyjęliście stopę procentową na poziomie 1%.

To jest pierwszy powód. Trzeba to przerobić.

To było 10%. W przyszłym roku ma to być 40%. 40% pieniędzy publicznych wydawanych przez rząd przechodzi poza kontrolą parlamentu. Nie wiem, jak państwo posłowie się do tego odnoszą.

Nie spełniacie w ogóle swojej konstytucyjnej funkcji. 40% - wiecie, ile to oznacza?

Budżet jest tak skonstruowany, że praktycznie nie ma w nim pieniędzy na rozwój ważnych obszarów usług publicznych i społecznych. Była mowa o zdrowiu.

Bo w ogóle nie wierzę w to, co państwo przedstawiacie, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia. Eurostat daje rzetelne statystyki. Nie ma wzrostu, a mamy pandemię. Mimo że mamy pandemię, to udział wydatków na zdrowie w Polsce nie rośnie. To jest pierwsza sprawa. Chcę państwu powiedzieć, jak to wygląda na tle Unii Europejskiej, bo warto się przyjrzeć. Jeśli chodzi o tak ważne obszary usług społecznych jak zdrowie, jesteśmy na 23. miejscu na 27 państw.

Ale są rankingi, w których jesteśmy wyżej. Wydatki na Policję - na 6. miejscu.

Nie mówimy o Białorusi, nie mówimy o tym roku, tylko mówimy o poprzednich latach. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której są pewne priorytety realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie wiem, czy one są akurat najważniejsze w oczach wszystkich Polaków. Mamy drożyznę, o której mówimy. Mamy kryzys zdrowotny, którego nie jesteście w stanie przełamać. Mamy kryzys ze szczepieniami, nie posuwacie się ani na krok w realizacji najbardziej skutecznej metody walki z kryzysem pandemicznym. W tej sprawie nie robicie nic. Mamy zapaść w inwestycjach, jesteśmy na 3. miejscu od końca, jeśli chodzi o poziom inwestycji prywatnych.

Szanowni Państwo! Bez inwestycji nie ma rozwoju, nie będzie rozwoju. My wszyscy jedziemy na ostatnich oparach paliwa, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. To jest cały czas wzrost finansowany dosypywaniem pieniędzy do konsumpcji. Przecież nie ma się co dziwić, że mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie, właśnie dlatego, że tyle pieniędzy trafia na rynek, a nie trafiają one na inwestycje, na rozwój zdolności wytwórczych, tak żeby w ślad za pieniądzem popytowym była także jakaś podaż.

To już chyba mamy załatwione, że w tym roku nie zobaczymy ani jednego euro. Macie jeszcze szansę, żeby się dogadać z Unią Europejską, ale jeżeli się nie dogadacie, naprawdę nie będziemy mieli pieniędzy na inwestycje.

To jest inflacja, ale to także jest rozwój gospodarczy. Ale my chcemy więcej. Polacy oczekują od was, żebyście rozwiązywali problemy. Chodzi o brak inwestycji, zapaść demograficzną, brak rąk do pracy, kryzys zdrowotny, kryzys, jeśli chodzi o edukację, transformację energetyczną, wszystko jest zawalone. Więc jak my mamy poprzeć ten budżet?

Proszę bardzo. Zacznę może od tego, że do tego dobrego budżetu - bo nie podzielam opinii mojego przedmówcy, jakkolwiek doceniam przygotowanie i merytoryczną wypowiedź, jedną z nielicznych, może jedyną - jeszcze garść poprawek, kilkanaście poprawek klubu Prawo i Sprawiedliwość, który popiera z całą mocą ten dobrze przygotowany dokument. Szanowni Państwo!

Proszę państwa, przecież my tych pieniędzy nie konsumujemy, tylko instytucje administracji państwowej, samorządy, poszczególni dysponenci. Proszę państwa, dysponenci budżetowi w czasach kryzysu czekają na pieniądze. Właśnie to, co cechuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest błyskawiczne dysponowanie pieniędzmi.

Nie chciałbym wracać do tego, jakie państwo mieliście pomysły, ale przypomnijmy sobie wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, jak inflacja urosła za waszych czasów do 5%. Proszę państwa, zaproponował wejście do strefy euro, co w naturalny sposób u naszych sąsiadów południowych zwiększyło ceny.

Podniesienie wieku emerytalnego - dla pań na wsi o 12 lat, dla pań w ogóle o 7 lat, dla panów plus 2% do 67. roku życia. Przez to straciliście władzę. Musicie jeszcze dosyć długo siedzieć i grzać ławy opozycji, żeby Polacy wam to wszystko zapomnieli. Wiem, że na to liczycie.

Proszę państwa, kwestia zielonego ładu.

Proszę państwa, pytanie jest inne: Czy Unię stać na wdrażanie dzisiaj polityki zielonego ładu w sytuacji, kiedy mocarstwa takie jak Chiny, Stany Zjednoczone, Bliski Wschód, Indochiny w ogóle z tego się wycofują, ewentualnie potakują? Po to, żeby zlikwidować konkurencyjność gospodarki europejskiej.

Potrafię to sobie wyobrazić, ale że Unia sama jako całość dzisiaj nie bierze tego pod uwagę, to budzi to moje lekkie zastanowienie. Szanowni państwo, zostało mi, jeśli dobrze liczę, jakieś 45 minut. Czy pan to zauważył? Proszę państwa, po raz kolejny podjęto próbę odpersonalizowania, zanonimizowania rzeczywistych osiągnięć rządów Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, chcę tylko jedną rzecz powiedzieć: strach i odwaga w tych wypowiedziach, które tutaj miały miejsce, mieszały się. Odwaga była po naszej stronie. My przyjęliśmy, chcemy przyjąć w tej Izbie dobry dokument. Proszę państwa, państwo epatowaliście obywateli strachem, a my mamy wielkie marzenia i nie paraliżujemy ich strachem. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy. Występuję dzisiaj w podwójnej roli. Mam zaszczyt być też sprawozdawcą sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Chciałem podziękować wszystkim klubom za to, że te poprawki. Nie zapominam o wnioskach mniejszości, których jest sporo. Dzisiaj mają już taki charakter dopinający, wyważony. Byłem bardzo mocno pocieszony deklaracją jednego z klubów, klubu Lewica, że zechciałby poprzeć budżet.

Z wnikliwą uwagą będę też jako przewodniczący komisji finansów próbował na ten temat rozmawiać. Chcę powiedzieć, że samo zadłużanie szpitali następowało przez lata. Przypomnę tylko, że to przecież nasz rząd podniósł właściwie o 100% wynagrodzenia lekarzy, którzy pracują w kontakcie z pacjentami COVID-owymi, żeby nie brakowało w jakimś ekstremalnym stopniu obsługi merytorycznej osób, które dzisiaj wymagają leczenia i wymagają opieki.

Mili Państwo! Jako przewodniczący od razu też proszę obecnych tutaj posłów uczestniczących w pracach naszej komisji o to, żeby jednak byli osobiście - nie będzie zwolnienia, jeśli chodzi o pracę zdalną, bez względu na słuszną decyzję pani marszałek - z uwagi na to, że chciałbym, żebyśmy przygotowali dobre sprawozdanie do trzeciego czytania.

Dziękuję bardzo.

Szanowni państwo. Ale proszę, panie pośle, nie robić takich uwag, bo mam wrażenie, że akurat nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wystąpienia i o pytania.

Jeżeli nie, to zamykam ją, ustalając czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Aleksander Mrówczyński. A zatem prosimy panią poseł Krystynę Skowrońską.

Drożyzna równa się PiS. Wasza wina, wasza wina, wasza wielka wina. Czy przez 6 lat ten rząd obniżył VAT? Nie. Każdego miesiąca każdego roku 8 mld z naszych kieszeni. Szukajcie porządnych argumentów. Budżet. Mówicie państwo o transformacji, o wyciąganiu pieniędzy z kieszeni. Jak wyciągniecie, to jak złodzieje nie oddacie.

W okresie kryzysu szpitale nie dostały pomocy. Nadmiarowe zgony, dłuższe kolejki i ludzie umierają przed szpitalami. Wasza wina, wasza wina, wasza bardzo wielka wina. Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Rafała Adamczyka. Wysoka Izbo!

Gospodarka wodno-ściekowa w Dąbrowie Górniczej. Budowa letniego basenu w Będzinie. Remont zamku w Będzinie i w Siewierzu i wiele, wiele innych. To jest kilkadziesiąt poprawek, które są złożone, podpisane. Pytanie otwarte: Czy posłanki i posłowie Wysokiego Sejmu poprą te poprawki? O lewą stronę jestem spokojny. Pytanie jest skierowane przede wszystkim do prawej strony. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Czesława Siekierskiego, Koalicja Polska.

Mówimy o raju wydatkowym, który jest nie tylko w rezerwach budżetowych, ale także w BGK, Polskim Funduszu Rozwoju, funduszu COVID-owym. To wszystko jest do dyspozycji premiera i rządu, poza kontrolą Sejmu.

Jakie przewidujecie wsparcie dla rolników w tej sytuacji, w której się znajdujemy? Wreszcie jeśli chodzi o poziom zadłużenia: Jaki jest rzeczywisty poziom zadłużenia państwa w ujęciu centralnym, rządowym, ale także w ujęciu samorządowym? Ile środków uzyskaliśmy ze sprzedaży uprawnień do emisji? Wreszcie: Jak szacujecie wielkość podatku inflacyjnego, który jednak wpłynął do budżetu, zapłacili go konsumenci? Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż różnica między prawicą a lewicą polega na tym, że lewica chce możliwie dużo dawać, żeby budżet był duży, żeby z niego można było dać. A prawica chce mieć budżet mały, żeby nie zabierać jednym i dawać drugim, tylko żeby ludzie te pieniądze po prostu mieli w kieszeni. Bo, po pierwsze, oni lepiej wiedzą, na co wydać, niż rząd. Nawet gdyby rząd nie kradł, nawet gdyby rząd chciał jak najlepiej, to i tak nie wie tego co ja. Po drugie, tworzy się warstwa ludzi, którzy tracą czas na pisanie podań o różne ulgi itd. To jest duża, ciężka praca. Ale, po czwarte, robi się ogromna kategoria ludzi, którzy żyją z tych dotacji kosztem innych. To, co wy robicie (Dzwonek), to nie jest polityka prawicowa, tylko lewicowa. Tylko to nie jest polityka prawicowa. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Michał Gramatyka. Wysoka Izbo! Miał być program dla Śląska. Miała być inteligentna kopalnia. Miały być gigantyczne farmy fotowoltaiczne w okolicach Jaworzna. Miało być Beskidzkie Centrum Narciarstwa za 500 mln zł. Miał być kompleks produkcji wodoru. Miał być poligon dla dronów na terenach Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński. Temat dronów najlepiej podsumował wasz minister, pan minister Dworczyk w tych mejlach, które niby nie są jego, nie są wasze i do których się nie przyznajecie. A temat waszego epokowego programu dla Śląska najlepiej podsumowała górnicza „Solidarność”, ojciec i matka chrzestni w jednej osobie, bo wycofała swoich przedstawicieli z rady wykonawczej programu. A szef tej „Solidarności” powiedział: nie rób pan propagandy - do pana premiera. Albo ten program realizuj, albo po męsku odpuść. Czy zatem zamierzacie realizować, czy po męsku odpuścicie? Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Ryszard Galla. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie chciałbym skierować do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki. W uzasadnieniu poprawki, o której mówiłem w swoim wystąpieniu, czyli dotyczącej obniżenia subwencji ogólnej w części oświatowej, wnioskodawca dokonał takiego zapisu.

Chciałbym zapytać pana przedstawiciela, pana ministra, jak to ma być zrealizowane. W jaki sposób państwo chcecie skonsumować tę poprawkę? Bo przecież mamy jeszcze klasy dwujęzyczne, z rozszerzonym językiem, mamy także inne przedmioty w języku niemieckim jako ojczystym. Jak państwo chcecie to fizycznie zrealizować? Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Janusz Kowalski jest na sali? Nie widzę. Pani poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej też nie ma. Zatem pan poseł Jan Szopiński, który na pewno jest.

Tak, dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie Marszałku! Nie ma sprawnego działania Policji bez pracowników cywilnych Policji. To duża, prawie 25-tysięczna grupa profesjonalistów, informatyków, finansistów, techników, analityków i innych specjalistów, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie ani Komendy Głównej Policji, ani komend i jednostek Policji żadnego szczebla i żadnej specjalności. Otóż w 2022 r. 25% spośród tych pracowników zarabiać będzie najniższą krajową. Złożyliśmy poprawkę oznaczoną numerem 478, która daje tym pracownikom nadzieję. Daje nadzieję na wyższe uposażenie. Panie i panowie posłowie, ta poprawka daje tym pracownikom nadzieję. Głosujcie za poprawką nr 478. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nasz klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił szereg poprawek obejmujących ważne obszary funkcjonowania naszego państwa. Wśród nich jest także obszar dotyczący infrastruktury. Ja konsekwentnie dopominam się o inwestycje z województwa łódzkiego, inwestycje drogowe, o które zabiegałem jako ludowiec, ale one były także potwierdzane przez państwa parlamentarzystów, a do dzisiaj niestety nie zostały zrealizowane. Dlatego pytam, czy w następnym budżecie znajdą się w końcu pieniądze na obwodnicę Radomska, na obwodnicę Skierniewic, na obwodnicę Tomaszowa Mazowieckiego, a także długo wyczekiwany remont drogi od Spały przez Inowłódz do miejscowości Poświętne i dalej, do końca województwa, drogi krajowej nr 48, na której zdarza się bardzo wiele tragicznych wypadków. To inwestycje od lat (Dzwonek) wyczekiwane przez mieszkańców województwa łódzkiego. Bardzo proszę, aby znalazły się pieniądze na tego rodzaju działania. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz, jeśli pan poseł pozwoli, panią poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską. Dziękuję bardzo, panie pośle. Najmocniej przepraszam - przyszłam prosto z komisji, naprawdę, a już szybciej nie umiałam. Panie i Panowie Posłowie! Przyszły rok nie rysuje się chyba oszałamiająco dla budżetu, a zwłaszcza dla Polaków, więc dobrze by było szukać jakichś oszczędności. Więc mam pytanie do prawej części sali: Czy poprzecie państwo naszą poprawkę, poprawkę Koalicji Obywatelskiej, która likwiduje kuriozalny zapis o przekazywaniu każdego roku 2 mld zł telewizji publicznej pana Jacka Kurskiego? Wydaje mi się, że pieniądze podatników nie powinny służyć kłamstwu, chamstwu i szczuciu (Dzwonek) Polaka na Polaka. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Debata budżetowa to zawsze jest debata na temat czczych obietnic i pobożnych życzeń partii rządzącej. Oczywiście rozmawiamy też tutaj o jakimś stopniu rozdawnictwa, więc idźmy w to i porozmawiajmy o tym, co rzeczywiście jest ważne. W styczniu tego roku wygłosiłem z mównicy sejmowej przemówienie w ramach oświadczeń poselskich na temat dzieci chorujących na SMA. Rozmawialiśmy wtedy o tym, jak gigantyczne koszty ponoszą rodzice tych dzieci i jak dramatyczna jest ich sytuacja: muszą zbierać pieniądze, żeby ich dziecko miało jakiekolwiek szanse na przeżycie i na życie w miarę normalny sposób.

Bardzo dziękuję panu posłowi. To przesuniemy. A teraz pan poseł Andrzej Kosztowniak. Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Jedno pytanie o inflację, w Polsce i w Europie: Ile państw w Unii Europejskiej od okresu rozpoczęcia COVID-19 zanotowało wzrost inflacji? Chciałbym porównać dwa okresy, które wydają się nieco podobne.

Słyszeliśmy Donalda Tuska, który mówił jasno, że gdyby miał ten guzik, toby bez przerwy wciskał, wciskał, a niektórzy mówią, że nawet zawijał później w papierki. Dziękuję bardzo. Czy można prosić o nieprowadzenie dyskusji z zadającym pytanie? Pan poseł Krzysztof Gadowski. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To, że dzisiaj uprawnienia kosztują 87 euro w stosunku do 2016 r., kiedy kosztowały 6 euro, to wasz problem. Wyście nic nie zrobili w zakresie zmiany, transformacji energetycznej. Zablokowaliście rozwój OZE, wiatraków na lądzie, blokujecie fotowoltaikę w zakresie własnego taniego prądu. Nic w tym zakresie nie robicie. Nie wybudowaliście sieci energetycznej do obsługi fotowoltaiki. Panie Ministrze! Obiecaliście, że do końca września powołacie Fundusz Transformacji Śląska - ustawą. Pytanie zasadnicze: Kiedy to zrobicie? Jakie środki finansowe na ten fundusz zabezpieczacie? Dziś nie doszacowaliście wpływów z emisji. Na co te pieniądze przeznaczacie? A przecież w tym roku to ponad 24 mld zł. A w przyszłym roku ile? Dziękuję bardzo.

To musi zabrzmieć głośno i wyraźnie. PiS w swoim budżecie zaplanował miliony na odprawy dla swoich zwalnianych notabli. Zaplanował też miliony na nie wiadomo co. Od miesięcy w zamrażarce leży moja ustawa o domach pomocy społecznej. Chodzi w niej o to, aby ludzie tam pracujący zarabiali choć odrobinę lepiej. Podczas pandemii widzieliśmy, jaka to ważna, odpowiedzialna praca. Ci ludzie ze swoimi podopiecznymi musieli tam podczas kwarantanny zamieszkać.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Mirosław Suchoń. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wśród poprawek, które zgłosiłem do budżetu, są niezwykle ważne związane z budową infrastruktury, m.in. budową Beskidzkiej Drogi Integracyjnej oraz skrzyżowań bezkolizyjnych w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach, z drogami wojewódzkimi m.in. w powiatach cieszyńskim, żywieckim i bielskim. Chciałem zapytać pana ministra, czy rząd poprze te poprawki, które wynikają z realnych potrzeb naszego regionu. Mówiąc wprost, jeżeli tych dróg nie będzie, jeżeli nie zostaną wyremontowane, to nie ma co liczyć na to, że w tym regionie nastąpi znaczące przyspieszenie gospodarcze, a przecież tego gospodarczego przyspieszenia potrzebujemy.

Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Sylwestra Tułajewa. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt budżetu państwa na rok 2022 to przede wszystkim bezpieczeństwo - bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tak skonstruowany projekt budżetu sprawia, że realizujemy nasze zobowiązania względem NATO. Przeznaczamy 57 800 mln zł na obronę narodową, realizujemy nasze zobowiązania względem NATO na poziomie 2,2% PKB. To bardzo ważne. Z drugiej strony mamy odpowiednie finansowanie Policji, przeznaczamy na nią blisko 11 mld zł, zwiększamy tę kwotę.

Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania panią marszałek Barbarę Dolniak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zjednoczona Prawica, idąc 6 lat temu do wyborów, mówiła o istotnych zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Dzisiaj, po 6 latach, nawet rządzący nie kwestionują tego, że jest źle. Proponujecie państwo wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych, kuratorów sądowych i pracowników prokuratury na poziomie, który nie pokryje nawet inflacji. Nie słuchacie państwo tych pracowników, którzy mówią, jak niskie wynagrodzenia obowiązują w sądach czy prokuraturze. Wyliczacie państwo jakieś średnie wynagrodzenia, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

czy pracowników prokuratury.

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Krzysztof Śmiszek. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W budżecie na 2022 r. zaplanowano pieniądze na wszystko - na fundusze, na instytuty, na synekury dla krewnych i znajomych królika. A na co nie zaplanowanych żadnych pieniędzy? Na podwyżki dla strajkujących od miesięcy pracowników administracyjnych sądów i prokuratur, dla osób, na których opiera się tak naprawdę nasz wymiar sprawiedliwości, dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi bardzo często niewidocznych, którzy tworzą, wraz z niezależnymi sędziami, polski wymiar sprawiedliwości. To są ludzie, dzięki którym nasze konstytucyjne prawo, prawo do sądu, jest realizowane nawet w tak ciężkich czasach, jak czasy Prawa i Sprawiedliwości, które rozmontowuje wymiar sprawiedliwości. To naprawdę niewiele w skali całego budżetu, ale bardzo wiele dla tych, dzięki którym Polacy mogą jeszcze liczyć na wymiar sprawiedliwości. Wzywam wszystkie siły polityczne, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, żeby poparły tę naszą poprawkę. Wymiar sprawiedliwości to nie tylko niezależni sędziowie, którym należy się szacunek i godność.

Pytanie zada pan poseł Wojciech Maksymowicz. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawiążę do wypowiedzi posła Wiesława Janczyka, którą w kontekście Funduszu Medycznego należałoby niestety odebrać jako żart. Cytuję: To, czym charakteryzuje się Prawo i Sprawiedliwość, to błyskawiczne dysponowanie pieniędzmi.

Czy nie ma potrzeb, czy raczej nie potrafią państwo tego rozdysponować? A może jest jeszcze gorzej, może postanowiono kumulować środki, bo potrzeby chorych na raka, umierające dzieci mogą poczekać? Czy to w ogóle jest możliwe? Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania pana posła Andrzeja Szlachtę. Wysoka Izbo! W 2018 r. minister infrastruktury zabezpieczył w budżecie na 2019 r. dodatkowe środki finansowe na szkolnictwo lotnicze studentów. Wynikało to z dynamicznego rozwoju rynku lotniczego.

Uczelnie oczekują, aby tę kwotę powiększyć o 10 mln zł. Dlatego zwracam się z pytaniem do pana ministra infrastruktury: Czy jest możliwość, aby w części 39: Transport dokonać takiego przesunięcia? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Tomasz Piotr Nowak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cóż widzimy w tym budżecie?

A co widzą?

Szanowni Państwo! Wyzwania, które stoją przed Polską, są wyzwaniami transformacyjnymi.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Dariusz Wieczorek. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Natomiast mam pytanie dotyczące tych słynnych funduszy. Prawda jest taka, że w tym budżecie, zresztą tak jak w poprzednich budżetach. Właściwie drugi budżet wydajemy w tych różnych funduszach i jednostkach zależnych. Jest taki Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Cena energii jest tak wysoka m.in. z tego względu, że odpisy z dywidend spółek Skarbu Państwa idą m.in. na ten Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Moje pytanie jest takie: Jakie są plany, jeżeli chodzi o zakup akcji spółek przez pana premiera i które spółki chcemy kupić? Czy to są kolejne spółki medialne, czy to jest koncern TVN? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Zbigniew Babalski. Wysoka Izbo! Mówicie: podnieście wyżej, będzie lepiej wyglądało. Panie Ministrze! Wracam do ustawy modernizacyjnej.

I na koniec pytanie retoryczne do opozycji, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć, a jest ono aktualne od dziesiątków lat. Co jest lepsze: niska inflacja (Dzwonek) i wyższe bezrobocie czy niższe bezrobocie i wyższa inflacja?

Bardzo dziękuję. Pytanie teraz zada pani poseł Ewa Kołodziej. Panie Premierze! Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłorocznym budżecie nie znalazła się poprawka Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy dotycząca grupy osób chorych na cukrzycę.

Szanowni Państwo! Cukrzyca nazywana jest pierwszą niezakaźną pandemią na świecie. To nie przypadek, dlatego że w Polsce zapadło na nią już 3 mln osób, natomiast 5 mln osób jest grupie ryzyka. Nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby uświadomić sobie, że 8 mln osób w Polsce choruje na tę chorobę bądź niebawem na nią zapadnie. W czasach pandemii, kiedy zmagamy się z koronawirusem, cukrzyca to pierwsza choroba współistniejąca, która predysponuje do ciężkiego przejścia COVID-19. W tym momencie nie pomagając cukrzykom, narażamy ich na utratę życia i zdrowia. Nie wyobrażam sobie, żeby ta poprawka nie uzyskała państwa akceptacji. Pytanie zada pan poseł Tomasz Trela. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Tych pieniędzy nie ma w tym roku i wszystko wskazuje na to, że nie będzie ich też w przyszłym roku. Dlatego złożyłem dwie poprawki.

Chciałbym zapytać pana ministra, czy samorządy, które nie dostaną pieniędzy w ramach funduszy europejskich ze względu na państwa nierozsądną, nieracjonalną politykę (Dzwonek) względem Unii Europejskiej, mogą liczyć na wsparcie pana ministra i większości Prawa i Sprawiedliwości? Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Pawła Rychlika. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Drodzy Polacy!

Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Nie ma. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Też nie widzę. Jest na sali pani poseł Maria Małgorzata Janyska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drogi Rządzie! Właściwie najdroższy rządzie, bo jest najdroższy od 2015 r., droższy o 664%. Mam wrażenie, że za marnotrawienie środków, za upychanie ich po funduszach na zewnątrz budżetu, żeby nikt was nie kontrolował, za upychanie długu na zewnątrz przez emisję papierów dłużnych, żeby nikt was nie kontrolował. Przez taką właśnie działalność Polacy za chwilę będą musieli iść na zakupy z torbami pieniędzy o wiele większymi niż torby z zakupami, które za te pieniądze zrobią. Gdzie jest KPO?

o obwodnice. Dlaczego? Dlatego że usłyszymy sakramentalne: chcielibyśmy. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Wiesław Buż. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Pandemia COVID-19 sprawiła, że transformacja cyfrowa ma ogromny wpływ na sektor publiczny i prywatny, a przede wszystkim na lokalne biznesy, w tym małą gastronomię i przewóz osób w systemie taksówek. Wielu przedsiębiorców zostało skazanych na łaskę globalnych gigantów cyfrowych i usługi wykonywane są za pomocą aplikacji. Światowi potentaci narzucają niekorzystne dla małych i średnich firm warunki współpracy.

Wskazują oni na fakt unikania ewidencjonowania transferu finansowego i unikania obowiązków podatkowych. Polska gospodarka powinna być odporna na działania cyfrowych gigantów.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Piotr Benedykt Zientarski. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy pan minister sprawiedliwości i jego najbliżsi współpracownicy rozumieją, jaki wpływ na funkcjonowanie sądów i prokuratur mają sekretariaty? Jako adwokat z ponadtrzydziestoletnim stażem przesiedziałem w sekretariatach tysiące godzin i byłem świadkiem tej ciężkiej, stresującej, odpowiedzialnej, wręcz benedyktyńskiej pracy.

Rotacja kadr jest zupełnie zrozumiała, ale wiąże się z odchodzeniem osób doświadczonych i przyuczaniem nowych. Fakt, że okres rozpoznawania spraw uległ za tego ministra sprawiedliwości przedłużeniu, często dwukrotnemu, wynika także z sytuacji płacowej pracowników sądów i prokuratur.

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Jerzy Hardie-Douglas. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jestem ze Szczecinka, miasta, które podobnie jak i jego okolice, jest uważane za jedno z miast, które są szczególnie wykluczone komunikacyjnie. Mamy bardzo daleko do najbliższych dróg szybkiego ruchu i wielką nadzieję od lat wiążemy z przebudową drogi ekspresowej S11. W tym roku ruszyła budowa na odcinku Koszalin - Bobolice. My w Szczecinku, a przypomnę, że jest to teren chyba najbardziej rozwinięty przemysłowo na Pomorzu Środkowym, czekamy cały czas na budowę odcinka Bobolice - Szczecinek.

Dlatego moja poprawka dotyczy zwiększenia finansowania tego odcinka drogi, który jest nam niezwykle potrzebny. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mówicie państwo często, że wysokie ceny energii to wina Donalda Tuska, ale gdy rządził Tusk, to pozwolenia na emisję były po 6 euro, a gdy rządzicie wy, są po 85. Mówię tak z pewną dozą złośliwości oczywiście, bo przecież sami sobie zdajecie sprawę, że to nie od tego zależy. Ale proponuję sprowadzić tę dyskusję do naprawdę merytorycznych argumentów. Chcę wam również powiedzieć, że 40% wydatków rządowych, które przechodzą poza parlamentem, poza tą Izbą i poza waszą kontrolą - wskazuję na panie posłanki i panów posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości - oznacza, że mamy do czynienia z brakiem kontroli nad olbrzymią częścią finansów publicznych. Krótko mówiąc, ponieważ wiemy, gdzie te pieniądze trafiają, one często trafiają właśnie do rozmaitych fundacji, chodzi np. o wspieranie (Dzwonek) Marszu Niepodległości, albo trafiają do o. Rydzyka. Chcę powiedzieć, że to jest naprawdę wielka pralnia pieniędzy i musicie z tym skończyć. Dwa sprostowania na koniec. Pani posłanka Masłowska mówiła, że w XX w. już mieliśmy wyższą inflację i podała jako przykład lipiec 2020 r. Chcę powiedzieć, że lipiec 2020 r. był w ubiegłym stuleciu, a nie w tym.

I ostatnie pytanie do pana ministra, jeśli jest. Chodzi mi o stawki FRA, które wyraźnie wskazują na oczekiwanie inflacyjne powyżej 3%. Proszę powiedzieć, jak Ministerstwo Finansów będzie finansować potrzeby pożyczkowe i jak to wpłynie na budżet? Bardzo proszę, pan poseł Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Widzę, że macie trzy zasady: łupić przedsiębiorców, zadłużać państwo i nakręcać inflację. Zapomnieliście o tym, że rolą państwa powinno być wspieranie ludzi najbardziej przedsiębiorczych i wyciąganie do nich ręki z pomocą, a nie po to, żeby zabierać kolejne podatki. Od przyszłego roku uderzycie w przedsiębiorców nowym ładem. Znam przykład stolarza, który od przyszłego roku zapłaci każdego miesiąca 400 zł więcej podatków przez wasze decyzje. Ostatnio opodatkowywaliście podwójnie wiele firm rodzinnych, a wiele przedsiębiorstw, takich, które mają wielkie hale produkcyjne, musi już nawet płacić podatek od deszczu. Jesteście współodpowiedzialni za tę inflację, bo nałożyliście szereg podatków: opłata mocowa, podatek handlowy, podatek od napojów słodzonych i taka jest prawda, że bierzecie za to współodpowiedzialność.

Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jako podlascy posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosiliśmy 27 poprawek do tego budżetu, regionalnych, bardzo ważnych poprawek. Dzisiaj chciałbym zaapelować do wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości, abyście ponad podziałami politycznymi spojrzeli na te poprawki, bo to są naprawdę bardzo ważne inwestycje dla województwa podlaskiego.

Jest to droga śmierci i jak najszybciej trzeba ją zrobić. Ale nie tylko to, bo również zwiększenie części oświatowej subwencji dla samorządów z województwa (Dzwonek) podlaskiego. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Ale również, szanowni państwo, oto poprawka, którą składam na prośbę pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Szanowni Państwo! Jeżeli chcecie dawać Bąkiewiczowi, dajcie też na pamięć o ludności cywilnej powstańczej Warszawy. Wysoka Izbo! Miały być nowe promy budowane w polskich, szczecińskich stoczniach, a jest rdzewiejąca stępka i międzynarodowy wstyd.

Miały być pieniądze dla psychiatrii dziecięcej, o co się upominamy cały czas. Co z tego zostało? Czarnkowy telefon zaufania. Nie potraficie realizować wielkich strukturalnych projektów, więc może dofinansujcie tych, którzy potrafią - samorządy? Wzywam posłów z PiS reprezentujących powiat gryficki o poparcie tej poprawki.

Wysoka Izbo! Z tego miejsca w imieniu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej chciałbym zaapelować o poparcie poprawki, którą przygotowaliśmy, według której należy przeznaczyć dodatkowe środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych zarówno jednostek Policji: komend wojewódzkich, komend powiatowych, jak i pracowników cywilnych Straży Granicznej. Jak państwo wiecie, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Policji wykonują bardzo ciężkie zadania i bardzo ciężką służbę w tej chwili na granicy. Od 1 stycznia funkcjonariusz średnio dostanie 677 zł podwyżki, natomiast jego kolega, pracownik cywilny - jedynie 167 zł. Oznacza to że blisko 30 tys. pracowników cywilnych komend powiatowych i wojewódzkich Policji będzie pracowało znowu za najniższą krajową. Tak być nie może. W imieniu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej bardzo państwa proszę, panie ministrze, o to żeby przyjąć poprawkę, która nada sens pracy pracowników cywilnych służb mundurowych, bo nie mogą pracować za tak strasznie niewielkie pieniądze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ileż to razy mówiliście o tym, że chcecie pomagać tym najsłabszym? Tymczasem fundujecie najdroższe w historii święta. Dzisiaj zakupy są dwukrotnie droższe niż w 2015 r., i to ci najsłabsi ponoszą największe konsekwencje tego, że mamy taką drożyznę, a wy nic z tym nie robicie.

To pokazuje, jak dbacie o tych najmłodszych, o tych najsłabszych. Na nich nie macie pieniędzy.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Szewiński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Taka sytuacja może doprowadzić wiele samorządów do upadłości. Przykład Częstochowy: subwencja oświatowa niższa o 150 mln od kwoty, jaką należy zabezpieczyć na realizację nałożonych zadań, zmniejszony podatek od osób fizycznych - 88 mln, do tego dochodzi koszt energii, podwyżek wynagrodzeń.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Tak nie może być. Trzeba coś z tym zrobić.

Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! PiS równa się drożyzna. PiS to galopujące ceny, to inflacja. Ale PiS to nie tylko drożyzna. PiS to również strata parudziesięciu miliardów złotych w KPO, dlatego że kłócicie się o izbę dyscyplinarną. PiS to również kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości. PiS to codziennie 500 osób, które umierają. Od początku pandemii to jest 150 tys. niepotrzebnych, nadwymiarowych śmierci. I przy tym wszystkim PiS to 4,89% PKB na ochronę zdrowia.

Poprzecie te poprawki?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Lasek, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Nieobecny Panie Premierze! Wysoka Izbo! Polskie lotniska w 2020 r. straciły 640 mln zł. W sytuacji gdy tak doświadczona pandemią branża lotnicza leczy rany, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwiększa wysokość opłat za świadczone przez siebie usługi terminalowe dla tych lotnisk. Kto za to zapłaci? Zapłaci pasażer. Bilety będą droższe, jak zresztą wszystko inne, zgodnie z waszym programem. Wspólnie z grupą posłów klubu Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy poprawkę przyznającą 50 mln dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie opłat terminalowych na dotychczasowym poziomie. Jeśli rzeczywiście zależy wam, aby polskie lotniska nadal były oknem na świat dla regionów, to poprzyjcie tę poprawkę. Branża lotnicza tego oczekuje. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten projekt budżetu jest skrojony pod działaczy i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na te wszystkie fundusze, instytuty są pieniądze. A co macie dla ludzi? Dla ludzi macie najdroższe święta od 20 lat. Otóż pomimo że jest bardzo wysoka inflacja - 7-procentowa - to jeśli ktokolwiek będzie chciał kupić karpia, zapłaci za niego 260% więcej niż rok temu, za dorsza zapłaci 220% więcej niż rok temu, za pomarańcze - 100% więcej niż rok temu, za rodzynki - 300% więcej niż rok temu, za śledzie - 50% więcej, za cukier - 25% więcej. Spełnia się niestety marzenie pana premiera Morawieckiego, który powiedział, że ludzie mają, delikatnie powiem, harować za miskę ryżu. Tak, bo nie ma nic innego do zaproponowania, nie zrobił nic, żeby ta inflacja i ta drożyzna były dużo lżejsze, tak jak jest w innych krajach. Chciałbym zapytać pana premiera Morawieckiego, ale nie ma go na sali.

Bardzo proszę, pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Dlaczego? Dlatego, że to jest najgorszy budżet, budżet drożyzny+, wirtualnej księgowości, rozpasany budżet, budżet wydatków na swoich, w tym na odprawy, zwiększenie wydatków dla premiera i prezydenta. Ograbianie samorządów, dla najuboższych dodatek osłonowy w wysokości 17 zł i na służbę zdrowia realnie, średnio ok. 5% w czasie pandemii. Domagamy się z tego z miejsca zwiększenia środków na służbę zdrowia o 20 mld, w szczególności na onkologię, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, szpitale powiatowe, oddziały pediatryczne w Puławach, Lubartowie, Janowie Lubelskim i na pokrycie wielu innych wydatków i kosztów inwestycji w województwach najuboższych na Lubelszczyźnie, która jest jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Podobno PiS ma nabożeństwo do tego, co narodowe, wszystkiego, co narodowe, ale jest wyjątek: chodzi o narodowe dziedzictwo kulturowe. Otóż mamy w Polsce 80 tys. zabytków nieruchomych, kilkaset tysięcy ruchomych.

Oczywiście nie muszę mówić, że większość tej kwoty idzie na obiekty sakralne. Gdyby nie praca samorządów, gdyby nie środki unijne, rozpadłaby się większość. To jest wstyd i hańba. Może wreszcie należałoby coś z tą hańbą narodową zrobić, aby to, co jest naszym dziedzictwem, to, co otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń, rzeczywiście było chronione. Województwo opolskie - 3366 zabytków. Ile ma wojewódzki konserwator zabytków? Bardzo proszę, pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Warszawiacy to nasi wspólni wyborcy, to pełnoprawni obywatele tego kraju, o których my w tej Izbie powinniśmy wspólnie zadbać. Tymczasem oni stali się jakąś waszą polityczną obsesją. Zamiast wyciągać konsekwencje, zmieniać swoje podejście, nastawienie, proponować inne rozwiązania, wy się na warszawiakach coraz bardziej chcecie odgrywać.

Dlatego chcielibyśmy wesprzeć Warszawę, zgłaszając poprawki.

Państwo macie szansę wyjść naprzeciw potrzebom warszawiaków i przestać ich traktować jako swoich politycznych przeciwników. My was sprawdzimy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jest drogo, ale wszyscy wiemy, że będzie jeszcze drożej. Rosną ceny żywności i to w szczególności niepokoi dziś Polaków. Dlaczego będzie drożej? Dlatego że rośnie także cena nawozów sztucznych. Co proponuje rząd? Wie pan minister? Pana kolega z rządu zaproponował izbom rolniczym, aby rolnicy przekierowali zainteresowanie na zwiększenie udziału w nawożeniu nawozami organicznymi. My proponujemy inne rozwiązanie: dopłaćmy rolnikom przy zakupie nawozów sztucznych. Zgłosiliśmy poprawkę. Proponujemy, żeby PiS (Dzwonek), jeżeli chcecie, aby żywność była tańsza, poparł poprawkę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak, tak. Proszę państwa, to nie jest dobry budżet dla Polski, to nie jest dobry budżet dla Polaków. Dlatego raz jeszcze apelujemy, byście państwo poparli nasze propozycje, żeby zwiększyć środki finansowe dla służby zdrowia, dla nauczycieli, dla pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej, prokuratury czy też sądów. Prosimy również i wnioskujemy o to, żeby znalazły się środki na dopłaty dla rolników, bo rolnicy są dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji, ale również na wsparcie dla samorządów, które są objęte stanem wyjątkowym.

Pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj na sali nie ma premiera Morawieckiego, ale kilka miesięcy temu tutaj był i tak mówił:

Nie pierwszy raz premier Morawiecki kłamał, okłamał Polki i Polaków, bo jest ostatnią osobą, której zależy na taniej energii, na tanim opale, na tanich produktach. Jest osobą, która za wszelką cenę chce zedrzeć z Polaków ostatni grosz, chce, aby im zostało tylko na michę ryżu. To jest prawdziwy obraz premiera Morawieckiego. Szanowni Państwo! To wasz znak firmowy, to jest znak firmowy PiS-u (Dzwonek), bo robicie wszystko, aby z podatku inflacyjnego do budżetu wpłynęło jak najwięcej. Pan poseł Michał Jaros, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Powtórzę po raz kolejny, bo mówię to ja i mówią eksperci: nie znacie się na gospodarce. Chyba nawet nie wiecie, co to jest gospodarka. Wydaje się wam, że to taka krowa, którą można wyłącznie doić, albo bank, z którego można wyłącznie brać pieniądze. W tym roku w rankingu systemów podatkowych państw OECD zajmujemy przedostatnie miejsce, za Włochami. Tym swoim Polskim Ładem uderzacie przede wszystkim w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, nie w korporacje, bo tych polskich firm nie stać na doradców podatkowych i na walkę o swoje prawa, o swoje pieniądze z fiskusem przez wiele lat. Pozostaje kilka pytań, szanowni państwo. Dlaczego niszczycie sukces gospodarczy kilku pokoleń Polek i Polaków? Dlaczego znacząco podnosicie obciążenia publiczne dla przedsiębiorców w tym bardzo trudnym i niestabilnym gospodarczo czasie? Dlaczego niszczycie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa? Dlaczego komplikujecie przepisy zamiast je upraszczać? Mam nadzieję, że znacie powiedzenie (Dzwonek), że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. A poza tym, pani marszałek, uważam, że Ostrołękę trzeba podliczyć i rozliczyć, a winnych ukarać. Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałam zapytać o przejrzystość finansów publicznych. Polakom ta informacja się należy. Wiemy, że 350 mld jest poza kontrolą Wysokiej Izby już dziś, a w tym budżecie na pięciu stronach, w 72 pozycjach jest prawie 40 mld zł ukrytych w różnych rezerwach, które zaraz po półroczu będą uruchamiane na różne wydatki, mniej lub bardziej potrzebne. Żądamy, aby tę kwotę przeznaczyć na realizację zgłoszonych przez nas poprawek. Ta kwota w zupełności wystarczy. Nie zgadzamy się, aby prawie 10% dochodów budżetu było ukryte w rezerwach. Są tu bardzo ciekawe zapisy, np. rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne (Dzwonek), w tym nowe zadania - tu są kolejne instytuty itd., itd. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Głogowski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałem zapytać o zabezpieczenie w budżecie na rok 2022 środków na likwidację bomb ekologicznych, czyli składowisk odpadów niebezpiecznych po byłych zakładach z branży chemicznej. Mam na myśli Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry, Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy, Zakłady Organika-Azot w Jaworznie czy Zakłady Przemysłu Barwników Boruta w Zgierzu. Na przykładzie pierwszego z nich, czyli Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry, mogę powiedzieć, że 2/3 prac przy zabezpieczeniu tych niebezpiecznych odpadów zostało już wykonanych, zrealizowanych w przeszłości, ale od roku 2015 żadne dalsze działania nie są realizowane, za to Ministerstwo Środowiska powołało specjalny zespół do spraw terenów zdegradowanych. W odpowiedzi na moją interpelację z lutego br. wiceminister klimatu i środowiska poinformował mnie, że rekultywacja terenów po tych zakładach przemysłu chemicznego będzie finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Polska już traci z tego tytułu pieniądze. Bardzo proszę, pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! W projekcie ustawy budżetowej nie znalazłam zapewnienia środków na podwyżki płac dla pracowników socjalnych, pielęgniarek, opiekunek, opiekunów, rehabilitantów, terapeutów w domach pomocy społecznej. Każda z tych grup zawodowych, obciążonych psychicznie i fizycznie szczególnie w okresie pandemii, wykonuje niezmiernie odpowiedzialną pracę, poświęca się dla osób niesamodzielnych, dla osób chorych, osób z niepełnosprawnościami. DPS-y nie są placówkami medycznymi i w związku z tym pracownicy, wykonując bardzo podobne obowiązki jak pracownicy zakładów opiekuńczo-leczniczych czy pielęgniarki na oddziałach szpitalnych, nie są objęci siatką płac obowiązującą w opiece zdrowotnej. Ta dysproporcja wynagrodzeń powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry z domów pomocy społecznej. Kiedy ten problem zostanie rozwiązany? Jutro? Pojutrze? W domach pomocy społecznej będą chorzy, będą osoby starsze, będą osoby z niepełnosprawnościami, ale nie będzie nikogo, kto będzie mógł tymi osobami się zająć, kto będzie je pielęgnował i będzie się nimi opiekował. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! To nie jest budżet robiony z myślą o Polakach, to jest budżet dla PiS-u. Ile jest tam pieniędzy ukrytych dla poprawy samopoczucia rządu PiS-u, tego dokładnie nie wiemy, proszę państwa, bo rząd się wyżywi - nawet jak będzie drożyzna, to rząd dodrukuje sobie po prostu pieniądze. Niedofinansowana jest służba zdrowia, która funkcjonuje już na krawędzi, rolnictwo chyli się ku upadkowi, energetyka jest w sytuacji krytycznej, ignorancja co do odnawialnych źródeł energii itd., itd. Koalicja Obywatelska złożyła doskonałe propozycje poprawek. Proszę je przyjąć. Budżet jest do poprawy w każdej części, bo to jest jedna wielka niewiadoma. Tak naprawdę nie wiemy, jakie jest zadłużenie naszego państwa, ale dla rządu w tej chwili to nic nie znaczy. Dziennie, proszę państwa, umiera pół tysiąca osób na COVID. Przerażające, bo wszyscy podeszli do tego jak do normalnej sytuacji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Elżbieta Gapińska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Nazwa waszej partii to synonim drożyzny.

Podoba wam się też budżet na przyszły rok. To budżet, w którym brakuje pieniędzy na wszystko: na zdrowie, na ekologię, na transformację energetyczną. Te pieniądze po prostu im się należą za to, że dbają oni o wasze dzieci, że wytrzymują w szkole, w której próbujecie ich indoktrynować i próbujecie indoktrynować dzieci. Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po pierwsze, PiS to drożyzna. Po drugie, ma rację pani poseł Skowrońska, która mówi, że to jest wasza wina, wielka wina. Po trzecie, szukam w budżecie na rok 2022 pieniędzy na drogi. Otwieram portal Ministerstwa Infrastruktury, zakładkę: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dawniej Fundusz Dróg Samorządowych, dawniej schetynówki, i szukam rozstrzygnięcia naboru wniosków na 2021 r. Tam gdzie są zadania obwodnicowe, nie ma rozstrzygnięcia, a wiem, że wszystkie procedury zostały już zakończone. Leży to na biurku u premiera Morawieckiego i czeka na podpis. Nie podpisuje. Dlaczego?

Czekają obwodnice w województwie lubuskim. Północna obwodnica Gorzowa, południowa obwodnica Zielonej Góry, obwodnice Słubic, Kożuchowa, Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą.

Bardzo proszę, pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek!

14 mln zł. Taka jest wasza prawdziwa twarz. Mówicie: przez 8 lat Platformy Obywatelskiej.

To są konkrety.

Sprawdźmy.

Bardzo proszę, pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Pani Marszałek! Panie Ministrze Mejzo! Mam pytanie do premiera Morawieckiego. Czy to prawda, że wysłał pan SMS-a do wysokiego urzędnika Komisji Europejskiej z prośbą o pomoc, aby Polska otrzymała pieniądze, i podpisał się pan, cytuję: ostatni Europejczyk w rządzie? Czy pan premier chciał przez to przekazać, że rządzą nami nie-Europejczycy? W czyim imieniu obecny rząd realizuje swoją antyeuropejską politykę? Rozmawiamy tu o budżecie. Wszyscy cierpimy z powodu wysokiej inflacji i drożyzny.

Kto w takim razie rządzi Polską? Panie Premierze! Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czy państwo w ogóle czasami chodzicie do sklepu spożywczego? Jeśli chodzicie, to doskonale wiecie, że to jest prawda. Przez ostatnie 6 lat waszych rządów ceny idą w górę, w sklepach spożywczych w sposób niewyobrażalny. Przez ostatni rok podstawowy koszyk zakupów podrożał o 35%. Fundujecie Polakom najdroższe święta Bożego Narodzenia od 20 lat. Co planujecie w budżecie na przyszły rok? Kolejne 214 mln zł wzrostu wydatków w kancelarii premiera. 2 mld zł na publiczną propagandę w TVP.

Nie.

Bardzo proszę, pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo! To jest właśnie wynik waszych działań, wynik tego, że drożyzna w Polsce jest zasługą Prawa i Sprawiedliwości. To, że mamy drogie paliwo, to, że mamy drogą energię, to, że produkty spożywcze są drogie, to jest również wynik pracy nie kogo innego jak szefa komisji energii i aktywów państwowych Marka Suskiego. Szanowni Państwo! To właśnie dzisiaj przez te rządy będziemy mieli najdroższe święta od 20 lat. Ale aby zrekompensować radomianom, mieszkańcom ziemi radomskiej te wielkie wydatki, mam wielką prośbę - tu przed chwilą był były kandydat na prezydenta Wojciech Skurkiewicz czy były prezydent Andrzej Kosztowniak - zagłosujcie za radomskimi poprawkami.

Panie Ministrze! Dlaczego opracowując projekt budżetu, nadal zapominacie o pracownikach sądów i prokuratur, o pracownikach cywilnych Policji? Poprzyjcie państwo poprawki w ich sprawie. Ale istotne jest pytanie, dlaczego Fundusz Medyczny nadal nie jest funduszem ratującym ludzkie życie, dlaczego nie jest funduszem pomagającym ciężko chorym. Obiecano w ramach tego funduszu ponad 4 mld zł, a w tym roku wydano zaledwie 170 mln zł. Dlaczego osoby dotknięte chorobami rzadkimi drżą z niepewności, drżą, czy będą objęte niezbędnymi terapiami, czy nagle zostaną ich pozbawieni. Proszę państwa, jak w ramach budżetu rząd chce pomóc chorym, np. na mukowiscydozę, jak chce w przyszłym roku pomagać tym, którzy cierpią na nocną napadową hemoglobinurię? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Proponuję zmianę nazwy waszej partii, bo nie macie nic wspólnego ani z prawem, ani ze sprawiedliwością. PiS to drożyzna. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 - już dziś można to powiedzieć - przynajmniej w części założeń jest nieaktualny. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest nad wyraz wysoka inflacja i jej konsekwencje. Do tego dochodzi kreatywna księgowość i przepuszczanie ogromnych środków poprzez różnego rodzaju agendy, które nie są ujęte w budżetowym planie. Tak ma wyglądać przejrzystość finansów publicznych. To wszystko pokazuje, że ustawa budżetowa już dawno przestała odzwierciedlać faktyczny stan finansów państwa.

Chciałam prosić o pisemną odpowiedź na te poprawki, które z uzasadnieniem na pewno zostaną nieprzegłosowane. Potrzebne jest bardzo wiele inwestycji na południu Polski i proszę o traktowanie południa Polski w inny sposób, nie tak jak traktujecie do tej pory, po macoszemu. Bardzo proszę, pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Kreatywna księgowość, wyprowadzanie pieniędzy poza budżet państwa, ogromne rozpasanie władzy. To widzimy, czytając ten budżet. Niestety pokazujecie także i tym budżetem, i swoją postawą tę sytuację. Widzimy tę drożyznę, otrzymując rachunki. Niestety jeśli tak dalej będziecie rządzić, będzie tylko gorzej. A Polacy dzisiaj zasługują na odpowiedzialną władzę, także odpowiedzialną władzę, która przyjmie Fundusz Odbudowy, która będzie działała zgodnie z prawem, przepisami prawa, na podstawie i w granicach tego prawa, która będzie przestrzegała praworządności, bo to podstawowa wartość, którą powinniśmy się szczycić i dumnie pokazywać. Dzięki temu możemy także pozyskać ważne środki dla przedsiębiorców, aby walczyć ze skutkami pandemii. Dzisiaj potrzebne są zmiany i przyjęcie poprawek dotyczących podwyżek dla pracowników cywilnych Policji, dla chociażby nauczycieli, ale także przyjęcie ważnych poprawek w sprawie Zagłębia Dąbrowskiego. na które czekają samorządy i mieszkańcy. Koniec rozpasania władzy, dzisiaj należy wspierać mieszkańców i obywateli. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Budżet na 2022 r. to najlepszy dowód na nieudolność PiS-u. To kolejne zadłużanie państwa o 140 mld zł, to nowe podatki. Wielu małych przedsiębiorców już dziś zastanawia się, czy w przyszłym roku nie będzie musiało ograniczyć bądź też zlikwidować swojej działalności gospodarczej. Nie ma pieniędzy na słuszne, właściwe podwyżki dla nauczycieli, dla pracowników administracji, sądów, prokuratur, pracowników Policji i Straży Granicznej czy pomocy społecznej. Nie ma pieniędzy na ochronę zdrowia, w tym na psychiatrię dziecięcą.

Zróbcie więc, proszę, najlepszy prezent: nie szkodźcie już więcej, zrezygnujcie i odejdźcie. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Pani Marszałek! Budżet państwa to powinna być nadzieja na lepsze życie rodzin pracowników budżetowych. Wielu z nich dziś otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w placówkach terenowych 60% z nich otrzymuje właśnie wynagrodzenie minimalne. Mówią tak: pora zmienić pracę, nie można tak ciągle do emerytury na płacy minimalnej. Czy w tym budżecie nastąpi radykalna poprawa sytuacji pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych pracowników budżetowych? Drugie pytanie: Czy w tym budżecie znajdują się środki na modernizację i remont drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno - Żydowo - Czeluśnin?

Szanowni Państwo! Budżet na rok 2022 będzie zawierał bardzo ważną pozycję, przełom po ostatnich 30 latach, jeżeli chodzi o kwestię finansowania nauki języka polskiego w Niemczech - aż 30 mln zł, po przyjęciu przez Sejm poprawki pana ministra Czarnka, z inicjatywy Solidarnej Polski.

To było ostatnie pytanie.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Wartość umów zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wtedy wynosiła 167 mln. To są materialne i złotówkowe efekty tego, jak wyglądają nakłady na psychiatrię dziecięcą.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonała retaryfikacji taryf w zakresie psychiatrii dziecięcej, psychiatrii.

Tylko w przeciągu 2 lat zwiększamy ten budżet o ponad 1 mld zł, co pokazuje w oczywisty sposób, że jest to dla nas priorytet, i to związany z wdrażaniem pewnych reform, i priorytet związany z finansowaniem tego obszaru. Te ponad 300 mln zł, o których mówiłem, w zakresie wzrostu wycen mamy zabezpieczone. Co więcej, myślę, że wielokrotnie w toku prac Komisji Zdrowia mówiliście państwo o dużym udziale wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Teraz nie jest to precedens, tylko jest to norma. Jest to norma, która wynika również z funkcjonowania ustawy 6%, ustawy gwarantującej określony poziom nakładów na ochronę zdrowia. Myślę, że warto wrócić się do kwestii dynamiki nakładów, bo dzisiaj z mównicy padało głównie hasło związane z tym, że liczymy nakłady w stosunku do 2 lat wstecz i że jest to nie efektywne, niekorzystne dla systemu ochrony zdrowia.

W 2010 r. kształtowały się na poziomie prawie 5% PKB liczonego według tej nomenklatury, o której mówię, czyli 2 lata wstecz.

Pani poseł, szanowni państwo, pomogliśmy wydatnie.

Te wydatki pochodzą albo z budżetu państwa, albo z rezerw celowych będących w dyspozycji ministra zdrowia czy innych dysponentów, albo z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.

To ogromne postępowania konkursowe.

Chcę przypomnieć, że gdy w roku 2014, w grudniu, Komisja Europejska przyjęła do realizacji Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko”, to ówczesne Ministerstwo Zdrowia pierwsze konkursy ogłosiło w październiku, po 10 miesiącach. Czy uważam, że to jest skandaliczne? Czy uważam, że były opóźnienia?

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z ustawą miała określony czas na przygotowanie wykazów technologii innowacyjnych. Jeden miał powstać pod koniec lutego, drugi pod koniec sierpnia 2021 r., potem były poddane analizie, a następnie skierowane jako pewne oczekiwanie i życzenie ministra finansów do firm farmaceutycznych, które mogą, ale nie muszą - bo nie jesteśmy w stanie ustawowo nikogo zmusić - złożyć stosowne wnioski refundacyjne.

Nie bardzo rozumiem, czy ma być skierowana na pomoc związaną z pandemią, czy na pomoc związaną ze świadczeniami COVID-owymi, czy ogólnie na wzmocnienie sektora ochrony zdrowia. Zachęcam do obiektywnej analizy tych zwiększeń, których dokonaliśmy w ostatnim roku, i przypominam jeszcze raz, że wzrost finansowania ochrony zdrowia w stosunku do tego, co było 2 lata temu, to prawie 30%.

To był wkład budżetu państwa w nakłady na sektor ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo.

Wysoki Sejmie!

Zatem nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy te poprawki uzyskają poparcie strony rządowej. W pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do problematyki inflacji.

Takie były prognozy rynkowe.

Inflacja jest obecnie problemem ogólnoświatowym. Podam przykład państwa strefy euro, naszego sąsiada, Litwy. Jest to członek strefy euro. Zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Cel inflacyjny EBC jest niższy niż Narodowego Banku Polskiego z przedziałem, a Europejski Bank Centralny nie podnosi stóp procentowych.

Myślę, że nie spodziewali się tak wysokiej inflacji. Wracając do przejrzystości, transparentności finansów publicznych, nie mogę się zgodzić z tezą, że 40% jest poza kontrolą.

Jeżeli chodzi o transparentność, to myślę, że transparentność finansów publicznych zapewniają rozwiązania unijne, tzw. statystyki ESA.

Padło tu również pytanie pana prof. Rosatiego o stawki forward rate agreement. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o narażenie na ryzyko dotyczące stóp procentowych, to jesteśmy dobrze przygotowani z tego względu, że ok. 3/4 długu Skarbu Państwa ma oprocentowanie stałe, więc zmiany stawek, przynajmniej w przyszłym roku, nie powinny mieć aż tak zasadniczego znaczenia. Padały również pytania o jednostki samorządu terytorialnego. Z tego miejsca mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa, niemal 100-procentową, oszacować, że rok 2021, podobnie jak rok 2020, jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo zamkną nadwyżką. Możemy tylko dyskutować, czy ta nadwyżka będzie 10-cyfrowa czy 11-cyfrowa, niemniej na pewno rok zamknie się nadwyżką.

W mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego dość powszechne jest, Wysoki Sejmie, odniesienie, że środków w jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza na inwestycje w tym roku, jest rekordowa ilość. Trzeba mieć na względzie dodatkowe 8 mld subwencji rekompensującej oraz 4 mld zł wydatków na sieci wodno-kanalizacyjne, które trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, gdzie ubytki w tej sieci były największe. Pojawiały się również pytania związane z podwyżkami, w szczególności w służbach mundurowych. Ustawa budżetowa zakłada wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 4,4%, odblokowanie 3-procentowego funduszu nagród. Ponadto nie należy zapominać o rozwiązaniu doraźnym w roku bieżącym, czyli dodatkowym 6-procentowym funduszu na działania promotywacyjne.

Również pracownicy cywilni będą mieli podwyżki w wysokości ok. 356 zł na etat. Dziękuję bardzo, panie ministrze. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja Infrastruktury przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1836.

Marszałek Sejmu proponuje, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowch oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (druki nr 1516 i 1821) Proszę pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, druk nr 1516.

Podczas rozpatrywania tej ustawy zgłoszono dwie poprawki, które zostały przez komisję przyjęte. W projekcie ustawy przewiduje się ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Proponowane zmiany przepisów wynikają z programu Polski Ład, w którym zapowiadano inicjatywę uwolnienia rolniczego handlu detalicznego. Celem ustawy jest przede wszystkim zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak sklepy, restauracje, stołówki. To terytorium całego kraju, obecnie jest to województwo. Chcemy to rozszerzyć na cały kraj, bo uważamy, że rolniczy handel detaliczny w Polsce dobrze się rozwija. Jest on przede wszystkim dedykowany rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Przyjęcie powyższego rozwiązania ograniczy liczbę osób obowiązanych do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a z drugiej strony umożliwi pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych. Procedowana ustawa jest oczekiwana przez rolników, którzy coraz częściej decydują się na rolniczy handel detaliczny, dzięki czemu my wszyscy, konsumenci, mamy zdrową żywność. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, druki sejmowe nr 1516 i 1821. Na posiedzenie Sejmu wraca bardzo istotny projekt ustawy będący realizacją inicjatywy nazwanej: uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, zawartej w dokumencie rządowym Polski Ład. Warto po raz kolejny podkreślić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zwiększyć możliwości rolników wynikające z wprowadzonego w 2017 r. rolniczego handlu detalicznego, który cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Przypomnę, że obecnie w Polsce taką formę sprzedaży żywności prowadzi kilkanaście tysięcy rolników. W przedmiotowym projekcie ustawy proponuje się ułatwienie dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz ulgi w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym celem proponowanych zmian jest wspomniane wcześniej zwiększenie możliwości rozwoju w Polsce działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Rozwiązania przewidziane w projekcie obejmują przede wszystkim, po pierwsze, rozszerzenie na cały kraj obszaru zbywania żywności niezwierzęcego pochodzenia wyprodukowanej w ramach RHD do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta, takich jak np. sklepy, restauracje czy stołówki, po drugie, zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom, po trzecie, podwyższenie kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego z obecnych 40 tys. zł do 100 tys. zł. W dniu 1 października 2021 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu na 38. posiedzeniu Sejmu RP, na którym projekt skierowano do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu 8 grudnia 2021 r. przyjęła projekt jednogłośnie. Jako członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwolę sobie poinformować, że w trakcie prac komisji przyjęto kilka poprawek do projektu ustawy, z których najistotniejsze dotyczyły uwzględnienia uwagi Komisji Europejskiej zgłoszonej w ramach procedury notyfikacji w celu zapewnienia zgodności proponowanych rozwiązań z przepisami prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz zmiany daty stosowania przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystnej dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. Komisja Europejska zgłosiła również uwagę do projektu dotyczącą obszaru, na którym może być zbywana żywność pochodzenia zwierzęcego wyprodukowana w ramach RHD do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta. Zdaniem Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dostawy takiej żywności w odróżnieniu od żywności pochodzenia niezwierzęcego powinny być prowadzone lokalnie, nie zaś na całym terytorium Polski, o ile do działalności RHD mają mieć zastosowanie uproszczone wymagania sanitarne. W wyniku przyjęcia poprawki uwzględniającej uwagę Komisji Europejskiej w projekcie zakłada się, że powiększony zostanie obszar - do terytorium całego kraju - na którym będą prowadzone dostawy żywności pochodzenia niezwierzęcego wytwarzanej w ramach RHD do innych zakładów. Z kolei obszar takiego zbytu w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego pozostanie bez zmian. Pozostałe najistotniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie, tj. dotyczące zniesienia maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom oraz podwyższenia kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego, nie uległy zmianie. Podsumowując, należy zdecydowanie stwierdzić, że projekt ustawy jest kolejnym dużym krokiem w celu udoskonalenia rolniczego handlu detalicznego. Znakomicie wpisuje się on w koncepcję skrócenia łańcucha dostaw: od pola do stołu. Podjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości inicjatywa ustawodawcza wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, ale również konsumentów. Przyjęcie projektu przedmiotowej ustawy sprawi, że dostęp do zdrowej, polskiej żywności będzie jeszcze lepszy, oraz ma dużą szansę pozytywnie wpłynąć na promocję rolniczego handlu detalicznego. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera proponowane rozwiązania i wnosi, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić przedmiotowy projekt ustawy. Bardzo proszę, pan poseł Kazimierz Plocke, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Zanim przejdę do omówienia projektu ustawy o rolniczym handlu detalicznym, najpierw kilka sprostowań. Po pierwsze, wbrew temu, co napisano w uzasadnieniu, proponowane przepisy nie wynikają z dokumentu rządowego Polski Ład. Jak wiadomo, rząd Polskiego Ładu nie przyjął jako swojego programu, a zatem jest to program partyjny Zjednoczonej Prawicy.

Naszym zdaniem tak się nie stanie. Z czego wynikają nasze obawy?

Zatem dedykowana ustawa ma objąć ok. 1% gospodarstw rolnych. Według obecnych przepisów produkcja żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego o wartości do 40 tys. zł jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. W postulowanych przepisach proponuje się podniesienie tej kwoty do 100 tys. zł. My w dalszym ciągu pytamy, dlaczego tej kwoty nie można podwyższyć np. do 200 tys. zł. Dziś wiemy, że kwoty 40 tys. zł nie da się utrzymać, ponieważ rząd planuje zwolnić z płacenia podatku dochodowego wszystkich obywateli osiągających dochody roczne do 30 tys. zł. Pozostawienie kwoty 40 tys. zł dla rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego byłoby groteską. Uważamy, że tę kwestię należy rozstrzygnąć w ten sposób i kwotę należy podwyższyć chociażby ze względu na galopującą inflację. Z dostępnych statystyk wynika, że rolnicy nie garną się do przekraczania przychodów na poziomie 40 tys. zł i uiszczania 2% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dlaczego tak mało? Jeśli to się zmieni, zainteresowanie rolników rolniczym handlem detalicznym z pewnością wzrośnie.

Przyznacie państwo, że to nie za wiele. To oznacza, że za 15,5 mln zł chcecie zachęcić rolników do wdrożenia skomplikowanego i obciążonego nadmierną biurokracją systemu. Warto zapamiętać, że w Polskim Ładzie wskazano ustawy, m.in. Kodeks rolny, akcyzę i prezentowany dzisiaj projekt ustawy o rolniczym handlu detalicznym. Naszym zdaniem to o wiele za mało. A zainteresowanych odsyłam do programu partyjnego Polski Ład, s. 78. Panie ministrze, jeszcze dwie kwestie. Komisja Europejska sformułowała uwagi w ramach notyfikacji tego projektu ustawy. Chciałbym zapytać: W jaki sposób i czy wszystkie uwagi komisji zostały uwzględnione? Czy nie istnieje konieczność poinformowania Komisji Europejskiej o uwagach wdrożonych do rzeczonego projektu ustawy przed głosowaniem? Druga kwestia to sprawa wejścia ustawy w życie. Zapis mówi, że to jest 14 dni od ogłoszenia ustawy, co oznacza, że ustawa będzie prawem obowiązującym na początku 2022 r. Natomiast chciałem spytać: Co z systemem podatkowym dla rolników, który powinien obowiązywać od 1 stycznia roku budżetowego? Podsumowując - mój klub poprze projekt ustawy, ale oczekujemy od pana ministra odpowiedzi na nasze wątpliwości i uwagi.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy wobec rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Rolniczy handel detaliczny to specyficzna, funkcjonująca od 2017 r. forma handlu detalicznego dedykowana rolnikom. Dane z Inspekcji Weterynaryjnej i inspekcji sanitarnej wskazują, że pod koniec 2020 r. rolniczy handel detaliczny prowadziło w ramach produkcji zwierzęcej ponad 11 tys. gospodarstw, a w ramach produkcji roślinnej ponad 1500 gospodarstw. Nie jest to duża skala - stanowi to niecały 1% wszystkich gospodarstw rolnych. Omawiany projekt ustawy zawiera kilka kluczowych zmian w funkcjonowaniu rolniczego handlu detalicznego. Po pierwsze, w projekcie ustawy proponuje się zniesienie maksymalnych limitów żywności w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym. Druga zmiana polega na podwyższeniu limitu przychodów ze sprzedaży zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Po trzecie, w projekcie ustawy proponuje się zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, do terytorium całego kraju. Obecnie obszar ten jest ograniczony do województwa oraz powiatów lub miast sąsiadujących z tym województwem. Po czwarte, zmianie ulega definicja pojęcia: rolniczy handel detaliczny. W przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik - np. przetworzone produkty mięsne, mleczne czy gotowe posiłki - wprowadzono zmianę, że żywność powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Co do zasady proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Ich celem jest wzmocnienie pozycji rolników na rynku spożywczym i skrócenie łańcuchów dystrybucji, tak aby rolnicy mogli przedstawiać swoją ofertę bezpośrednio konsumentom.

W trakcie pierwszego czytania zwróciłam uwagę na ryzyko nadużyć, które mogą wynikać ze zmiany definicji rolniczego handlu detalicznego. Ta zmiana mówi o tym, że żywność powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. Ta zmiana powoduje, że jeżeli w gotowym posiłku z własnej uprawy są tylko rzodkiewki, a reszta to np. ryż z Chin, soja z USA, mięso i pomidory z Hiszpanii, to taki posiłek będzie można sprzedawać bez podatku dochodowego. Na tę samą kwestię zwróciła uwagę Krajowa Rada Izb Rolniczych w swojej opinii z 17 września. Rada podaje przykład rolnika, który uprawia tylko groszek i dodaje go do potraw w różnej formie, albo rolnika utrzymującego kilka tuczników słoninowych i dodającego tłuszcz z tych tuczników do wszystkich potraw. Zgodnie z tym projektem ustawy, nawet jeżeli wszystkie inne składniki pochodzą z zakupu z innych źródeł, taki producent potraw będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Krajowa Rada Izb Rolniczych proponuje także konkretne rozwiązania zmian w projekcie ustawy, np. zapis, że jeden z dwóch głównych składników produktu złożonego winien pochodzić w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Ewentualnie mogłoby też być określenie procentowe stosowane w innych krajach. Niestety ta sprawa nie została naprawiona w projekcie ustawy i uważam, że jest to duże niedopatrzenie. Pomimo tego Lewica zagłosuje za tą ustawą, gdyż naszym zdaniem korzyści z niej płynące przewyższają ryzyka z nią związane. Pan poseł Mirosław Maliszewski, Koalicja Polska. Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie!

To jest kontynuacja, tylko pod zmienioną nazwą. Cóż to takiego jest ta sprzedaż bezpośrednia albo rolniczy handel detaliczny? Czym to się różni od podstawowej produkcji rolnej?

Zawsze było takie niebezpieczeństwo, że produkty wytworzone na bazie produktów zwierzęcych, np. mleka czy mięsa, muszą spełniać określone warunki higieniczne, ponieważ one podlegają skomplikowanej obróbce i mają specyficzne właściwości. A więc aby ludzi nie narażać na niebezpieczeństwo, zawsze zwracamy uwagę na to, aby przetwarzanie produktów zwierzęcych odbywało się zgodnie z zasadami higieny i wymogami weterynaryjnymi czy bezpieczeństwa produkcji żywności. Trochę inaczej to wygląda w przypadku produktów roślinnych, gdzie ta obróbka jest łatwiejsza.

Dlatego trzeba stopniowo uwalniać rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią, po to aby to miejsce na rynku, które mają duże podmioty, pomału zajmowali rolnicy, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w formie przerobionej.

Dzisiaj on dotyczy głównie małych rolników, którzy posiadają gospodarstwa rozdrobnione i którzy ze względu na mały wolumen produkcji muszą zająć się przetwórstwem, po to aby zwiększyć wartość dodaną, aby uzyskać dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży produktów przetworzonych do swojego gospodarstwa.

Po drugie, te produkty dotyczą wąskiego wycinka działalności rolniczej, dlatego że jest bariera w racjonalnym sprzedaniu tych produktów. Nie ma dzisiaj dużego odbiorcy, który byłby w stanie od rolnika trochę większego niż mały, drobny kupić te produkty i je zagospodarować.

Pozostaje więc pytanie: Czy nie warto - ono jest retoryczne, bo na pewno warto - rolników wesprzeć w relacjach handlowych wobec dużych odbiorców, dużych graczy na rynku?

Jeżeli te wszystkie rozwiązania byśmy wprowadzili w życie, to moglibyśmy uznać, że ten rodzaj produkcji rolnej ma pewną szansę.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Wysoka Izbo! Natomiast dzisiaj w Sejmie powinniśmy dyskutować o tym, co nadchodzi, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, a co jest sygnowane nazwiskiem polityka PiS-u, który jednocześnie wywodzi się z PSL-u, czyli pana Janusza Wojciechowskiego. A nadchodzi trzęsienie ziemi nie tylko w polskim, ale i europejskim rolnictwie, szanowni państwo, pod nazwą: Europejski Zielony Ład. Tak, chodzi o Europejski Zielony Ład, o którym służba naukowa Komisji Europejskiej napisała, że doprowadzi on do dramatycznego załamania rolnictwa i produkcji rolnej w skali całego kontynentu. Europejski Zielony Ład, który doprowadzi do tego, że Europa z eksportera żywności stanie się znaczącym importerem żywności. Europejski Zielony Ład, który doprowadzi do tego, że dziesiątki, setki tysięcy gospodarstw w Polsce, gdzie i tak nie jest lekko, staną na skraju bankructwa, przestanie opłacać się produkcja. Będzie likwidacja do kilkudziesięciu procent, jeśli chodzi o produkcję mięsa, o produkcję zwierzęcą, o hodowlę, również jeśli chodzi o mleczarstwo, prognozowany spadek jest nawet kilkunastoprocentowy. To jest, proszę państwa, ta kwestia, nad którą dzisiaj Sejm powinien debatować.

Jaka jest debata? Gdzie jest krzyk rozpaczy, który powinien być tutaj wydawany, i gdzie jest sprzeciw wobec tego europejskiego, unijnego szaleństwa, które dzisiaj uderza w branżę i które konsoliduje opór rolników na terenie całej Europy? To są poważne wyzwania, to jest poważna odpowiedzialność wobec samowystarczalności żywnościowej kraju, wobec kolejnych pokoleń Polaków, którzy zmierzą się z kolejnymi utopijnymi projektami Unii Europejskiej. Dzisiaj trzeba z tego miejsca bardzo stanowczo powiedzieć: dosyć, dosyć tego unijnego szaleństwa sygnowanego przez Janusza Wojciechowskiego, przez PiS-owskiego komisarza z PSL-owskim rodowodem.

Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Szanowni Państwo! Tak jak tu już było powiedziane, deklarowanym przez rząd celem ustawy jest wprowadzenie pewnych ułatwień w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Proponuje się szereg zmian, które według rządu mają dać impuls do zwiększenia dochodów mieszkańców terenów wiejskich, m.in. zmianę definicji rolniczego handlu detalicznego, rozszerzenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności, czy doprecyzowanie kwestii pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Efektem tej ustawy ma być również skrócenie w niektórych obszarach drogi z pola na stół. Oczywiście cele te są bliskie Polsce 2050. Pytanie jest jednak takie, czy ta nowelizacja rozwiąże problemy, które trapią dziś polską wieś. Z pewnością ten pomysł rządu nie jest remedium na wszystkie problemy polskiej wsi, choć myślę, że nie możemy tutaj wszyscy oprzeć się wrażeniu, że pan minister mówił o tej ustawie tak, jakby to był Święty Graal rolnictwa. Po pierwsze, wąski zakres obowiązywania zmian. Z rolniczego handlu detalicznego skorzystało zaledwie 12 876 gospodarstw, czyli stosunkowo niewielka grupa, a koszt tych zmian to zaledwie 15,5 mln zł.

Myślę, że te problemy, panie ministrze, są o wiele głębsze, a na to nakłada się dzisiejsza sytuacja, czyli szalejąca drożyzna, wysoka inflacja, brak odwagi w kreowaniu rozwiązań. Niestety ten projekt tego wszystkiego nie zapewnia. Podczas prac nie wyjaśniono też części naszych wątpliwości dotyczących tego, czy przypadkiem nie dojdzie do takiej sytuacji, w której pod rolniczy handel zostaną podciągnięte takie działalności, gdzie wykorzystuje się składniki importowane, co byłoby oczywiście ze szkodą dla rolnictwa. W tych sytuacjach Polska 2050 Szymona Hołowni będzie zdecydowanie walczyła o prawa polskiej wsi, o prawa rolników. Te rozwiązania (Dzwonek), choć wąskie, idą w dobrym kierunku. W związku z tym Koło Parlamentarne Polska 2050 będzie ten projekt ustawy popierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytanie? Zamykam listę. Jako pierwszy pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. 1 minuta na zadanie pytania. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska.

Szanowni Państwo! Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o kondycji polskiej wsi, rozmawiamy o kondycji gospodarstw domowych indywidualnych rolników. Ostatnio byłem w Namysłowie, ostatnio byłem w Kluczborku, ostatnio rozmawiałem z rolnikami w Głubczycach i wszyscy rzeczywiście martwią się rosnącymi cenami, szczególnie cenami paliwa, cenami gazu, który jest bardzo często wykorzystywany do różnych czynności związanych z produkcją na wsi. Dla nas, szanowni państwo, dzisiaj jest bardzo ważny wniosek: tym, co jest największym zagrożeniem dla polskiej wsi, jest unijny regulacyjny green deal.

Na to nie możemy pozwolić. Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła opinię na temat ustawy i prosiłbym o pisemne odniesienie się do stwierdzenia, które zacytuję: Pewne wątpliwości może budzić zaproponowany przepis dotyczący pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności innej niż pierwotna, stanowiący, iż żywność produkowana w ramach RHD zawierająca więcej niż jeden składnik powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Chciałbym zapytać pana ministra o metody weryfikacji oraz ewentualne sankcje, które mogą spotkać rolników działających z naruszeniem uchwalonych przepisów.

Kto i na jakiej podstawie będzie stwierdzał, czy kiełbasa sprzedawana na przydrożnym straganie została zrobiona ze świni hodowanej w gospodarstwie tego rolnika czy jego sąsiada? Jakie metody weryfikacji ustawodawca proponuje, aby stwierdzić, czy jabłka stanowiące przedmiot transakcji urosły w sadzie pana Kowalskiego, a nie w sadzie pana Nowaka? Uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedź w tej sprawie na piśmie w związku z wieloma pytaniami, które otrzymuję. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

To przesłania zarówno władzy, jak i większości z Prawa i Sprawiedliwości sprawy polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa i bardzo źle oddziałuje na państwo polskie.

Dotyczy ono kontroli.

Pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa jest w swoim założeniu słuszna.

Po pierwsze, jaka jest skala środków w ramach planu strategicznego nowej polityki rolnej, aby wspierać rolników m.in. w proponowanych zakupach sprzętu? Czy będą np. ośrodki doradztwa rolniczego?

W jakim zakresie ta ustawa wejdzie w życie? Od kiedy tak naprawdę ustawa zacznie obowiązywać z uwagi na zmiany podatkowe w Polsce? Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam trzy uwagi krytyczne.

Uważam, że na tym etapie tę kwotę trzeba podnieść. Trzeci element.

Pozytywy. To jest rzecz niezwykle ważna. Z pola na stół.

Bardzo proszę, pani poseł Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Na pewno rolniczy handel detaliczny nie uzdrowi całego rolnictwa. Jest to jeden z elementów, który umożliwia rolnikom podniesienie opłacalności produkcji. Panie Ministrze! Czy przygotowane są rozporządzenia, które zwiększą kwoty na przetwórstwo w ramach rolniczego handlu detalicznego? Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Czy resort ma jasną diagnozę? Czy ta interwencja legislacyjna rzeczywiście rozwiązuje problemy? Bo wydaje się, że mamy taką sytuację: rolnik ma co sprzedać, ale nie ma komu sprzedać, nie ma gdzie sprzedawać, czyli chodzi o infrastrukturę, i czasami nie ma kiedy. Tzn. mówimy o sytuacji, że w Europie taką sprzedażą zajmują się pewne kooperatywy, uzgodnienia pomiędzy rolnikami, może nawet stowarzyszenia.

Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przed chwilą poseł Konfederacji w płomiennym wystąpieniu krytykował zielony ład, który jest popierany przez wszystkie praktycznie związki zawodowe drobnych rolników w całej Europie.

Bardzo proszę, pan poseł Kazimierz Plocke, Koalicja Obywatelska. Mam dwa pytania do pana ministra. Pierwsze pytanie. W ustawie zapisaliśmy, że gospodarstwa rolne wytwarzające i wprowadzające żywność na rynek będą podlegały urzędowej kontroli ze strony inspekcji weterynaryjnej, inspekcji sanitarnej. Czy to oznacza, że małe gospodarstwa rolne będą podlegały takim samym procedurom jak firmy, przedsiębiorstwa wytwarzające żywność w sposób przemysłowy? Czy minister rolnictwa podejmie negocjacje z Ministerstwem Finansów w zakresie zmiany załącznika nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie określenia limitów produkcji?

Pan poseł Leszek Galemba, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Podważacie, jakbyście nie wiedzieli, że na każdym produkcie jest etykieta. Rolniczy handel detaliczny to przyszłość rolnictwa. Podważacie ilość powstałych podmiotów. To jest ok. 50 gospodarstw w powiecie, 330 powiatów razy 50 daje nam tę liczbę. Czyli rozwija się to wszystko. Panie Ministrze! Zwiększy się. Nie. Chcemy racjonalnie: z 40 tys. do 100 tys., a potem 2%. Każdy ma prawo sprzedawać, ile zechce. Surowce naprawdę pochodzą z tych gospodarstw rolnych. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica.

Wysoki Sejmie! Ta ustawa idzie we właściwym kierunku, zwłaszcza że jak sobie przypomnimy, 2 czy 3 tygodnie temu uchwalaliśmy ustawę, która mówi o tym, że samorządy będą miały obowiązek wyznaczenia miejsc handlu, m.in. handlu detalicznego dla rolników.

Czy jako element obrotu.

Dziękuję. Ostanie pytanie, pan poseł Romuald Ajchler. Wysoka Izbo! Lewica poprze projekt ustawy, bowiem uważamy, że nie możemy mówić już dzisiaj na wsi o tym, że jest drożyzna, tylko że wkradła się bieda i że rolnicy walczą z biedą. Cała komisja rolnictwa przyjęła projekt jednogłośnie. Lewica popiera każdą ustawę, która idzie w tym kierunku, że mianowicie próbuje zwiększyć dochody rolników.

Jak wy szacujecie, jakie ewentualnie dobrodziejstwa wynikające z tej ustawy popłyną na wieś? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana ministra Lecha Kołakowskiego.

Wysoka Izbo!

Państwo polskie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom.

Przechodzę do pytań.

Podwyższać kolejne progi będziemy mogli w następnych etapach, jeżeli będzie taka potrzeba. Pochylamy się nad tym problemem. Odnośnie do Komisji Europejskiej - wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Jest to przedmiotem drugiego czytania. System podatkowy jest zgodny z prawem. Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się, że zmiany podatkowe mogą być wprowadzane, jeżeli są korzystne dla rolników.

Ograniczenie procentowe ustanowione jest w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. I rolnicy korzystają z tej możliwości. Pan poseł Mirosław Maliszewski. Tak jak wcześniej wskazałem, kontrola jest to nadzór. Chodzi tu o kontrolę inspekcji. Chcę również dodać, że tu występują też elementy edukacyjne odnośnie do wsparcia z PROW, działania 4.2. A w ogóle chcę bardzo podziękować panu posłowi za deklarację poparcia tego dobrego projektu. Chcę powiedzieć, że kierować będziemy się polską racją stanu i dobrem polskiej wsi, producentów żywności. Tu chcę powiedzieć, że jest to kolejny krok w kierunku poprawy sytuacji ekonomicznej rolników. Pan poseł Piotr Borys.

W planie strategicznym jest to 200 tys. zł i to jest na wniosek. Jest to bardzo prosta procedura. Należy tylko złożyć wniosek do powiatowego lekarza weterynarii lub inspekcji sanitarnej. Prościej się nie da, ale bardzo dziękuję. Pan poseł Ryszard Wilczyński.

Chodzi o bezpieczeństwo żywności i obywateli. Tak że pewne kwestie muszą być uregulowane prawnie. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Tutaj chcę podkreślić szczególną rolę też ustawy wspierającej, o handlu w piątki i soboty. Jest to bardzo potrzebne i oczekiwane zadanie. Pan poseł Romuald Ajchler. Zakładano, że tym programem w roku 2017 objętych będzie 10 tys. rolników. Dzisiaj widzimy, że jest ich 14 tys., czyli jest ich o 40% więcej.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, druk nr 1837. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 1822 i 1837) Bardzo proszę pana posła Krzysztofa Lipca o przedstawienie sprawozdania komisji.

Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który został przedstawiony w druku nr 1822.

Projekt został uzasadniony przez posła, który reprezentował środowisko posłów, którzy przedłożyli ten projekt ustawy.

Muzeum nie posiadało osobowości prawnej, zostało powołane, jak wspomniałem, na zasadzie zarządzenia i funkcjonowało w ramach struktury organizacyjnej Służby Więziennej. Muzeum to jest zlokalizowane przy ul. Rakowieckiej 37, a więc każdy polski patriota wie, o czym mówimy w tej sprawie. To jest miejsce kaźni wielu pokoleń Polaków, którzy za to, że chcieli żyć dla Rzeczypospolitej i działali na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej, byli tam męczeni i katowani przede wszystkim w okresie stalinowskim przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ale również i w późniejszym okresie, aż do, można powiedzieć, roku 1990, kiedy to odzyskaliśmy jako państwo byt państwa niepodległego.

Rzecz dotyczy również jednego obiektu, natomiast te kwestie nie zostały, że tak powiem, zrealizowane z tego względu, że w czasie pandemii brakowało środków inwestycyjnych.

Wysoka Izbo!

To jest dobre rozstrzygnięcie i bardzo polecam, zachęcam, aby ponad podziałami politycznymi Wysoka Izba zechciała uchwalić ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dziękuję, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy pan poseł Dariusz Olszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od zakończenia II wojny światowej minęło już 76 lat, ale bardzo powoli przebija się do świadomości Polaków wiedza o tym, że po latach niemieckiej okupacji wkraczająca na polskie ziemie Armia Czerwona nie niosła Polsce i Polakom wolności i pokoju. Oddziały NKWD i Smiersz przynosiły ze sobą niewyobrażalne tortury i śmierć zadawane wszystkim niepokornym i nieposłusznym nowej komunistycznej władzy, wszystkim, którzy nie akceptowali siłą narzuconego ustroju.

Czyniono wszystko, aby w narodzie polskim osłabić tożsamość narodową, świadomość historyczną, patriotyzm i wiarę katolicką.

Wielu z nich przeszło niewyobrażalne tortury w więzieniach NKWD i aresztach śledczych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Obok tzw. Łączki na terenie Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach, więzienia Toledo na Pradze, więzienia w Rembertowie symbolem zniewolenia oraz terroru wobec żołnierzy i polskiego społeczeństwa jest przede wszystkim areszt śledczy na warszawskim Mokotowie. Pawilon X tego aresztu był miejscem niewyobrażalnych tortur, jakie spotkały polskich patriotów. Przez tego rodzaju miejsca utworzone na terenie całego kraju przeszły setki tysięcy ludzi, a dziesiątki tysięcy - straciły życie. Nie tylko dlatego, że nie zgadzali się oni na Polskę bolszewicką, ich jedyną winą było to, że chcieli Polski polskiej, rządzonej przez Polaków. Temat ten dopiero od początku lat 90. powoli zaczął docierać do świadomości Polaków. Ujawnienia prawdy o ofiarach domagają się ostatni żyjący wyklęci oraz rodziny poległych i pomordowanych. Poznanie prawdy historycznej jest szczególnie ważne dla prawidłowego ukształtowania postaw i charakterów młodego pokolenia dla zakorzenienia w nich miłości do ojczyzny i czci wobec obrońców polskości. Teren więzienia przy ul. Rakowieckiej, a zwłaszcza jego budynki, są niemymi świadkami wydarzeń tamtych lat. Ściana straceń z licznymi dziurami po kulach zmusza do zadumy i pamięci o ofiarach reżymu komunistycznego. Wraz z rodzinami żołnierzy wyklętych chciałbym w tym miejscu podziękować panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze za rozpoczęcie procesu upamiętniania żołnierzy wyklętych i za podjętą decyzję o przekształceniu więzienia mokotowskiego w państwową jednostkę muzealną poświęconą tak licznym ofiarom zbrodniczego reżymu. Dzięki tej odważnej inicjatywie dowody zbrodni komunistycznych i mordów sądowych zostaną zabezpieczone i wyeksponowane. Prawda historyczna będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym, a dowody licznych zbrodni zostaną zaprezentowane w świetle dziennym. Oczywiście zrozumiałe jest, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest już właściwym organem do prowadzenia placówki muzealnej, i najlepszym krokiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest kolejna decyzja, tym razem o przekazaniu muzeum żołnierzy wyklętych pod zarząd Instytutu Pamięci Narodowej. Pozwoli to na prawidłowy rozwój tej placówki, utrzymanie założonego jej charakteru oraz kontynuowanie badań historycznych i dokumentowanie prawdy historycznej. Muzeum powinno być miejscem ukazującym i dokumentującym tragedie i dramaty z szacunkiem i uznaniem dla cierpienia oraz zadumą nad poświęceniem uczestników walki o wolność i niezawisłość ojczyzny. Winno służyć refleksji nad dramatem minionego czasu, poznaniu nieznanych zdarzeń czy uzyskaniu wiadomości o losach bliskich. Dawać możliwość opowiedzenia czy udostępnienia ich losów szerszej publiczności oraz odnalezienia grobów i miejsc tajnych pochówków. Ważnym elementem jest także umożliwienie nawiązania kontaktów z towarzyszami walki i cierpienia. Muzeum powinno pokazywać, że Polska chce pamiętać o swoich bohaterach i wyjaśnić, dlaczego wyklęci byli wyklęci. Wysoki Sejmie! Klub PiS popiera ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i będzie głosował za przyjęciem ww. ustawy. Bardzo proszę, pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Witam pana ministra Kaletę, ale chciałbym przede wszystkim przywitać nieobecnego dzisiaj ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Piotra Glińskiego. Bo, Wysoka Izbo, wtedy kiedy rozmawiamy o muzeach, na sali posiedzeń powinien być minister kultury. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz na samym początku.

Ale ta debata nie jest o tym, czy tam powinno być muzeum, bo to sprawa oczywista. Pytanie jest dzisiaj zasadnicze: W jaki sposób powinno być zorganizowane, przez kogo powinno być prowadzone i czy projekty ustaw, które są przekazywane Wysokiej Izbie, powinny być przykładem niechlujstwa, bałaganu i niekompetencji? Bo tak trzeba po prostu, Wysoka Izbo, nazwać projekt poselski pisany na kolanie, złożony 2 grudnia przez grupę posłów, przede wszystkim Solidarnej Polski. Dzisiaj nieobecność ministra kultury na posiedzeniu połączonych komisji jest przykładem niepoważnego traktowania tego projektu i niepoważnego traktowania tego zagadnienia. O tym chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć. Szanowni Państwo! W zamyśle, jak rozumiem, wnioskodawców jest przekazanie tego muzeum Instytutowi Pamięci Narodowej. Ale zadajmy sobie podstawowe pytanie: Czy Instytut Pamięci Narodowej jest właściwą jednostką do prowadzenia muzeów w Rzeczypospolitej Polskiej? W mojej opinii nie. Jest ustawa o muzeach, jest ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. A pierwszą rzeczą, którą widzimy w tym projekcie, jest co? Jest wyłączenie stosowania tych ustaw, w szczególności jeśli chodzi o ustawę o muzeach, chcecie wykreślenia działania z art. 6 ust. 1, czyli tego, że statut muzeum jest uzgadniany z ministrem kultury. Chcecie wyrzucić art. 8 ustawy o muzeach, czyli nadzór ministra kultury nad tym muzeum. Chcecie, żeby minister kultury nie miał jakiegokolwiek wpływu na obsadzenie rady muzeum, która przy muzeum powstanie. Chcecie wyłączyć art. 23, który mówi o tym, że muzea państwowe i samorządowe mogą dokonywać zamiany, sprzedaży, darowizn muzealiów, czyli wpływać na podnoszenie wartości tej jednostki.

I chcecie wyłączyć udział ministra kultury przy ewentualnej likwidacji muzeum. Taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość. Nie ma na sali, szanowni państwo, również prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tak naprawdę w żaden sposób, w sposób oficjalny powołany przez Sejm i przez Senat prezes IPN w tej sprawie nie zabrał głosu, czyli tak naprawdę nieznane jest stanowisko instytucji w tej sprawie. Czy rzeczywiście w ciągu 30 dni od momentu ogłoszenia ustawy chciałby przejąć tę instytucję? Instytucję rozgrzebaną z niezakończonym procesem inwestycyjnym, z pięcioma decyzjami administracyjnymi, których termin ważności kończy się na początku przyszłego roku, czyli może innymi słowy część przepisów tej ustawy wejdzie z mocą wsteczną wtedy, kiedy decyzje dotyczące rozbudowy muzeum czy też rozbiórek nie będą już po prostu obowiązywać. Wysoka Izbo! Legislatorzy sejmowi na tym projekcie nie zostawili suchej nitki. To jest kolejna rzecz, którą należy podkreślić. Chciałbym zapytać, jaka jest rzeczywista chęć wspierania przez was pożytecznych, wartościowych inwestycji dotyczących patriotyzmu, dotyczących propagowania ważnych rzeczy z punktu widzenia historii. Bo mamy, szanowni państwo, Fundusz Patriotyczny - 30 mln zł. Ogłoszono, że to są środki na to, żeby pielęgnować pamięć o naszych bohaterach. Szanowni państwo, mamy „Cele bezpieki” w byłym resorcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - to jest obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy Wysoka Izba wie, z kim Muzeum Powstania Warszawskiego przegrało w konkursie o pieniądze z Funduszu Patriotycznego? Z Bąkiewiczem, ze Strażą Narodową, ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. Czy tak chcecie prowadzić sprawy dotyczące również tego muzeum?

Bardzo proszę, pani poseł Anna Maria Żukowska, Lewica. Pani Marszałek! Jako Lewica byliśmy przeciwko powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej. Złożyliśmy projekt ustawy o likwidacji tegoż instytutu, w związku z czym nie widzimy powodów, by dawać kolejne kompetencje temu instytutowi. Uważamy, że muzeami w Polsce powinno się zajmować ministerstwo kultury. Nie jest to instytucja, która powinna być w jakikolwiek sposób związana z bieżącą polityką, dlatego jesteśmy przeciwko tej ustawie i będziemy głosowali przeciwko. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Ona nie zawsze była tylko i wyłącznie patriotyczna. Bardzo żałuję, że ten projekt nie jest projektem rządowym, bo taki powinien być.

To jest resort powołany do tego, aby sprawował nadzór, opiekę nad muzeami w Polsce. Wiem, że to nie jest rozwiązanie, które funkcjonuje wszędzie, ale tak powinno być, a my, stanowiąc prawo, powinniśmy to prawo stanowić dobrze.

Rzeczą niedobrą jest to, że nie poznaliśmy nawet szacunkowych kosztów. Jeżeli mówimy o czymś, to powinniśmy wiedzieć, za ile zamierzamy coś zrealizować.

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni czy patrioci, ci, którzy walczyli z minionym systemem, byli w każdym z naszych obozów politycznych. Szkoda, że państwo tak bardzo mocno to zawłaszczacie i nie pozwalacie, żebyśmy pracowali nad tym wspólnie. Bardzo mnie smuci to, że pan minister kultury jest dzisiaj nieobecny, ale jest dzisiaj również niemy.

Mając to na względzie, szanowni państwo, nie wiem jeszcze, jaką rekomendację ostatecznie przekażę moim koleżankom i kolegom. Uważam, że idea jest słuszna, natomiast sposób wykonania niestety po raz kolejny jest słaby, mierny, a niektórzy mówią bardziej dosadnie.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Michał Urbaniak w imieniu koła Konfederacja. Zapraszam, panie pośle. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Prawdą jest też, że ta ustawa nie w pełni określa stosunek muzeum choćby do ministra kultury.

Stoi na straży historii naszego narodu, stoi na straży prawdy.

Trzeba pamiętać też o tym, że gdyby zmieniła się władza, IPN mógłby być bardziej niezależną instytucją niż minister kultury, bo w tym wypadku, jeśli zmieniłby się minister kultury, to w zasadzie z dnia na dzień mógłby zamknąć takie muzeum i nikt by nic pewnie z tym nie mógł zrobić.

Zatem mam wrażenie, że chodzi głównie o walkę polityczną, a nie o realne działanie na rzecz upamiętnienia bohaterów, którzy stracili życie m.in. przez zbrodniarzy PRL. Pan poseł Tomasz Zimoch w imieniu koła Polska 2050. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Po raz kolejny posiedzenie komisji pokazało, jak trudne jest obecnie sejmowanie. Nie są przyjmowane argumenty, głosy przeciwne odnośnie do niektórych propozycji są ignorowane, osoby mające prawo wyrażać własne poglądy są niestety obrażane, a uwagi sejmowych legislatorów są lekceważone i pomijane. Przy procedowaniu nad tym projektem nie ma sejmowej współpracy, a przecież powinno wszystkim zależeć, właśnie tu, w polskim parlamencie, na przywróceniu wspólnotowej pamięci o podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej. Właśnie w Sejmie, omawiając takie projekty ustaw, nie powinniśmy poszerzać budowanej od kilku lat propagandy historycznej. Rację mają ci historycy, którzy domagają się, by pamięć o podziemiu powojennym nie przesłaniała przecież działania Armii Krajowej czy późniejszych zrywów sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. Po dzisiejszym posiedzeniu komisji mam wrażenie, że rację mają też nauczyciele, mówiąc, że w programie szkolnym żołnierze wyklęci stają się centralnymi figurami polskiej historii XX w. Projekt przenosi Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w gestię Instytutu Pamięci Narodowej. W związku z tym jego prezesowi daje pełną władzę nad tą placówką. Przecież kierujący obecnie Instytutem Pamięci Narodowej, najdelikatniej mówiąc, nie radził sobie w Gdańsku z prowadzeniem Muzeum II Wojny Światowej, a IPN karnie wykonuje politykę historyczną. Koło Parlamentarne Polska 2050 będzie głosować przeciwko tej ustawie, bo naszym zdaniem rozszerza zakres kompetencji instytucji, do której nie tylko my nie mamy pełnego zaufania. Przechodzimy do pytań. Bardzo proszę.

Szanowny Panie Ministrze!

Czyżby nagle projektodawcy, zwracam się do wnioskodawców, uznali, że minister kultury i dziedzictwa narodowego - myślę że ten obszar jest elementem dziedzictwa narodowego - powinien być prowadzony właśnie przez ministra kultury, a nie przez Instytut Pamięci Narodowej? Dlatego też chciałbym zapytać, jakie są argumenty merytoryczne ze strony wnioskodawców, że przewidują powierzenie funkcjonowania tego szczególnego muzeum właśnie Instytutowi Pamięci Narodowej.

Dziękuję. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W tym wielkim sporze o kształt polityki historycznej Polski, która odzyskała niepodległość po sowieckiej okupacji, zwyciężył śp. Lech Kaczyński, a nie obściskujący się ze zbrodniarzem, mordercą i sowieckim kolaborantem Wojciechem Jaruzelskim Adam Michnik.

To muzeum powstaje. Dobrze, że znajdzie się w Instytucie Pamięci Narodowej, że tam zostanie zbudowane. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Projekt ten daje nadzieję, że IPN przez prawie 25 lat swojej działalności zdążył już rozliczyć wszystkie osoby, które dopuściły się czynów noszących znamiona przestępstwa, i powoli w miejsce prokuratorów zacznie zatrudniać muzealników oraz konserwatorów zabytków. Czy wraz z przekazaniem kompetencji nastąpiło przekazanie środków między Ministerstwem Sprawiedliwości a IPN-em? Czy może minister przekazał nadzór nad muzeum bez uszczuplania swojego budżetu, a na jego działalność przeznaczone zostaną nowe środki z budżetu państwa? Uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Panie Ministrze! W projekcie ustawy czytamy: Rada Ministrów w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy podejmie uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie” Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie” stanowi załącznik do niniejszej ustawy. Bardzo proszę o pisemną odpowiedź na pytanie, jakie środki zostaną przeznaczone na zacytowany przeze mnie program w poszczególnych latach. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Czy w związku z przejęciem muzeum wzrośnie budżet Instytutu Pamięci Narodowej i o jaką kwotę? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Posłowie! Poseł sprawozdawca apelował, żeby przyjąć tę ustawę ponad podziałami. To bardzo dobra idea i jestem za. Tylko że jeżeli chce się coś przyjmować ponad podziałami, to należy słuchać wszystkich. Jako żywo nie bardzo wiem dlaczego, ani nie było ministra kultury, ani nie było stanowiska ministerstwa kultury, ani nie było przedstawiciela ministerstwa kultury. Wszystkie nasze wnioski i apele o tym, żeby jednak poprosić o taką opinię i poczekać na nią, jak gdyby poszły w powietrze. Mam takie pytanie do wnioskodawców: Czy naprawdę najszczytniejszą ideę musicie spaprać? Bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego zgłaszacie projekt, w którym mówicie o muzeum, które muzeum nie jest?

Wysoka Izbo! Padły tutaj pytania: Dlaczego nie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Drodzy państwo, naprawdę tak.

Teraz najważniejsza kwestia, bo czas goni.

Wszyscy mogli to poznać. Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Ministrze Mejzo! Przy tworzeniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL chcę podkreślić: szacunek dla tych, którzy walczyli o wolność i za nią ginęli, ale pogarda dla tych, którzy pod tymi szczytnymi hasłami mordowali ludność cywilną, zajmowali się rozbojem lub antysemityzmem. Oprócz prawdziwych patriotów i bohaterów byli też bandyci. Pytam więc, czy w tym muzeum zamierzacie fałszować historię. Czy będzie tam sala Burego, który ponosi odpowiedzialność za szereg zbrodni wojennych? Z jego rozkazu rozstrzeliwano jeńców litewskich, ludność cywilną narodowości białoruskiej lub wyznania prawosławnego. Czy będzie sala Łupaszki, który oskarżany jest o to, że jego oddział dokonał masakry na litewskiej ludności cywilnej w Dubinkach? Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Jasne. Pani poseł, niech pani już przestanie się kompromitować, bo to, co przed chwilą usłyszeliśmy, to słowa haniebne. Nie przystoi posłowi Rzeczypospolitej Polskiej takich tekstów kłamliwych, obrażających bohaterów Rzeczypospolitej Polskiej wygłaszać. Panie Ministrze! Panie Prezesie! Czy prawdą jest, że Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest urzędem państwowym o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych, poszukiwawczych? Dzisiaj podczas obrad w komisji wspólnej: kultury i sprawiedliwości był obecny pan wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Jest również obecny teraz, mamy przyspieszenie obrad Sejmu, więc proszę nie kłamać, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest nieobecny. Bardzo serdecznie pragnę podziękować pani poseł Anicie Czerwińskiej za pomysł, aby takie muzeum powstało, Ministerstwu Sprawiedliwości za to, że tego dokonało i że Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL istnieje w naszym kraju.

Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Chciałbym zadać konkretne pytania. Czy były prowadzone rozmowy między ministrem sprawiedliwości a ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w kwestii ewentualnego przejęcia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL? Jeśli tak, prosimy o terminy, prosimy o ustalenia. Jeśli pan dzisiaj tego nie przekaże, będziemy wnioskować o dokumenty w tej sprawie. Kolejne pytanie: Czy w tej sprawie były prowadzone rozmowy z ministrem kultury?

Z punktu widzenia ustawy o muzeach, z punktu widzenia tego artykułu bardzo ważna jest możliwość, którą on kształtuje, dotycząca współpracy między muzeami i możliwość dokonywania zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów. Kolejna, ostatnia rzecz, pani marszałek: Jaki będzie związek między funkcjonującym Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce a docelowym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Nie wnikając w szczegóły tej ustawy, uważam, że wszystkich patriotów i organizacje, które w przeszłości tych patriotów gromadziły, powinniśmy traktować w sposób równy i sprawiedliwy.

Jeśli przywracamy dzisiaj to godne miejsce, to powinniśmy (Dzwonek) przywracać wszystkim. Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Nikt tutaj nie kwestionuje celowości powstania tego muzeum i tego, co powiedział poseł Szczerba, że rzeczywiście są to rzeczy święte dla wszystkich Polaków. Ale, po pierwsze, bardzo bym chciała, żeby historią zajmowali się historycy, a nie politycy. To bardzo nam ułatwi znalezienie porozumienia. Naprawdę nic by się nie stało, gdybyśmy mieli czas na porozmawianie z ministrem kultury, który może przedstawiłby nam swoją rację, gdybyśmy posłuchali, czy istnieje możliwość współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z ministrem kultury, co wydawałoby się zasadne, ponieważ instytut ma inne zadania, a zupełnie inaczej prowadzi się muzeum, to są także trochę inne cele. Wydaje mi się, że powodem jest to, że Ministerstwo Sprawiedliwości wie, że nie zdąży zrealizować tych wszystkich terminów i odrzuca to muzeum jak palący kartofel (Dzwonek), żeby nie brać za to odpowiedzialności. Dziękuję, pani marszałek. Pan poseł Dariusz Bąk, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Chwała Instytutowi Pamięci Narodowej za to, że wydobyła z ciemności prawdziwych bohaterów i przywraca właściwą pamięć Polakom. Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej wiemy, kto był bohaterem, a kto zdrajcą, wiemy, kto był ofiarą, a kto katem.

To muzeum pozwoli w sposób bardziej dogłębny poznać prawdziwą historię narodu polskiego, oświecić Polaków, żeby się uszlachetnili.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! To jest zupełnie niepotrzebne. Mam kilka pytań do pana, choć widzę, że pan rzeczywiście notuje dosyć wnikliwie, słuchając naszych wypowiedzi. Dlaczego nie zostały policzone - a jeśli zostały, to dlaczego nie zostały nam przedstawione - koszty powstania muzeum albo przekazania tego muzeum, tak to nazwijmy, do IPN-u? Czy bierze pan pod uwagę, że wszelkie sprawy związane z tą inwestycją w przyszłości będą - albo inaczej: powinny być - regulowane już tylko ustawami? Jeszcze jedno pytanie: Gdyby pan był ministrem kultury, to czy dzisiaj nie poczułby się pan trochę dotknięty tym, że to nie właśnie panu oddano władzę nad tym muzeum?

Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To muzeum to muzeum jeszcze niezabliźnionych ran - ran, które na tkance narodu polskiego jeszcze nie zdążyły się zabliźnić, bo jeszcze żyją bliscy tych, którzy byli tam mordowani. Konieczna jest pamięć o tych ludziach, którzy ponieśli śmierć lub doznali cierpień za to, że chcieli wolnej Polski, chcieli żyć w normalnej ojczyźnie.

że powstał pomysł przeniesienia własności tego muzeum do Instytutu Pamięci Narodowej, bo tam jest jego miejsce. O udzielenie odpowiedzi na pytania pań i panów posłów uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Sebastiana Kaletę. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ponieważ żyli prawem wilka/ historia o nich głucho milczy”, „nie opłakała ich Elektra/ nie pogrzebała Antygona/ i będą tak przez całą wieczność/ w głębokim śniegu wiecznie konać” W ten sposób o dramacie żołnierzy wyklętych w wierszu „Wilki” pisał Zbigniew Herbert. W Polsce już wolnej dosyć długo trwa spowodowanie, by historia przestała w pełni pisać o tym, co Herbert określił jako głuche milczenie. Żołnierze wyklęci nie porzucili nie tylko swojej miłości do ojczyzny, kiedy zakończyła się II wojna światowa, ale nie porzucili także broni. Nie porzucili z tego powodu, że m.in. mieli świadomość tego, że jeśli to zrobią, mogą zostać zamordowani. Tak w istocie się działo. To właśnie robili komuniści w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie - strzałem w tył głowy. Dziś, po dziesiątkach lat, udało się nawet znaleźć ślady po kulach na murach więzienia. W tej właśnie sprawie spotykamy się dziś w Sejmie, by historia przestała głucho milczeć o swoich bohaterach i by pokryte tynkiem dziury po kulach odkryć i pokazać lekcje historii, pokazać historię opresji i terroru, historię walki i zniewolenia, historię marzeń, które przez krew i pot znalazły swoją ścieżkę ku wolności. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL działa od 2016 r. Decyzją ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przystąpiono do zamknięcia funkcjonującego aresztu i podjęcia działań, by ten betonowy pomnik ociekający krwią polskich bohaterów był miejscem hołdu dla ich poświęcenia. Przeprowadzono konkursy architektoniczne, uzyskano pozwolenia na budowę.

Jest to miejsce wyjątkowe w skali Polski i Europy. W celach tych komuna trzymała Jacka Kuronia, Antoniego Macierewicza, Andrzeja Czumę, Karola Modzelewskiego, Jana Lityńskiego i setki, tysiące innych opozycjonistów czasów PRL. To muzeum nie obejmuje swoją pamięcią wyłącznie żołnierzy wyklętych, szanowni państwo, Wysoki Sejmie, to muzeum opowie o zmaganiach milionów Polaków, by komunę odrzucić również po okresie stalinowskim. To będzie pierwsze i wyjątkowe miejsce w Polsce, które w całości opowie tę dramatyczną walkę Polaków o wolność. Te mury nie rozróżniały barw politycznych i historia wszystkich tych osób jest i będzie opowiadana w tym muzeum. Historia dziś może przestać głucho milczeć.

Wiele pytań dotyczyło dotychczasowego funkcjonowania muzeum. Mam nadzieję, że poprzez przekazanie tych informacji przekonam państwa i państwa kluby, byśmy wspólnie tę ustawę przyjęli, i że uznają państwo wyjaśnienia, które przedstawię, za wystarczające, byście państwo z nami wspólnie poparli tę ustawę, byśmy wspólnie wysłali taki sygnał, jaki wysyłali więzieni tam Polacy. Tam wszyscy byli równi, wszyscy chcieli wolnej Polski. Mam nadzieję, że w tej Izbie również. Zatem przechodzę do szczegółów podnoszonych w pytaniach. To wyłączenie wynika z faktu, że IPN jest instytucją państwową, ale niezależną od rządu. Ta ustawa zakłada zachowanie tej zasady. Obawiam się, że gdyby tych przepisów nie było, państwo moglibyście podnieść zarzut, że właśnie dochodzi do zwiększenia wpływu rządu na funkcjonowanie IPN-u.

Pani marszałek Kidawa-Błońska powiedziała, że tą sprawą powinni się zajmować historycy, a nie politycy.

Dlaczego? Ponieważ od pierwszego dnia funkcjonowania muzeum to historycy IPN byli wiodącymi postaciami w pracach badawczych, w przygotowywaniu wystaw tymczasowych czy też różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych, które muzeum cały czas organizuje. To historycy IPN są w gremiach decyzyjnych, które podejmowały decyzje o projektach, o koncepcjach.

Pan prof. Krzysztof Szwagrzyk przeprowadził ze swoim zespołem szereg prac badawczych, odkryto, ekshumowano szczątki osób, które były tam mordowane w różnych okresach, również w czasach okupacji niemieckiej. Dzięki tej placówce działalność IPN z pewnością się rozwinie.

Tak, od 5 lat w tej sprawie rozmawiamy.

Również ta komórka przeprowadziła konkursy, o których mówiłem. Również ta komórka przeprowadziła proces pozyskania pozwoleń na budowę.

Dzisiaj to się, można powiedzieć, krystalizuje z tego powodu, że jesteśmy w kluczowym momencie, momencie, w którym wszystko, co trzeba było zrobić przed przetargiem, jest wykonane. Jest odebrana dokumentacja, są pozwolenia, jest jasna koncepcja, jest już kilkanaście tysięcy eksponatów zgromadzonych przez muzeum. Teraz trzeba po prostu zrewitalizować budynek i zorganizować wystawę, a w związku z tym - ustalić finansowanie. Padały pytania o koszty. Dokumentacja jest już znana w przeciwieństwie do ustawy, którą państwo przywołaliście. Tutaj nie rozmawiamy o, można powiedzieć, szacunkach, ale już o pewnych konkretach wynikających z projektów budowlanych, które są odebrane. Powiem, jakie są to kwoty.

Jest to plan realizacji wieloetapowej inwestycji z różnymi etapami oddawania również do użytku, jeśli będzie taka możliwość, wystaw, bo jest tu kilka budynków. Oczywiście jeśli chodzi o etapowanie tej inwestycji i czas realizacji, to również tutaj Rada Ministrów będzie się nad tym w niedługim czasie pochylała.

Wbrew niektórym opiniom czy głosom, które były dzisiaj przedstawiane, to nie jest utworzenie, to jest przekazanie czegoś, co działa, czegoś, co ma już swój dorobek, podstawy i filary, łącznie z prawem do nieruchomości. Wstęp do tego muzeum mają tylko zorganizowane grupy, natomiast od kilku lat są tam organizowane najważniejsze uroczystości państwowe związane z kluczowymi rocznicami, wokół których, można powiedzieć, skupia się praca muzeum: 1 marca i 13 grudnia.

Czy to nie jest taki symbol, na którym powinno nam dzisiaj zależeć? Te uroczystości są organizowane konsekwentnie.

Pojawiło się pytanie, dlaczego pilnie.

Gdyby tej ustawy nie było, być może ta inwestycja mogłaby dopiero wystartować pomimo tak dalekich wysiłków i tak dalekich punktów, które osiągnęliśmy, z opóźnieniem, czego nie chcemy. Na koniec, jeśli mógłbym poprosić.

Rzeczywiście pytania były personalnie kierowane do pana prezesa, zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania pań i panów posłów.

Szanowna Pani Marszałek!

Otóż dzisiaj wręcza w Lublinie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji demokratycznej Krzyże Wolności i Solidarności. Przepraszamy. Odnosząc się do tego, o czym państwo wspomnieli, chciałbym na wstępie zacytować fragment preambuły, która została uchwalona w tej sali 23 lata temu, za 4 dni będą 23 lata: Mając na względzie czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w obronie wolności oraz godności ludzkiej ustawa reguluje.

W 2006 r. decyzją Wysokiej Izby doszedł pion lustracyjny, a w 2016 r. - pion upamiętnień walk i męczeństwa.

Chciałbym podziękować za to zaufanie wobec władz Instytutu Pamięci Narodowej. To jest tak, że my, szanowni państwo, akurat tą działką, tą historią, zajmujemy się od samego początku i temat żołnierzy wyklętych, więźniów politycznych leżał u podstaw powstania Instytutu Pamięci Narodowej.

To dowód na to, że Instytut Pamięci Narodowej umie i potrafi sobie radzić także z zadaniami, które dotyczą muzealnictwa.

Padły pytania, jeśli chodzi o kwestię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy były jakieś formalne rozmowy między Instytutem Pamięci Narodowej a ministerstwem kultury.

Jest ono rzeczywiście szczególne w historii Polski.

Chodzi tu o nazwiska, które są podręcznikowe, a także o nazwiska, które dzisiaj współtworzą naszą demokrację, czy to patrzymy na prawą stronę, czy to patrzymy na inną część sali. Także z tej strony - tutaj patrzę na Platformę Obywatelską - jest bardzo wiele osób, które były tam więzione, a które współtworzą państwa formację. Zresztą dotychczasowe doświadczenia obecnego kierownictwa też wskazują, że nie jest tak źle, jeśli chodzi.

A więc może jak troszeczkę czasu minie, zobaczycie państwo, że nie będzie to w żadnym sensie muzeum polityczne.

Natomiast odpowiadając jeszcze szczegółowo na pytanie posła z Polskiego Stronnictwa Ludowego pana Krzysztofa Paszyka powiem tylko, że jeśli chodzi o Bataliony Chłopskie, to nie jest to temat zapomniany, bo jest on poruszany w otwartym niedawno też przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Tak że jest tych inicjatyw bardzo dużo, a jeśli państwo mają jeszcze jakieś inne pomysły, ale też zarzuty, to pan prezes dr Karol Nawrocki naprawdę jest osobą otwartą, nie zważającą nawet na ataki. Myślę, że mogę w jego imieniu powiedzieć, że nie tylko chętnie się z państwem spotka przy okazji corocznych sprawozdań z działalności i składania wniosków o środki budżetowe, ale także zaprasza do swojego gabinetu wszystkich, od prawej do lewej strony. Dziękuję bardzo, panie prezesie. O głos prosił również sprawozdawca komisji pan poseł Krzysztof Lipiec.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dla porządku rzeczy chciałem tylko wyjaśnić jedną kwestię, albowiem tak samo na posiedzeniu połączonych komisji, jak i dzisiaj, podczas tej debaty był czyniony zarzut, że nie jest obecny minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W toku prac legislacyjnych nad projektem tej ustawy rząd delegował ministra sprawiedliwości, którego reprezentował dzisiaj sekretarz stanu pan Sebastian Kaleta.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1835 i 1836) Uprzejmie proszę pana posła Piotra Króla o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1835. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury będzie miało nr 1836.

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 9 grudnia 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania. Chciałbym powiedzieć, że podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęto osiem poprawek, a odrzucono sześć poprawek. Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu tego pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu ustawy oraz rozpatrzeniu poprawek wnosi, by Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Anna Milczanowska. Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w zakresie złożonego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1835. Celem projektu ustawy jest transpozycja do polskiego systemu prawnego przyjętej, funkcjonującej w europejskim prawodawstwie dyrektywy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I. Wedle założeń unijnego prawodawcy przyjęty pakiet ma na celu tworzenie bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego. Ponadto celem dyrektywy jest zapewnienie równowagi pomiędzy poprawą warunków socjalnych i warunków pracy kierowców a zwiększeniem swobody świadczenia usług transportu drogowego w oparciu o uczciwą konkurencję między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami, co w konsekwencji ma przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej. W projekcie zaproponowano także niezbędne zmiany w dotychczas istniejących przepisach, mające na uwadze potrzebę wyeliminowania niejasności oraz poprawy czytelności norm prawnych sprawiających trudności w interpretacji. Należy wskazać, iż regulacja kwestii transportu drogowego, transportu ciężkiego na terenie Unii Europejskiej z uwagi na zastrzeżenia Polski co do przyjętych rozwiązań jest przedmiotem licznych działań polskiego rządu przeciwdziałających utracie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z branży transportowej. Warte podkreślenia jest również otwarcie Ministerstwa Infrastruktury z przebywającym z nami tutaj, na sali panem ministrem Rafałem Weberem na dialog z przedsiębiorcami zajmującymi się transportem drogowym.

Z uwagi na konieczność przystosowania polskiego prawa do prawomocnych regulacji Pakietu Mobilności I klub Prawa i Sprawiedliwości popiera proponowany projekt ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Paweł Papke. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Druk nr 1835 to projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z motywem dyrektywy zmierza ona do utworzenia bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego. Ponadto celem dyrektywy jest zapewnienie równowagi między poprawą warunków socjalnych i warunków pracy kierowców a zwiększeniem swobody świadczenia usług transportu drogowego w oparciu o uczciwą konkurencję między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami, co w konsekwencji powinno przyczynić się do poprawnego funkcjonowania rynku transportu drogowego w całej Unii Europejskiej. Projektowana ustawa wprowadza także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Niestety należy zwrócić uwagę na opieszałość rządu i implementację powyższej dyrektywy w ostatniej chwili. Utrudni to przedsiębiorcom z branży transportowej właściwe przygotowanie się do nowego prawa. Należy jeszcze zwrócić uwagę na porażkę rządu w negocjacjach z Unią Europejską, aby jak najlepiej zabezpieczyć polskie firmy transportowe. Niestety w czasie szalejącej w Polsce inflacji, drożejącego paliwa i pandemii COVID-19 firmy stracą rentowność, co może grozić upadłościami i stratami miejsc pracy. Zapewne przewoźnicy przerzucą koszty działalności na swoich kooperantów. Na końcu oczywiście jest ostatnie ogniwo, czyli konsument. Posłowie wraz ze środowiskiem transportowym na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Infrastruktury zaproponowali sześć bardzo ważnych poprawek, które znacząco ułatwiłyby przetrwanie i zapewniły konkurencyjność finansową polskich firm transportowych. Niestety, wszystkie te poprawki zostały odrzucone. Padła na szczęście deklaracja ze strony rządowej, z ust pana ministra Webera, że w czasie prac w Senacie rząd ze stroną społeczną i Senatem wróci do nich i po ich dokładnym przeanalizowaniu, przemyśleniu, przyjmie je. 288 stron to taka gruba książka. Parlamentarzyści mieli tylko kilkadziesiąt godzin, żeby zapoznać się z tym projektem i go zaopiniować. Chyba nie tak powinna wyglądać praca w Sejmie. Na podstawie powyższego Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska warunkowo poprze proponowaną nowelizację ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1835. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu klubu Lewica głos zabierze pan poseł Maciej Kopiec. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy wobec ustawy z druku nr 1835. Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. pakiet mobilności.

Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy. Wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

Wprowadzone zmiany przede wszystkim poprawiają sytuację finansową kierowców, natomiast będą generować dodatkowe koszty dla przedsiębiorców. Przedstawiciele branży zwracali w trakcie trwania posiedzenia Komisji Infrastruktury uwagę, że należy jak najszybciej wprowadzić nieuniknione zmiany legislacyjne, aby przedsiębiorcy mogli przygotować się do czekających ich zmian oraz faktycznie wdrożyć w życie nowe rozwiązania, co bezpośrednio związane będzie z dostosowaniem umów o pracę z kierowcami. Ministerstwo twierdzi, że wprowadzone zmiany mają również na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego. Branża transportowa jest świadoma, że wprowadzenie Pakietu Mobilności I jest nieuniknione, jednak, jak zwracaliśmy uwagę w trakcie posiedzenia komisji wspólnie z posłem Mirosławem Suchoniem z Polski 2050, prosimy o poparcie poprawki mającej na celu okrojenie do tylko niezbędnych kar w nowym taryfikatorze. Wprowadzone zmiany nie powinny wykraczać poza implementację prawa Unii Europejskiej i nadmiernie obciążać przedsiębiorców. Pakiet Mobilności I to jedno z największych wyzwań dla branży transportowej w ostatnim czasie. tego, że Ministerstwo Infrastruktury dopiero teraz rozpoczęło szczegółowe prace nad tym projektem w Sejmie, przedstawiciele branży, mając świadomość rewolucyjnego poziomu wprowadzanych zmian, już w grudniu ub.r. zwracali się do ministerstwa o jak najszybsze rozpoczęcie prac legislacyjnych, aby był czas na spokojną dyskusję i analizę wszystkich kontrowersji. Szkoda, że tak długo trwały prace legislacyjne nad tym projektem. Ubolewam, że z większą uwagą nie mogliśmy przeanalizować wszystkich zapisów zawartych w projekcie przedstawionym przez ministerstwo. Pan minister na posiedzeniu komisji raczył przyznać, że projekt nie jest dopracowany, a ministerstwo chce go jeszcze poprawić w Senacie, co deprecjonuje powagę Komisji Infrastruktury.

Tutaj pojawia się pytanie do pana ministra: Czy rozważaliście państwo zwiększenie poziomu finansowania inspekcji transportu drogowego? Należy pamiętać, że branża transportowa jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki. Jeżeli chcemy funkcjonować na rynku europejskim, zachowując konkurencyjność, powinnyśmy jak najszybciej i w jak najbardziej transparentny sposób wdrożyć unijną dyrektywę, nie pozostawiając miejsca na dwuznaczności w kwestii interpretacji. Klub Lewicy wspiera poprawki opozycji i poprze projekt ustawy.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści wobec sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1835.

W sierpniu 2020 r. wprowadzono pierwsze zmiany dotyczące przepisów Pakietu Mobilności. Kierowca powinien wrócić do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

Pojawiła się możliwość odbywania dwóch z rzędu skróconych odpoczynków tygodniowych w transporcie międzynarodowym, trzeba jednak spełnić szereg warunków.

Postój ten ma odbywać się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. Wyrównanie do wysokości pensji minimalnej nie będzie obowiązywało w przypadku tranzytu oraz transportu bilateralnego w zakresie dwóch dodatkowych operacji: załadunku i rozładunku. Zmian jest sporo. Przepisy nakładają od 20 maja 2022 r. na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. A zatem zmian jest dosyć dużo i dotkną one w znacznej części przedsiębiorców transportowych, którzy zapowiadają, że wskutek podwyższenia wynagrodzeń kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy koszt tych wynagrodzeń może wzrosnąć nawet o 100%, co spowoduje, że krajowe firmy staną się mało atrakcyjne na rynku.

Zastosowanie się do nowych przepisów spowoduje wzrost kosztów ponoszonych przez firmy transportowe. W celu uniknięcia strat firmy transportowe z pewnością będą podnosiły ceny, a co z tym się wiąże, ceny wzrosną, koszty usług wzrosną, więc różnice te pokryjemy my jako konsumenci końcowi.

Wysoka Izbo! Polska była liderem transportu drogowego w Europie. Byliśmy liderem w zakresie kabotażu we Francji, w Niemczech i Unia Europejska chciała to ograniczyć. Nie jest to dziwne.

Czy to jest poważne traktowanie Sejmu i legislacji w Polsce? To jest naprawdę niepoważne traktowanie tego wszystkiego.

Kto za to zapłaci?

Zamknie im to możliwość rozwoju taborów, zamknie im to możliwość wprowadzenia podwyżek dla pracowników, w związku z czym pewnie część pracowników przeniesie się za granicę, a może nawet i całe firmy się przeniosą. Implementacja tego prawa oznacza w dużej mierze upadek polskiego transportu drogowego za granicą. Dlatego jako Konfederacja składamy wniosek o odrzucenie w całości tego rządowego projektu. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Wysoka Izbo!

Jednak nie mogę się oprzeć refleksji, że to jest za późno, że jednak prace można było rozpocząć wcześniej.

Niemniej jednak dzisiaj należy podejmować decyzje, ponieważ jesteśmy u progu wejścia w życie przepisów. Kiedy te prace ruszyły, to pierwszy projekt przypominał granat. Ten granat, gdyby rzeczywiście dotrwał do dnia dzisiejszego, z pewnością wysadziłby w powietrze całą branżę transportową i pewnie trzeba by było wrócić do jakiegoś transportu konnego, bo w takich warunkach, jakie były pierwotnie w projekcie, z pewnością branża nie dałaby rady. Nie możemy uciekać od skutków gospodarczych. Efektem Pakietu Mobilności niestety jest pogorszenie warunków działania polskich firm i za to winę ponosi rząd. Jest to bezpośrednia wina rządu, który zamiast zajmować się dbaniem o interesy gospodarcze, tak jak robią to Francuzi, Niemcy, uwikłał się w bezsensowną i przegraną wojnę polityczną dotyczącą kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj ministerstwo i rząd oburzają się, że Niemcy, Francuzi walczą o swoje. Ale wymagamy od rządu - walczcie o polskie firmy, walczcie o polską gospodarkę, a nie politykujcie, bo od tego naprawdę są inne miejsca. Tak jak powiedziałem, ten projekt ewoluował, więc tutaj pana ministra docenię, że wyszedł naprzeciw wielu oczekiwaniom branży transportowej, ale do załatwienia pozostało co najmniej sześć spraw, które uzgodniła cała branża, i przedstawiła w jednolitym stanowisku.

Drugie czytanie, panie ministrze, to jest ten moment, w którym trzeba podjąć męską decyzję, wesprzeć polską branżę transportową i przyjąć poprawki branży transportowej, które niniejszym na ręce pani marszałek pozwalam sobie złożyć. Zamykam listę osób chcących zadać pytanie. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Andrzej Szewiński, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Podczas konsultacji społecznych padły argumenty, iż wprowadzenie w życie przedmiotowego projektu spowoduje, iż diety i ryczałty kierowców w firmach transportowych będą traktowane jako element wynagrodzenia i będą podlegały opodatkowaniu i dodatkowym opłatom na poczet składek na ubezpieczenie społeczne. Efektem takich zmian dla kierowców nieobjętych delegowaniem w międzynarodowym transporcie będzie średni wzrost kosztów pracy o ponad 17%. Dla kierowców delegowanych w transporcie międzynarodowym będzie jeszcze wyższy wzrost kosztów, co wpłynie na obniżenie konkurencyjności polskich firm przewozowych. Szanowny Panie Ministrze! Czy można wprowadzić w życie przepisy dostosowujące polskie prawo do unijnych regulacji, tak aby polscy przedsiębiorcy nie byli poszkodowani? Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Celem tej zmiany ustawy o transporcie drogowym jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

Jednym z podmiotów, który będzie realizował część kontrolną rozwiązań prawnych zawartych w ustawie jest Inspekcja Transportu Drogowego, a również jej oddziały wojewódzkie. Są też zadania dla samorządów. Ustawa przewiduje dodatkowe środki finansowe właśnie dla inspekcji i dla jej oddziałów ze względu na zwiększone zatrudnienie. Chciałbym zapytać, jakie nowe zadania będzie realizował w związku z tym samorząd powiatowy i gdzie są zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań prowadzonych przez samorząd powiatowy?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wprowadzenie do porządku obrad tego punktu kilka godzin po przedłożeniu Sejmowi 500 stron ustawy świadczy o niepoważnym traktowaniu posłów. Co gorsze, świadczy również o niepoważnym traktowaniu całej branży transportowej. Rząd miał prawie 2 lata na przygotowanie stosownych przepisów oraz na wprowadzenie ich w życie. Zamiast tego rząd zajmował się walkami o stołki, tworzeniem nowych ministerstw i obsadzaniem nowych ministrów Mejzów na tych stanowiskach. Ustawa zmienia znacząco warunki funkcjonowania podmiotów związanych z transportem i to powinno być przedmiotem obrad i przedmiotem analiz Wysokiej Izby.

Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych ustaw - oczywiście z zaskoczenia, wczoraj, po półtorarocznej pewnie ciężkiej pracy ministerstwa.

Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Otóż w wielu innych państwach branża transportowa otrzymuje wsparcie dla swojej działalności. To wsparcie jest związane choćby z możliwością pewnych dotacji do taboru, odnowienia taboru, pewnych dotacji związanych z ograniczaniem emisyjności oraz tworzeniem nowych rozwiązań, które można finansować w ramach dostępnych środków finansowych.

Czy będzie wsparcie dla branży transportowej? Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nareszcie zrobiliście coś, żeby uporządkować kilka drogowych patologii, o których mówimy od dawna. Polscy kierowcy traktowani są jak woły pociągowe, których jedynym celem jest przewożenie jak największej ilości towarów w jak najkrótszym czasie za jak najniższą cenę. W końcu zwróciliście uwagę na problem przerw w pracy. Kierowcy komunikacji miejskiej przez cały dzień jeździli praktycznie bez odpoczynku - czy służbowych delegacji, i to przez przepisy, które służymy temu, by kierowcom międzynarodowym płacić jak najmniej. Dzięki tej ustawie sytuacja zawodowa grupy liczącej kilka tysięcy osób stanie się lepsza, dlatego ją popieram. Ale to tylko jedna strona medalu. W budżetówce od wielu miesięcy trwają protesty, m.in. pracowników cywilnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego czy Państwowej Inspekcji Pracy, a więc osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo na drogach. Kiedy to zauważycie? Kiedy zaczniecie cenić ich pracę? Pan poseł Jerzy Paul, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że transport drogowy jest ważną częścią polskiej gospodarki. Polskie firmy transportowe przebojem podbijały zachodnie rynki swoją sumiennością, dotrzymywaniem terminów i dobrym taborem samochodowym. Sukcesy polskich kierowców na rynku europejskim stały się solą w oku zachodniego kosztownego transportu kołowego. Niestety dzisiejsze propozycje zmian w ustawie są w większości wymuszone przez Unię Europejską, która na siłę chce obarczyć polskich kierowców dodatkowymi wymogami, ograniczeniami i kosztami, co niestety ma z powrotem przynieść większą konkurencyjność francuskim czy niemieckim firmom transportowym. W imieniu swoim, ale i kierowców pragnę podziękować za dziesiątki spotkań z przedstawicielami firm transportowych, dzięki którym udało się wypracować ustawy możliwie najmniej dotykające branże polskiego transportu kołowego, a zarazem polskich kierowców. Panie Ministrze! W związku z dzisiejszymi propozycjami zmiany ustawy mam (Dzwonek) pytanie: Którzy polscy europarlamentarzyści w Unii Europejskiej bronili polskiego transportu drogowego, a którzy milczeli i los polskich kierowców był im obojętny? Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, koło Konfederacja.

Jak już w Unii Europejskiej odegraliście państwo teatralny sprzeciw wobec tych regulacji, to teraz przykładnie je wdrażacie.

Widzę, że skusiło jednak i wolimy łupić swoich kierowców, niż ich bronić przez durnymi regulacjami z Unii Europejskiej. Dlaczego? Pan poseł Krystian Kamiński, Konfederacja.

Wysoka Izbo!

Czemu łupicie polskie firmy, żeby potem 370 mln zł reinwestować w to, żeby jeszcze im kary dowalać? Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Polskie firmy transportowe rządzą na rynku Unii Europejskiej. Swoją przewagę zbudowały na solidności, inwestycjach w sprzęt i niższych niż na zachodzie Europy wynagrodzeniach. Dziś transport wypracowuje aż 7% polskiego PKB i daje pracę 700 tys. osób. Procedowana ustawa, choć dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych tworzących tzw. Pakiet Mobilności I i dotyczy zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, uznając ich za pracowników delegowanych, to w ocenie samych zainteresowanych stanowi realną groźbę likwidacji tysięcy miejsc prac w transporcie. Pytanie zasadnicze brzmi: Co rząd zrobił, jakie środki dyplomatyczne przedsięwzięto, aby ochronić interesy (Dzwonek) polskich firm transportowych na forum unijnym w tej materii? Pan poseł Marek Dyduch, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Dzisiaj w Europie jednym z najlepszych, najbardziej poszukiwanych towarów jest praca i wykwalifikowani pracownicy. Transport jest kluczem do obsługi gospodarki, do dostaw towarów. Widzimy po Wielkiej Brytanii, że wszystko się mogło załamać na skutek niedoceniania transportu - i kooperacja, i różne inne kwestie związane np. z obrotem towarowym. A więc jest to bardzo ważna dziedzina życia publicznego, gospodarczego. Chciałem zapytać, patrząc na ogromną konkurencję, która jest w Europie: Ilu polskich kierowców szacunkowo może pracować w innych firmach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii? I drugie pytanie: Co może zagrozić polskim firmom transportowym, jeżeli chodzi o konkurencję, utrzymanie się na rynku europejskim? Pan poseł Paweł Papke, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, to ok. 300 stron. A polski parlament miał kilkadziesiąt godzin, żeby zapoznać się z powyższymi propozycjami regulacji, z opiniami i z innymi dokumentami, które mają świadczyć o tym, że ta ustawa jest niezbędna. Pan jest też parlamentarzystą. Stąd wynika pytanie: Dlaczego tak długo trwały konsultacje społeczne z branżą transportową i dlaczego prace rządowe nad tym projektem tak długo trwały, że mamy tu, w parlamencie, tak mało czasu, aby zdążyć przed 2 lutego 2022 r. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zajmujemy się dziś tą ustawą, dlatego że wdrażamy rezultat prac w Unii Europejskiej nad Pakietem Mobilności. Ale w pracach nad tym pakietem polski rząd doznał klęski i dziś powinniśmy zastanawiać się, jak branżę transportu drogowego objąć tarczą. Jakie pomysły ma w tym zakresie rząd, żeby poprawić sytuację przedstawicieli branży transportowej? Ta branża to potęga w Europie. Dziś możemy tak jeszcze powiedzieć. Ale jak będzie po lutym, gdy te przepisy wejdą w życie? Wszyscy zadają sobie to pytanie, a pan minister musi na to pytanie odpowiedzieć. Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Odnoszę wrażenie, że to nie jest Pakiet Mobilności, tylko braku mobilności, skoro kierowcy są delegowani do danego kraju, że tak powiem, na stałe i tam zarabiają. Ale mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy sporów, które istnieją w tym zakresie. Te sprawy były nieuregulowane i bardzo często do biura zgłaszają się przede wszystkim właściciele niewielkich firm, którzy mają spory z kierowcami. Czy to rozwiązanie wpłynie na rozwiązanie tych sporów?

Zapraszam. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pani marszałek, nie myślałem, że kiedykolwiek zgodzę się z panem posłem Franciszkiem Sterczewskim. Tak, zgadzam się, są przypadki nadużyć, wykorzystywania polskich kierowców przez polskich przewoźników. Przecież tutaj, w Warszawie, mieście stołecznym rządzonym przez wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, mamy przypadki grubych nadużyć, tragedii związanych właśnie z nieprawidłowym naliczaniem godzin pracy przez kierowców. Dlatego dobrze, że w końcu te zapisy ustawy regulują i porządkują zasady zatrudnienia kierowców. Panie ministrze, czy omawiany projekt wprowadza zasady wynagradzania kierowców wykonujących transport międzynarodowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, pod warunkiem że uzna się ich za pracowników delegowanych? Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Ale dzisiaj pół dnia trwała debata budżetowa.

Czy takie środki, i w jakiej wysokości, pójdą w ślad za uchwaleniem tej ustawy? To z pewnością będzie miało miejsce. Taka konkluzja po wysłuchaniu debaty budżetowej i obecnej dyskusji: jeśli jest tak dobrze i ma być tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Rwą włosy z głowy, że będzie tragicznie, że będą plajty. Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy zapytałem o tempo, pan minister w sposób nawet niegrzeczny odpowiedział mi na posiedzeniu komisji. Pamiętamy niedawną dyskusję na temat likwidacji opłat na bramkach, wprowadzania e-TOLL, możliwości zakupu biletów, e-biletów, papierowych biletów. Dziś, po 2 tygodniach funkcjonowania, widzimy, jak to działa. Wystarczy wejść na portale, wystarczy obejrzeć filmy na portalach społecznościowych o tym, co dzisiaj kierowcy sądzą o waszych rozwiązaniach. Bubel pogania bubel, za co zapłacą ostatecznie kierowcy, bo nie mogą kupić biletów, bo bilety papierowe nie są dostępne, a na koniec dostaną odpowiednie wezwanie i zapłacą 400 czy 500 zł.

Panie Ministrze!

Z iloma podmiotami był konsultowany ten projekt ustawy? Chodzi mi o podmioty, przedsiębiorców transportowych, ale także o stronę społeczną. Ile ich opinii zostało zaakceptowanych przez rząd? Uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Rafała Webera o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Wysoka Izbo! Rozpocznę może od wniosku, który został złożony, który polega na odrzuceniu tego projektu w drugim czytaniu, bo nic bardziej szkodliwego państwo nie mogą wymyślić. Nic bardziej się nie wpisuje w scenariusz niemiecki czy francuski jak właśnie taka propozycja. Bo właśnie o to chodzi, żeby od 2 lutego w Polsce nic się nie zmieniło, aby Pakiet Mobilności nietknięty przez polskie prawodawstwo mógł wejść w życie, bo wtedy koszty, które potencjalnie byłyby ponoszone przez polskich przewoźników drogowych w każdym innym kraju Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, byłyby dużo wyższe niż to, co my proponujemy w przepisach ustawy. Kiedyś bym zapytał, czy ten wniosek został napisany cyrylicą, ale on nie został napisany cyrylicą. On został napisany przez was po niemiecku albo po francusku i widać, czyje interesy reprezentujecie. Natomiast jeżeli chodzi o sam Pakiet Mobilności, to, szanowni państwo, tym, którzy mówią, że rząd był bierny, że rząd nie walczył z tymi przepisami, chcę bardzo jasno powiedzieć, że Pakiet Mobilności jest dzieckiem Platformy Obywatelskiej, jest dzieckiem Lewicy, jest dzieckiem PSL-u, jest dzieckiem tych frakcji politycznych, które w Parlamencie Europejskim należą do EPP, należą do liberałów i należą do socjaldemokratów. To te frakcje parły jak szalone do tego, aby te przepisy w końcu weszły w życie i niestety próbowały bardzo mocno ograniczyć rynek przewozowy czy bardzo mocno ograniczyć firmy transportowe, które przez ostatnie lata tak wspaniale się rozwijały. Między 2015 a 2019 r. królem czy prezydentem Europy, a formalnie przewodniczącym Rady Europejskiej, był niejaki Donald Tusk. Proszę wskazać choć jeden cytat z tego pana, w którym odnosiłby się do Pakietu Mobilności, jeden cytat, w którym skrytykowałby te przepisy, jeden cytat, w którym by podkreślił, że będą one dyskryminujące dla polskich przewoźników. Ja takiego sformułowania nie znalazłem. Donald Tusk, jeżeli chodzi o Pakiet Mobilności, wywiesił białą flagę. To rząd polski przygotował skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to rząd Prawa i Sprawiedliwości zachęcił do tego dziewięć innych państw: siedem zrobiło to indywidualnie, dwa pozostałe przyłączyły się do Polski, jeżeli chodzi o tę skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Piłeczka jeszcze jest w grze. Używaliśmy w tych skargach nie tylko argumentów gospodarczych, ekonomicznych czy prawnych - prawnych w sensie ograniczenia konkurencyjności - ale używaliśmy również ostatnio bardzo modnych argumentów ekologicznych. Bo Pakiet Mobilności jest pseudoekologiczny, jest antyekologiczny, jest aklimatyczny.

I co Komisja Europejska robi z tą analizą? Na razie jeszcze nic nie robi, aczkolwiek cały czas wywieramy wspólnie z państwami like-minded presję na to, aby ten dokument został użyty do mocnej rewizji Pakietu Mobilności. Skoro argumenty gospodarcze, ekonomiczne, finansowe, prawne nie pomagają, to może w końcu te cudowne argumenty ekologiczne wezmą górę i wskażą drogę postępowania. Tak że piłeczka w ocenie Ministerstwa Infrastruktury jest jeszcze w grze. Jeżeli wygra zdrowy rozsądek, jeżeli wygra logika, to w odniesieniu do Pakietu Mobilności albo w pewnym zakresie powinien zostać on uznany za niewłaściwy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, albo wcześniej Komisja Europejska czy komisarz do spraw transportu pani Vălean powinna sama podjąć inicjatywę legislacyjną, aby przynajmniej te w części szkodliwe przepisy zmienić. I mam podskórne przekonanie, że tak będzie.

Proszę nie obrażać posłów, dobrze?

Jeżeli chodzi o wsparcie dla branży, również zachęcam do odrobienia pracy domowej i do podliczenia, ile w trakcie pandemii COVID-19 branża transportu drogowego uzyskała wsparcia z tarczy antykryzysowej.

Myślę, że wyjdą tutaj bardzo ciekawe liczby.

I to właśnie polskie firmy transportowe z tego dobra będą korzystać. Jeżeli wskazujecie państwo na jakieś nadmierne obciążenia przewoźników czy wszystkich tych, którzy operują w Polsce, to proszę porównać opłaty drogowe, które w tej chwili są w naszym kraju, do opłat, które występują w innych państwach nie tylko Unii Europejskiej, ale też szerzej - w państwach, które nie są zrzeszone w Unii Europejskiej.

Warto też zaznaczyć fakt, że waloryzacji, rewaloryzacji czy podwyższania opłat drogowych w ostatnich latach, przynajmniej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie było. Jeżeli chodzi o kwestie konsultacji, o które pytali państwo posłowie, one odbywały się faktycznie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ministerstwo Infrastruktury złożyło projekt ustawy z prośbą o wpis do wykazu prac rządu jeszcze w kwietniu tego roku, czyli ponad 8 miesięcy temu. Tak trudna i skomplikowana, ale przede wszystkim nowa materia wymagała miesięcy wspólnej pracy ze środowiskiem przewoźników, wcześniej oczywiście ze środowiskiem związków zawodowych, które reprezentowały kierowców. Coś, co leży w interesie przedsiębiorcy, nie do końca leży w interesie związku zawodowego i odwrotnie. Musieliśmy te wszystkie racje zbalansować. Jak część z państwa mogła dzisiaj usłyszeć na posiedzeniu Komisji Infrastruktury nie ode mnie, tylko od przewoźników, którzy byli dzisiaj tam reprezentowani, te przepisy są do przyjęcia, są najmniejszym złem, które w tej chwili może im się przydarzyć. Przechodząc do szczegółów, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń, to regulujemy je dokładnie w taki sam sposób, w jaki są uregulowane zarobki, w jaki jest uregulowany model wynagrodzeń pracowników delegowanych we wszystkich innych dziedzinach, we wszystkich innych zawodach. Tutaj zawód kierowcy, jeżeli chodzi o sposób wynagradzania, będzie podlegał takim samym przepisom jak każdy inny zawód. W Polsce ta sytuacja będzie miała miejsce oczywiście od 2 lutego przyszłego roku. W związku z nowym modelem wynagradzania najwięcej wpływów będzie kierowanych do ZUS i do NFZ, ale to są środki finansowe, z których później kierowcy, czy to przechodząc na emeryturę lub rentę, czy to korzystając ze zwolnienia chorobowego, będą mieli oddawane.

Podobnie - składki na Narodowy Fundusz Zdrowotny. Im większa podstawa odprowadzenia składek, tym większe świadczenie chorobowe w razie niedyspozycji pracownika.

Wykorzystując kilka godzin przerwy między posiedzeniem komisji a drugim czytaniem na sali plenarnej, przepracowaliśmy te poprawki.

To zrobimy.

A, szanowni państwo, dlaczego przez ostatnie lata transport drogowy w Europie się rozwijał? Możemy jeździć swobodnie, nie musimy prosić się o zezwolenia drogowe, tak jak to się działo wtedy, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej.

Właśnie dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, polscy przewoźnicy odnieśli sukces. Gdyby nie bytność w Unii Europejskiej, nawet z tymi wszystkimi - powiedzmy - negatywnymi rzeczami, które się w międzyczasie dokleja, polscy przewoźnicy nie odnieśliby takiego sukcesu.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury celem przedstawienia sprawozdania. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1692) Uprzejmie proszę Przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Marcina Zielenieckiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt - a zarazem jest to duża przyjemność - przedstawienia Wysokiej Izbie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych emerytury stażowej.

Projekt ustawy, jak również jego uzasadnienie, został napisany przez życie.

Chciałbym przedstawić państwu dwie z takich historii. Historia pana Czesława: Mam 62 lata.

Przez 3 lata nauki w zawodzie mechanika samochodowego w szkole przyzakładowej przez 3 dni w tygodniu uczyłem się zawodu, a przez kolejne 3 dni tygodnia pracowałem. Po odbyciu służby wojskowej zacząłem pracować jako mechanik samochodowy, a od 1983 r. - w wytwórni silników wysokoprężnych jako monter hamownik silników spalinowych. Jest to praca w szczególnie szkodliwych warunkach: duży hałas, liczne szkodliwe substancje i związki chemiczne pochodzące z pracy silników. Dawniej posiadałem prawo do dodatku za pracę w szkodliwych warunkach, dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej, a nawet posiłków regeneracyjnych i mleka, aż zakład został sprywatyzowany. Zabrano mi wszystkie dodatki i dziś, mimo że pracuję w jeszcze bardziej szkodliwych warunkach, nie mam nic prócz gołej stawki godzinowej wynagrodzenia. W ciągu 47 lat pracy tylko raz otrzymałem nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Byłem przekonany, że po ukończeniu 60. roku życia będę mógł przejść na emeryturę w obniżonym wieku ze względu na szkodliwe warunki pracy, ale znów się zawiodłem. Okazało się bowiem, że ostatni rocznik, który mógł przejść na ten rodzaj emerytury, to ten, który urodził się w 1958 r. Znów zabrakło mi szczęścia albo raczej taki mamy sprawiedliwy system społeczny w tym kraju. Kiedy wmawia mi się, że mimo 47 lat ciężkiej pracy nie mogę przejść na emeryturę stażową, i wymaga się ode mnie pracy przez 50 lat, to zastanawiam się, czy żyję jeszcze w Europie, czy w jakimś kraju trzeciego świata. Jaki przykład państwo daje młodemu pokoleniu, jak chce je zachęcić do sumiennej pracy, skoro nie ma jakiegokolwiek poszanowania i wdzięczności dla tego pokolenia, które uczciwie i od najmłodszych lat pracowało, pracuje i chyba dalej będzie pracować jak niewolnicy do śmierci? I drugi przykład, przykład pani Katarzyny: W 1983 r. w wieku 15 lat rozpoczęłam naukę zawodu w przyzakładowej szkole zawodowej o profilu: ceramika użytkowa. Przez 3 dni uczyłam się w szkole, przez 3 dni pracowałam na wydziale produkcyjnym, wykonując pracę w szczególnych warunkach. Od 38 lat warunki mojej pracy nie uległy zmianie. Wysoka temperatura, ręczne odlewanie form, ręczne przenoszenie odlewów ceramicznych, dźwiganie i przenoszenie ciężkich desek z odlewami. Od 1986 r. do dziś wykonuję ten sam rodzaj pracy. Gdyby nie to, w wieku 55 lat, po 40 latach pracy, mogłabym przejść na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Dziś nie mam ani prawa do wcześniejszej emerytury, ani prawa do emerytury pomostowej. Zarówno ja, jak i inne panie pracujące w moim zakładzie pracy przy tej ciężkiej, monotonnej pracy narzekamy na problemy z układem ruchu.

ZUS odmawia nam prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jestem wrakiem człowieka. Jestem spracowana, zmęczona. Pracuję w warunkach ciągłego bólu, na lekach przeciwbólowych, bo z czegoś muszę żyć. Wynagrodzenie, jakie osiągam, ani nie daje mi satysfakcji, ani nie rekompensuje mi cierpienia. Zapraszamy do naszego zakładu. Z perspektywy biurka w Warszawie nikt nie jest w stanie ocenić, jak wygląda nasza praca i nasze życie. Przejdę teraz do przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego, zarówno powszechnego jak i rolniczego, emerytury przysługującej wyłącznie z tytuły osiągniętego okresu ubezpieczenia, zwanej dalej: emeryturą stażową. Jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Wprowadzenie tego rozwiązania zapowiedziane zostało przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 r. Od wielu lat z postulatem wprowadzenia emerytur przysługujących z tytułu wysługi występowały związki zawodowe, a Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wprowadził ten postulat do umowy programowej zawartej z prezydentem Andrzejem Dudą w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej. Wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r. system emerytalny, tzw. system zdefiniowanej składki, uzależnia prawo do emerytury od spełnienia przez ubezpieczonego wyłącznie jednego warunku, tj. od osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Staż ubezpieczeniowy w tym systemie nie ma waloru przesłanki nabycia prawa do świadczenia. W rezultacie każda osoba, która przez choćby najkrótszy czas podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu, z chwilą osiągnięcia tego wieku nabędzie prawo do emerytury. Długość okresu opłacania składek wpływa jednak na wysokość emerytury, a także na objęcie ubezpieczonego gwarancją uzyskania świadczenia w wysokości nie niższej od kwoty najniższej emerytury. Taka gwarancja przysługuje wyłącznie ubezpieczonym, którzy legitymują się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. W teorii polityki społecznej od dawna pozytywnie ocenia się fakt posługiwania się przez systemy emerytalne przesłanką stażu ubezpieczeniowego. Okres ubezpieczenia pełni w nich rolę miernika, który pozwala ocenić wkład ubezpieczonego w tworzenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on także stwierdzić, że dochód utracony w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia losowego, w tym przypadku w wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego, osiągany przez ubezpieczonego ma charakter normalny, stały i podstawowy, a nie przejściowy i dodatkowy, i pozwala też wyeliminować z kręgu osób uprawnionych osoby, których przynależność do wspólnoty ryzyka miała charakter incydentalny. Włączenie stażu ubezpieczeniowego do układu warunków nabycia prawa do emerytury jest wyrazem uwzględnienia elementów związanych z wysługą. System emerytalny powinien opierać się na założeniu, że po wielu latach pracy człowiek ma prawo zaprzestać aktywności zawodowej i pozostałą część swojego życia spędzić bez pracy, choćby zachował jeszcze zdolność do zarobkowania. Obawy związane z pozbawieniem wysługi charakteru przesłanki nabycia prawa do emerytury w nowym systemie emerytalnym znajdują potwierdzenie w danych statystycznych dotyczących struktury emerytur wypłacanych przez ZUS w ramach nowego systemu emerytalnego. W ciągu ostatnich 10 lat lawinowo wzrosła w naszym kraju liczba przyznanych i wypłacanych emerytur niższych od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego. Jeszcze w 2011 r. liczba takich emerytur wynosiła niecałe 24 tys., a udział takich emerytur w ogólnej liczbie przyznanych i wypłaconych emerytur z nowego systemu wynosił ok. 4%. W 2020 r. liczba takich emerytur wynosiła czy wynosi już 310 tys., a ich udział w ogólnej liczbie przyznanych i wypłaconych świadczeń wzrósł do prawie 10%. Oznacza to blisko trzynastokrotny wzrost liczby takich świadczeń w ciągu ostatnich 10 lat. Zdaniem wnioskodawców powyższe dane jednoznacznie wskazują na to, że stosowane do tej pory w nowym systemie emerytalnym wyłącznie ekonomiczne zachęty do regularnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, które wpisane są w formułę ustalania wysokości emerytury, okazują się niewystarczające. Ubezpieczeni albo nie dostrzegają korzyści wynikających z systematycznego opłacania wysokich składek, albo traktują te korzyści jako odległą i niepewną perspektywę. W rezultacie konieczne jest zastosowanie nowych, dodatkowych bodźców i taką rolę właśnie mogłoby pełnić wprowadzenie do systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej, która przysługiwałaby ubezpieczonym, którzy osiągnęli odpowiednio długi okres ubezpieczenia jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Możliwość przejścia na taką emeryturę byłaby swego rodzaju nagrodą dla ubezpieczonych, którzy w młodym wieku zaczęli wykonywać pracę zarobkową, a następnie przez wiele lat regularnie opłacali składki na ubezpieczenie emerytalne. Stanowiłaby także wyraz docenienia przez państwo ubezpieczonych legitymujących się długim okresem ubezpieczenia. Mógłby on, nie składając wniosku o taką emeryturę, bez jakiegokolwiek ograniczenia kontynuować wykonywanie pracy po osiągnięciu okresu ubezpieczenia uprawniającego do emerytury stażowej. Konsekwencją długiego i przerwanego okresu wykonywania pracy zarobkowej jest jednak w wielu wypadkach utrata sił uniemożliwiająca jej kontynuowanie do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego - i w tych przypadkach ubezpieczony mógłby zakończyć wykonywanie pracy i cieszyć się z zasłużonej emerytury. W projekcie proponuje się, aby w powszechnym systemie emerytalnym emerytura stażowa przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., tj. objętym nowym systemem emerytalnym, czyli systemem zdefiniowanej składki, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Nabycie prawa do takiej emerytury byłoby uzależnione od jej wysokości. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie byłaby niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego. Ponieważ wysokość emerytury obliczonej według tej formuły zależy przede wszystkim od takich czynników jak wartość składek na ubezpieczenie emerytalne wpłacone w okresie aktywności zawodowej, jak również średnie dalsze trwanie życia osób w wieku osoby przechodzącej na emeryturę, prawo do emerytury stażowej przysługiwałoby ubezpieczonym, którzy legitymują się długim okresem składkowym i nieskładkowym pod warunkiem opłacania za nich składki na ubezpieczenie emerytalne od odpowiednio wysokiej podstawy wymiaru. W systemie rolniczym ten projekt zakłada również objęcie osób objętych systemem ubezpieczenia społecznego rolników prawem do takiej emerytury stażowej. Tak że w tym systemie prawo do tej emerytury przysługiwałoby osobom legitymującym się okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu wynoszącym 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Emerytura stażowa również (Dzwonek) w ich przypadku nie mogłaby być niższa od najniższego świadczenia emerytalnego. Dwa słowa na temat skutków finansowych. W uzasadnieniu tego projektu macie państwo dokonane szacunki dotyczące kosztów finansowych tego projektu. One zostały przygotowane w oparciu o dostępne dane dotyczące właśnie skutków finansowych wprowadzenia emerytury stażowej dla osób, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. Ale te szacunki nie uwzględniają tego ograniczenia, o którym wspominałem, tzn. ograniczenia zakresu podmiotowego tego prawa do emerytury stażowej do osób, które wypracowały sobie emeryturę w kwocie najniższej emerytury. Te skutki zostały wyliczone w dwóch wariantach, tzn. w wariancie, w którym z takiego świadczenia skorzystałaby tylko połowa osób uprawnionych, i w wariancie, w którym wszyscy uprawnieni skorzystaliby z tego rozwiązania.

Już kończę.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zwracam się do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wprowadzającej do polskiego systemu ubezpieczenia społecznego emeryturę stażową. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Janusz Śniadek. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam honor w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczonej Prawicy przedstawić stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, druk nr 1692. Przyznaję, że dzisiaj staję tutaj z wyjątkowo ciężkim sercem, bo chciałbym móc zadeklarować, że jest jednoznaczne stanowisko Zjednoczonej Prawicy, zgodnie z apelem pana Zielenieckiego w imieniu komitetu wzywającego do poparcia tej ustawy.

W roku 2008, kiedy toczyliśmy bój o emerytury pomostowe, przegrany zresztą na wiele miesięcy, po raz pierwszy zaczął się pojawiać, już jako ogólnozwiązkowy, postulat emerytur stażowych. On się przewijał dalej, ale działo się to wszystko właśnie w momencie wycofania postulatu czy uprawnień do emerytur pomostowych wbrew deklaracjom wyborczym w 2011 r. W 2012 r. nastąpiło podniesienie wieku emerytalnego o 2 lata dla mężczyzn, 7 lat dla kobiet, 12 lat np. dla kobiet w KRUS-ie.

Również jeśli chodzi o politykę społeczną, to Prawo i Sprawiedliwość wykonało wiele działań, m.in. można przytoczyć przykłady corocznej wypłaty trzynastej emerytury od 2020 r. czy wzrostu najniższej emerytury od 2015 r. do dzisiaj, sięgającego ponad 40%. Przedstawiany projekt zakłada, że zgodnie z dodawanym ubezpieczeniem urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. będzie przysługiwała emerytura, jeżeli okres składkowy i nieskładkowy wyniesie co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn, oraz że emerytura przysługująca z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określona w art. 26, łącznie z okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z funduszu określona w art. 26 jest co najmniej równa kwocie najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ustawy. Przyznam jednak, że to uzależnianie prawa do emerytury od wysokości świadczenia wynikającego ze zgromadzonego kapitału jest trochę problematyczne. Spoglądam na czas, a chciałem choć troszkę odnieść się jeszcze do kosztów, o których wspominał pod koniec pan Marcin Zieleniecki.

W każdym razie zakończę tylko podsumowaniem, że są wyliczone szacunkowe łączne skutki finansowe w okresie 10 lat od wejścia w życie proponowanych zmian przepisów w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2020 r. w cenach stałych z tego roku.

Wysoka Izbo, wnoszę o skierowanie tego projektu do dalszych prac. Pani poseł Joanna Frydrych w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawiam stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Obywatelski projekt ustawy zakłada wprowadzenie emerytur, do których prawo uzależnione jest od stażu pracy ubezpieczonego niezależnie od jego wieku. Udowodniony okres składkowy i nieskładkowy wynosiłby dla kobiet 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat. Wysoka Izbo! System emerytalny ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Rozwiązania funkcjonujące w Polsce uzależniają przyznanie prawa do emerytury od osiągnięcia wieku emerytalnego. Zasady dotyczące ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego oparte są na modelu zdefiniowanej składki. Im więcej do systemu odprowadził ubezpieczony w postaci składek, tym więcej z systemu otrzyma jako świadczeniobiorca. System ten należy ocenić jako nowoczesny i odpowiadający na wyzwania demograficzne. Każdy ubezpieczony powinien ocenić, jakie świadczenie otrzyma i co powinien zrobić, aby je pomnożyć. Trzeba mieć jednak świadomość, że z roku na rok rośnie skala ubóstwa emerytalnego w Polsce. Pod koniec grudnia 2015 r. 76 tys. emerytów pobierało emerytury niższe od minimalnej. Polityka rządu PiS spowodowała, że pod koniec 2020 r. liczba takich emerytów wzrosła do 310 tys. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wzrost liczby osób wykluczonych społecznie.

Tyle osób żyje dziś poniżej granicy skrajnego ubóstwa, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Mówimy w tym momencie o życiu za mniej niż 20 zł dziennie. Jedną z obietnic był np. wzrost emerytur. Kłamaliście, a jedyne co wam wyszło, to drożyzna, inflacja i horrendalne liczby zgonów. Jeżeli Polki i Polacy skorzystają z emerytur wprowadzonych przedmiotową ustawą, wielu z nich będzie skazanych na niskie świadczenia.

Jeżeli ten mężczyzna skorzysta z emerytury stażowej, otrzyma świadczenie w wysokości 2564,61 zł, czyli o 619,59 zł miesięcznie niższe. Natomiast średnia emerytura dla kobiety przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat wynosi 2127,81 zł. Jeżeli ta sama kobieta skorzysta z emerytury stażowej, otrzyma świadczenie w wysokości 1743,18 zł, czyli o 384,63 zł miesięcznie niższe. Jeżeli poddamy analizie dokładne dane, różnice te mogą być większe. Dlatego wprowadzając nowy komponent do systemu emerytalnego, należy wprowadzić elementy kształtowania świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie, żeby ubezpieczony w pełni świadomie dokonywał swojego wyboru rezygnacji z aktywności zawodowej i miał pełną wiedzę o wysokości przyznanego świadczenia, żeby to był jego wybór, a nie wypychanie go z rynku pracy. To jest obowiązek oraz odpowiedzialność rządu. Kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej wśród Polaków będzie wyrażało troskę o wysokość przyszłych świadczeń oraz zwiększy zainteresowanie pracowników wykonywaniem pracy rejestrowanej, zmniejszy skalę zatrudnienia w szarej strefie, co przełoży się na zgromadzenie większego kapitału emerytalnego i uniknięcie pogłębiania się ubóstwa emerytalnego. Ponadto rząd musi odpowiedzialnie prowadzić politykę demograficzną oraz politykę migracyjną, by nie zachwiać rynkiem pracy. To też są bardzo ważne obszary, które świecą się na czerwono, bo obecny rząd w tych obszarach również nic nie robi. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z racji tego, że jest to projekt obywatelski i jest duże oczekiwanie (Dzwonek) społeczne, jeśli chodzi o wprowadzenie emerytur stażowych, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska składam wniosek o skierowanie tego projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Emerytury stażowe są przede wszystkim sprawiedliwym rozwiązaniem. Osoba, która pracuje 35–40 lat, która odprowadza składki i uczciwie płaci przez te wszystkie lata podatki, powinna móc odejść na zasłużoną emeryturę niezależnie od tego, czy po 40 latach pracy ma 55 czy 65 lat. Dlatego Lewica oczywiście popiera ten projekt. Potrzebujemy jako społeczeństwo od was, od posłów i posłanek partii rządzącej, jak również od posłów i posłanek opozycji myślenia o tym, jak zagwarantować nam wszystkim godne życie na europejskim poziomie, a nie kombinowania, jakby tu najmniej wypłacić, jak oszczędzić na obywatelach, na emerytach, na pacjentach. Niestety, takie spojrzenie, mam wrażenie, dominuje na tej sali od lat. Z takim podejściem Lewica nigdy się nie zgodzi. Związki zawodowe od przeszło dekady walczą o emerytury dla osób z najdłuższą wysługą lat. PiS wraz ze swoim kandydatem na prezydenta obiecywał je w kolejnych kampaniach. Ze związkowcami spotykał się premier Morawiecki.

Procedujemy dziś nad projektem obywatelskim nie dlatego, że chcieliście, ale dlatego, że musicie tego wysłuchać. Domagają się tego obywatele. Projekt jak żaden inny cieszy się poparciem miażdżącej większości społeczeństwa. Wiemy z doświadczenia, że obiecaliście obywatelom i związkowcom emerytury stażowe, ale nie macie najmniejszej ochoty ich wprowadzić. Po dzisiejszej debacie dowiemy się, czy będziecie dalej cynicznie kłamać w żywe oczy, czy będziecie nadal nad tym procedować, czy wbrew własnym zapewnieniom odłożycie to do zamrażarki. Tymczasem pragnę zwrócić uwagę koleżanek i kolegów z obu stron sali na to, że samo wprowadzenie emerytur stażowych bez zagwarantowania ich godnego poziomu ponownie wykluczy z tego rozwiązania osoby najciężej pracujące, które często otrzymują niskie wynagrodzenia.

Państwo - mimo że tak chwalicie się swoim prosocjalnym podejściem - nie zrobiliście absolutnie nic, żeby tamte błędy naprawić. Ten pomysł, który zgłosiliśmy, także leży w zamrażarce.

W Polsce potrzebujemy systemu emerytalnego, który zapewni godne emerytury na poziomie adekwatnym do kosztów życia. Potrzebujemy ich, by zachęcić do podejmowania legalnego zatrudnienia i co za tym idzie - płacenia podatków. Potrzebujemy godnych emerytur także do tego, by utrzymać koniunkturę na rynku, bo do 2035 r. już 27% Polaków będzie pobierało emerytury.

Wiemy, że rozwiązania gwarantujące Polkom i Polakom dobre emerytury, dobrą edukację, dobrą ochronę zdrowia, życie na europejskim poziomie są możliwe, są opłacalne i jak najbardziej wykonalne - dziś, tu, w Polsce. Świadczą o tym sukcesy podobnych rozwiązań w innych krajach europejskich, opinie ekspertów i matematyka, bo to wszystko wyliczyliśmy. Jedyne, czego brakuje dziś rządzącym - w przypadku emerytur stażowych widać to bardzo dokładnie - to wola, aby te rozwiązania wprowadzić, aby zrealizować obietnice i wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec społeczeństwa. Nam na lewicy tej woli nie brakuje i dlatego popieramy obywatelski projekt wprowadzający emerytury stażowe. Dziękuję, pani poseł. Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawię stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw z druku nr 1692. Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia, tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Godna emerytura to niezbywalne prawo każdego ciężko pracującego człowieka, a ustawa ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników i jest odpowiedzią na ich głosy. 35 lat opłacania składki przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn to wystarczający okres, żeby zgromadzić środki na co najmniej minimalną emeryturę, a tylko do takiej dopłaca budżet państwa w przypadku jej nieosiągnięcia. Należy docenić tych, którzy odprowadzają składki i ciężko pracują, często fizycznie, od najmłodszych lat, i dać im prawo wyboru, czy chcą dalej pracować, czy chcą skorzystać z prawa do emerytury. Emerytura stażowa to wybór, nie konieczność, dlatego każdy, kto będzie czuł się na siłach, aby dalej pracować, będzie miał taką możliwość, co - jak pokazuje sytuacja na rynku pracy - jest dobrym rozwiązaniem dla emerytów, ale również dla pracodawców, którzy nie tracą doświadczonych pracowników. Ustawa ta, co jest niezwykle istotne, nie dyskryminuje rolników, którzy również mają szansę skorzystać z emerytury stażowej, bo to oni, pamiętajmy, ciężko pracują od najmłodszych lat i jak wynika ze statystyk, mają niestety najniższe emerytury. Pokazuje bowiem, że kapitał na przyszłą emeryturę należy budować już od samego początku pracy zawodowej.

Ten projekt niestety, drodzy państwo, trafił do zamrażarki, w której jest do dzisiaj. Gdyby wszedł w życie w ubiegłym roku, to już przez ten cały rok przyszli emeryci mogliby z tego korzystać. Dlatego klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera projekt tej ustawy i skierowanie go do dalszych prac. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Z przerażeniem słucham tej debaty i tego zalewu demagogii z państwa strony.

W 2060 r. liczba emerytów może wynieść ok. 12 mln. Kurczy nam się baza pracujących, powiększa się baza emerytów, w wiek emerytalny wchodzą roczniki najbardziej liczne. Jest wielka, gigantyczna dziura w środku naszego budżetu, a wy rozmawiacie o jej powiększeniu. Uchwalanie takiej ustawy to jest działanie na pograniczu zdrady stanu po prostu. 1/3 wszystkich wydatków sektora publicznego już w tej chwili stanowią emerytury.

Jeśli zsumujemy wydatki na emerytury, to będą one równe łącznym wydatkom na bezpieczeństwo wewnętrze, czyli policję, sądy, więziennictwo itd., bezpieczeństwo zewnętrzne, czyli armię, ochronę zdrowia i całe szkolnictwo, łącznie ze szkolnictwem wyższym.

Ale ten ktoś oprócz tego, że będzie musiał utrzymać z pracy siebie i płacić na wszystkie obecne wydatki państwowe, będzie musiał jeszcze utrzymać pana Czesława i panią Jadwigę. Do tego chcecie doprowadzić.

Za 35 lat pracy dostanie 29 lat emerytury.

70 mld zł w ciągu 10 lat ma kosztować ten pomysł.

Uprzejmie dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Szanowni Państwo!

Oczywiście ten projekt ustawy może stanowić głos w dyskusji. Jest to rozwiązanie, które umożliwia pracownikom posiadającym określony staż pracy odejście na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Wnioskodawcy proponują, aby na emeryturę mogły odejść kobiety po przepracowaniu 35 lat i mężczyźni po przepracowaniu 40 lat.

To bardzo wysoki koszt, biorąc pod uwagę to, że już w 2015 r. według GUS-u ten ukryty dług emerytalny wynosił niemalże 4960 mld zł. To jest potężny koszt, który jest nałożony na barki naszych dzieci i wnuków, bo kiedyś te pieniądze trzeba będzie wypłacić.

Co prawda wnioskodawcy przewidują pewien mechanizm zabezpieczający, niemniej jednak dla kobiet będzie to zazwyczaj albo minimalna, albo zbliżona do minimalnej wysokość. Na dodatek rząd Prawa i Sprawiedliwości chce pozbawić członków otwartych funduszy emerytalnych 15% zgromadzonych kapitałów, czyli znów oznacza to pomniejszenie emerytur. Dzisiaj potrzebna jest oczywiście bardzo szeroka dyskusja na temat aktywizacji zawodowej jak największej liczby Polaków. Mamy poczucie, że tutaj brakuje propozycji. Można skorzystać z tych, które są zawarte w programie gospodarczym Polski 2050, związanych z przeznaczeniem 8-procentowej składki rentowej na składkę emerytalną czy też wypłaceniem wszystkich utraconych emerytur, 13. emerytur osobom, które zdecydują się na późniejsze przejście na emeryturę, [[Dzwonek]] niemniej jednak dzisiaj obywatele oczekują wyższych emerytur i stabilnych warunków w systemie emerytalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Dzisiaj debatujemy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, pod którą podpisało się 235 tys. obywateli popierających ten projekt ustawy. Projekt ten jako cel główny przyjmuje osiągnięcie okresu ubezpieczeniowego do uzyskania emerytury z powszechnego i rolniczego systemu emerytalnego. Wykorzystanie okresu ubezpieczeniowego jako miernika pozwala ocenić wkład ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeniowego i ma pozytywny odbiór społeczny. Bardzo zła tendencja do przechodzenia na emeryturę osób otrzymujących świadczenia emerytalne niższe od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego świadczy o tym, że obecne rozwiązania polegające na zachęcaniu do regularnego opłacania składek są niewystarczające. 310 tys. osób w roku 2020 otrzymywało emerytury niższe od najniższego świadczenia emerytalnego. Jest to trzynastokrotny wzrost w porównaniu do roku 2011. Mając na uwadze takie zachowania ubezpieczonych, należy szukać nowych rozwiązań w celu osiągania długiego okresu ubezpieczenia jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przejście na emeryturę po 35 latach dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn okresu składkowego i nieskładkowego, przed osiągnięciem wieku emerytalnego - będzie nagrodą dla ubezpieczonych i docenieniem przez państwo za długoletnie okresy ubezpieczenia. Kolejnym wyzwaniem jest niedopuszczenie, aby emerytura stażowa była niższa od najniższego świadczenia emerytalnego. Emerytura stażowa będzie uprawnieniem, a nie obowiązkiem ubezpieczonego, dlatego może on kontynuować pracę po osiągnięciu okresu ubezpieczenia uprawniającego do emerytury stażowej. Musimy pamiętać także, że są zawody czy rodzaje pracy wykonywane przez ubezpieczonych, gdzie sprawność psychofizyczna jest niezbędna dla bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy. Szanowni państwo, nie wszyscy są pracownikami na stanowiskach nierobotniczych. Podam własny przykład. Praca w systemie 4-brygadowym, na trzy zmiany, na mrozie, na wysokościach, 30 m - jako młody człowiek przez 11 lat taką pracę mogłem wykonywać, ale w wieku 60 lat nawet bym nie miał co się do tej pracy zbliżać. A więc trzeba wziąć pod uwagę, że są ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują. Nie wszyscy mogą skończyć studia i mieć zawody, pracować na stanowiskach nierobotniczych.

Przechodzimy do pytań. Jednocześnie proszę, byście państwo nie przekraczali określonego czasu, bo jest sporo osób, które zapisały się do pytań. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Nie widzę. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Chciałam zapytać, bo pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że nie ma stanowiska rządu, dlaczego tego stanowiska nie ma i kiedy to stanowisko będzie, żebyśmy się dowiedzieli, jak państwo wypowiadacie się w sprawie tej inicjatywy. Wnioskodawców chciałam zapytać, czy dobrze zrozumiałam, że nie każdy będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, z emerytury stażowej - jeżeli jego zgromadzone składki nie pozwolą na osiągnięcie emerytury minimalnej, wtedy on nie przechodzi na emeryturę, on będzie musiał dalej pracować. Może w tym przypadku trzeba pomyśleć o innym rozwiązaniu?

Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski z klubu Lewica zada kolejne pytanie.

Mamy 29 osób. Pani Marszałek!

Pewno miejsce siedzenia zmienia punkt widzenia. 22 lipca 2010 r. poseł Stanisław Szwed, reprezentujący klub Prawa i Sprawiedliwości, o emeryturach pomostowych w czasie pierwszego czytania tej ustawy mówił: „Budżet państwa, budżet ZUS nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów, chyba że w wyjątkowych przypadkach, gdy ktoś nie ma środków wypracowanych na minimalną emeryturę, wtedy budżet państwa musiałby dopłacić. Nie przypuszczam, żeby była to jakaś znaczna grupa osób” W odpowiedzi na moją interpelację 1 grudnia tego roku pan minister pisze, że koszty to w pierwszym roku 7,4 mld zł. W związku z powyższym pisze pan również, że będzie stanowisko rządu. Czy to będzie stanowisko rządu, które przekazał pan w interpelacji? Czy będzie zmiana stanowiska ministerstwa pracy na rzecz korzystnego stanowiska rządu? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Sytuacja jest jasna.

To oznacza, szanowni państwo, że będzie coraz gorzej, jeśli chodzi o rynek pracy. To oznacza, że przy wydłużającej się, cały czas się zwiększającej, pomijając ostatnie 2 lata, średniej długości życia w Polsce będziemy mieli miliony emerytów. Cały wysiłek legislacyjny, cały wysiłek państwa polskiego musi być skoncentrowany na tym, żeby jak najdłużej ludzie mogli być aktywni zawodowo, a nie na tym, żeby jak najszybciej odsyłać ich z rynku pracy na emeryturę. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szanowni Panowie Przedstawiciele Wnioskodawców!

I pytanie do pana ministra: Czy prawdą jest to, co zostało przedstawione w opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że projekt przedstawiony przez grupę społeczną jest sprzeczny z celami tzw. Polskiego Ładu oraz planami aktywizacji zawodowej, co do której chyba wszyscy się tutaj zgadzamy, że jest to niezwykle potrzebne? Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To pokazuje, że żyjemy w państwie obywatelskim, nie tak jak było za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy prawie 300 tys. związkowców manifestowało przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Nie było miejsca na żadną debatę za waszych rządów. Cieszę się z tego, że „Solidarność” się do tego przyczyniła, składając projekt obywatelski, który pozwoli na poziomie komisji sejmowych, na poziomie polskiego parlamentu na debatę dotyczącą miejsca emerytur stażowych w polskim systemie emerytalnym. Mamy też projekt prezydencki.

Czy jest szansa, aby pracować jednocześnie nad tymi dwoma projektami? Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wnioskodawcy! W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że wprowadzenie tego rozwiązania zapowiedziane zostało przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 r. Od wielu lat z postulatem wprowadzenia emerytur przysługujących z tytułu wysługi występowały związki zawodowe, a NSZZ „Solidarność” wprowadził ten postulat do umowy programowej zawartej z prezydentem Andrzejem Dudą w trakcie ostatniej kampanii wyborczej. Jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Tak. Uważam, że to rozwiązanie powinno być korzystne dla wielu osób. Przypomnę tylko przy okazji, że oczekiwań społecznych jest dużo więcej, np. niezawisłe i szybko pracujące sądy, [[Oklaski]] prawo do rzetelnej informacji, pomoc ludziom poszkodowanym przez systemy bankowe. Tym ludziom pan prezydent też obiecywał wsparcie. Jakoś nie wyszło.

W związku z tym mam pytanie, na ile rzetelne są te obliczenia, skoro nie uwzględniają grupy społecznej, czyli rolników.

Wysoka Izbo! Dzisiejszą debatę można zdefiniować w sposób następujący: pan Duda zrobił niedźwiedzią przysługę panu Dudzie. Chodzi o rozwiązanie, które prezydent obiecał przecież wszystkim Polakom podczas kampanii wyborczej. Panie Prezydencie! Od zakończenia kampanii wyborczej mijają 2 lata. Czy faktycznie w tym czasie cała Kancelaria Prezydenta z budżetem ponad 200 mln zł rocznie nie była w stanie przygotować tego projektu? Czy 420 zatrudnionych w Kancelarii Prezydenta pracowników nie znalazło czasu na przygotowanie lub zlecenie przygotowania ustawy spełniającej wyborcze obietnice prezydenta naszego kraju? Może trzeba zrewidować omawiany w dniu dzisiejszym budżet pana prezydenta? Dzisiaj podziękowania należą się panu przewodniczącemu Dudzie. Bardzo proszę. Kiedy państwa brały się za wdrażanie systemów emerytalnych, na jednego pracującego przypadało kilku, nawet kilkunastu pracujących. Ludzie do emerytury przeważnie nie dożywali, a jak dożywali, to byli na niej kilka lat. W tej chwili ludzie żyją coraz dłużej, wchodzą na rynek pracy coraz później, m.in. przez lansowaną przez państwo modę na studiowanie na koszt podatnika. Efekt jest taki, że niedługo, w 2060 r., na 12 mln emerytów będzie przypadało 17 mln pracujących, jak dobrze pójdzie. Już w tej chwili, żeby ten system się trzymał, jesteśmy zmuszeni importować siłę roboczą z zagranicy, ale w ten sposób tylko opóźniamy katastrofę i powiększamy ją na przyszłość, bo ci ludzie, pracując tutaj, po prostu nabywają prawa do emerytur.

Jaki macie pomysł, jedni, drudzy, trzeci - wszyscy na wyjście (Dzwonek) z tego impasu, a nie na pogłębianie go? Panie Ministrze! Projekt ustawy obywatelskiej przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego zarówno powszechnego, jak i rolniczego tzw. emerytury stażowej. Projekt ustawy proponuje, aby emerytura stażowa przysługiwała osobom urodzonym po 1 grudnia 1948 r., które osiągnęły wysokość stażu pracy dla kobiet - 35 lat i dla mężczyzn - 40 lat. Panie Ministrze! Mam pytanie, czy ministerstwo posiada na chwilę obecną wyliczenia kosztów dotyczących wprowadzenia tejże emerytury stażowej oraz czy przejście na emeryturę stażową będzie dobrowolne dla osób, którym, powiedzmy, stan zdrowia nie pozwala (Dzwonek) na to, aby w dalszym ciągu pracować. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie zauważyłam, aby zmianie ustawy emerytalnej towarzyszyła niezbędna zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie ochrony przedemerytalnej, która obecnie jest przewidziana w art. 39. Co to oznacza? W praktyce nic nie będzie stało na przeszkodzie, by pracodawca zwolnił pracownika z uwagi na emeryturę stażową, do której nabył on prawo. I tu rodzą się pytania i wątpliwości. Czy emerytura stażowa będzie uprawnieniem socjalnym, czy nabyciem właściwej emerytury? Czy przepisy Kodeksu pracy nie powinny jednoznacznie wskazywać, że nabycie prawa do wcześniejszej emerytury stażowej objęte zostanie uprawnieniami ochronnymi i czy nie powinien obowiązywać w tym wypadku zakaz wypowiadania umowy o pracę do czasu osiągnięcia właściwego wieku emerytalnego, odpowiednio 60 i 65 lat? To ubezpieczony sam (Dzwonek) powinien decydować po uzyskaniu uprawnienia, czy z niego skorzysta, czy też nie, a uprawnienia do emerytury stażowej nie są i nie powinny być przesłanką do rozwiązania stosunku pracy. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Wysoka Izbo! Panie Przewodniczący! W ramach procesu legislacyjnego otrzymaliśmy opinię Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 8 grudnia 2021 r., gdzie rada rolników zwraca uwagę, że proponowane zmiany w przedmiotowym projekcie ustawy będą generować dodatkowe koszty związane z modyfikacją systemów informatycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które nie zostały uwzględnione w budżecie kasy.

Pan poseł Mariusz Trepka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Dlatego uważam, że ta ustawa powinna wejść w życie.

Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska, zada kolejne pytanie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Ta ustawa wyklucza pewną dużą grupę osób i dlatego o sprawiedliwości historycznej, dziejowej chyba nie można mówić.

Gdy odchowała dzieci, a mama zmarła, mogła pójść do pracy i miała 43 lata.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Bólem każdego rządu jest ilość pieniędzy wpływających do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego od kilkudziesięciu lat kombinujemy jak konie pod górę, jak te pieniądze zdobyć, i manipulujemy, ile ich wypłacić dla emerytów i rencistów. I dlatego Donald Tusk wziął kilkadziesiąt miliardów złotych z komercyjnych funduszy emerytalnych, dlatego PiS dokończył tego dzieła. Każdy rząd się martwi, ile ma do funduszu dopłacić.

Dzisiaj mamy warunki bardzo dobre, bo bezrobocie jest znikome, Polacy zarabiają coraz więcej. To kiedy mamy wprowadzić systemowe rozwiązanie, że wprowadzamy drugie kryterium otrzymywania emerytur i rent? Właśnie teraz trzeba to zrobić. Ale jak będziemy bogatszym krajem i będziemy bogatsi, to sobie z tym poradzimy. Trzeba ludziom dać szansę. Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość - z przeprosinami, że pana pominęłam. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Posłowie opozycji zarzucają, że ten projekt jest niesprawiedliwy.

Wtedy jako student farmacji w Poznaniu prowadziłem akcję zbierania podpisów, prowadzoną przez związek „Solidarność”

Pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Ale właśnie pan ciągle coś mówi, panie pośle. Bardzo pana proszę o spokojne przysłuchiwanie się obradom, a nie ciągłe dziamgolenie. Panie pośle, zwracam panu uwagę. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo. Bardzo proszę, pani poseł, dodam czas. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nikt z przedmówców z Koalicji Obywatelskiej nie powiedział, że ten projekt jest niesprawiedliwy. Wszyscy mówią, że jest absolutnie wart dalszych prac w komisji. Takie rozwiązania funkcjonują w różnych krajach zachodnich, tylko oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, więc musimy głęboko się zastanowić nad konkretnymi zapisami, bo oprócz dawania ludziom możliwości przechodzenia na świadczenia po przepracowaniu określonego stażu trzeba również tworzyć system zachęt do pozostania na rynku dla tych, którzy chcą na nim zostać. W 2017 r. została podana informacja o przygotowywanych przez rząd propozycjach. Wtedy pani premier Szydło mówiła, że to jeden z dyskutowanych wariantów. Bo jakoś żadnego z nim nie ujrzeliśmy. Rząd nie zrobił nic, by wesprzeć system emerytalny.

Przepraszam. Pani poseł, bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! Pan poseł Śniadek, sprawozdając stanowisko klubu Zjednoczonej Prawicy, powiedział, że właściwie klub nie ma zdania. Szczerze mówiąc, nie mieści mi się w głowie, jak można nie mieć zdania o obywatelskim projekcie, który poprawia sytuację osób, które naprawdę ciężko pracowały przez całe życie i powinny móc z tej swojej pracy skorzystać. Jak rozumiem, to trochę wyjaśnia też to, dlaczego np. projekt Lewicy zapewniający emeryturę minimalną tym osobom, które lata przepracowały na umowach-zleceniach, na śmieciówkach i na starość będą dostawać kilkaset złotych emerytury, również jest w zamrażalce sejmowej. Dlatego że nie mają państwo zdania o tym, że ludzie powinni dostawać na starość godne pieniądze. Dobry wieczór państwu. Pani poseł Ewa Kołodziej, Koalicja Obywatelska. Zapraszam serdecznie wieczorową porą. To może zagwarantować jedynie godna emerytura, która seniorom zarówno pozwoli zapłacić wszystkie finansowe zobowiązania, jak i pozwoli przynajmniej na drobne przyjemności. W związku z tym moje pytania.

Z czego wynika ta różnica? Czy przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej mają wiedzę, czy macie państwo jakieś takie wstępne symulacje, ile będzie wynosiła ta emerytura stażowa? Czy mają państwo również wiedzę, jakieś symulacje, ile osób skorzysta z tej emerytury? Bo my podejrzewamy, że to będzie kwota niestety bardzo niska, wynosząca 1250 zł (Dzwonek), która będzie wpędzała seniorów w ubóstwo. Ludzie będą popadać w tarapaty finansowe, w związku z czym będą być może żałowali swoich decyzji. Będą mamieni waszymi obietnicami wysokich emerytur, a potem będą chcieli wrócić na swoje stanowiska pracy, a to stanowisko pracy będzie już zajęte, bo ktoś już zajmie ich miejsce. W związku z tym co przewidujecie dla tych ludzi, którzy niestety zostaną oszukani obietnicą dużych pieniędzy z waszej strony, a życie okaże się brutalne i te emerytury będą bardzo niskie? Czy przewidujecie jakieś świadczenia socjalne dla tych osób, które będą mieć te emerytury stażowe?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiciele Inicjatywy Ustawodawczej! To całkiem niezły projekt obywatelski o emeryturach stażowych. Ten pozytywny to możliwość wyboru po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 przez mężczyzn. Jak najbardziej, każdy powinien mieć prawo wyboru, czy chce pozostać na rynku pracy, czy chce skorzystać ze świadczenia emerytalnego. Ta druga strona to jednak fakt, że z rynku pracy może zniknąć blisko 400 tys. osób, niezwykle cennych dla rynku pracy. Dlatego pytam, jakie są analizy rządu w tym zakresie. Dlaczego rząd nie ma stanowiska? Czy dlatego, że jest to projekt obywatelski?

Zapraszam panią poseł. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Projekt ustawy stażowej umożliwia Polakom wybór terminu przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobiety, a 40 lat przez mężczyzn. Wiele kobiet i mężczyzn pracuje bardzo długo. Niektórzy już od 15. roku życia, zwłaszcza wtedy kiedy rozpoczynali naukę w szkołach zawodowych, równolegle z nauką pracowali.

Zapytam o grupę ludzi, którzy pracują w rzemiośle, pracują bardzo długo. Płacili i płacą niskie składki, ale uważam, że (Dzwonek) ta sprawa musi być rozpatrzona szczególnie. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowni Wnioskodawcy! Ubóstwo, ubóstwo osób starszych jest coraz większym problemem w Polsce. Ubóstwo kobiet jest problemem narastającym. Kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę, te emerytury są mniejsze, a kobiety żyją dłużej. Pytanie do państwa jest takie - bo postulat, żeby każdy mógł sobie wybrać w każdym obszarze życia jest słuszny - w jaki sposób państwo zamierzacie przeciwdziałać ubóstwu kobiet, przeciwdziałać wypychaniu ich z rynku pracy, proponując takie rozwiązania.

Jakie są programy przeciwdziałające temu, by Polki na emeryturze nie były biedne i nie były głodne? Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Szczerba. Jeżeli nie ma pana posła Michała Szczerby, to znaczy, że jest z nami pan poseł Dariusz Joński. To znaczy, że mam 2 minuty? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do wnioskodawców, dlatego że mam umowę programową „Solidarności” z wtedy kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Nie jest ona zbyt długa, ale jest tutaj zobowiązanie dotyczące m.in. właśnie emerytur stażowych. Minęło 5 lat, nic się w tej sprawie nie stało. Przed kolejną kampanią pan prezydent Duda znowu podpisał z państwem porozumienie, obiecując, że będą emerytury stażowe. Co prawda chwilę później już udzielił wywiadu i powiedział, że postulat ten jest bardzo trudny do spełnienia z punktu widzenia systemu ubezpieczeń społecznych.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Małgorzata Niemczyk, Koalicja Obywatelska.

Szanowni Państwo! Chyba wiem, dlaczego klub PiS-u nie ma stanowiska w tej sprawie, dlaczego rząd nie ma stanowiska w tej sprawie. Dlatego że oni po prostu już nie mają pieniędzy. Chciałbym się z tej mównicy upomnieć o tych, którzy pracują. Dzisiaj czytałem raport dotyczący dostępności mieszkań dla ludzi pracujących, młodych, którzy nie mają własnego mieszkania. Połowa z nich nie ma szansy na własne mieszkanie, nigdy, a państwo proponujecie ustawę, która nakłada kilkadziesiąt miliardów zobowiązań, nikt nie wie, czy 20 czy 50, która zmniejsza liczbę ludzi pracujących i nakłada obowiązki na ludzi pracujących. Wy po prostu nie macie na to pieniędzy. Wtedy „Solidarność” powstała dlatego, że państwo zbankrutowało. Dzisiaj to nie jest „Solidarność” Wałęsy, tylko to dzisiaj „Solidarność” podcina gałąź i wydaje pieniądze, których nie ma. To się skończy dokładnie taką samą katastrofą gospodarczą, bo ludzie nie będą w stanie tego waszego systemu niby-socjalnego utrzymać. Skończycie dokładnie jak Polska w roku 1989, która zbankrutowała, bo ludzie nie będą w stanie na ten system zarobić.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że postulat zapewnienia pracownikom o długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego cieszy się bardzo wysokim poparciem społecznym. Zaletą procedowanej ustawy jest również fakt, iż ewentualna decyzja o przejściu na emeryturę pozostawałaby w gestii samych zainteresowanych, a w przypadku braku usatysfakcjonowania wysokością świadczenia taka osoba mogłaby zdecydować o dalszej pracy. Wsłuchując się w argumenty obu stron na temat celów tej ustawy, proszę wnioskodawców o odpowiedź na pytanie, czy tzw. emerytura stażowa nie spowoduje obniżenia ogólnego poziomu emerytur i zmniejszenia podaży pracy osób w wieku przedemerytalnym, które spełniałyby (Dzwonek) warunek stażu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Mam pytanie do przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, do pana ministra Marcina Zielenieckiego. Szanowny panie ministrze, mówił pan, że prezydent obiecał emerytury stażowe i że zostało podpisane porozumienie z „Solidarnością” Dzisiaj prezydent Andrzej Duda złożył projekt dotyczący emerytur stażowych, ale zdecydowanie różni się on od obywatelskiego. Warunkiem przyznania emerytury według prezydenckiego projektu jest 39 lat stażu pracy dla kobiety i 44 lata pracy dla mężczyzny. Do niedawna był pan wiceministrem w Ministerstwie Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny. Wielokrotnie, nawet wspólnie, uczestniczyliśmy w konferencjach Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Był pan przecież członkiem zarządu. Jest pan fachowcem w dziedzinie polityki społecznej, przede wszystkim systemu ubezpieczeń społecznych. Dlaczego, będąc w rządzie, nie wykazywał pan inicjatywy rządowej w sprawie emerytur stażowych? Czy PiS nie chciał wówczas emerytur stażowych, skoro dzisiaj również nie ma opinii o danej sprawie i stanowiska? Pytanie do strony rządowej: Czy wydacie pozytywną opinię na temat obywatelskiego projektu ustawy, czy raczej będziecie państwo popierać projekt prezydencki? Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt może być dobrym projektem, ale muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki. Po pierwsze, ciągłe budowanie świadomości emerytalnej, a po drugie, zachęty. Mówię o ciągłym budowaniu świadomości, żeby ludzie dokładnie wiedzieli - jeśli pójdą wcześniej na emeryturę - jakie będą brać później emerytury. To ma być permanentny proces uczenia. Mamy w tym zakresie dość duże zaległości. Drugi element, proszę państwa. Mają być wszelkiego rodzaju zachęty.

Bo stosunek ludzi pracujących do niepracujących będzie się pogarszał. Mówię o tym celowo, bo niektórych danych nie da się zafałszować.

W ostatnim okresie - mówię o generalnym ubóstwie - liczba ta wzrosła o 400 osób. Do tego nie możemy dopuścić. Dziękuję bardzo. Pan poseł Przemysław Koperski, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Część moich kolegów się skusiła.

Dzisiaj zbliżają się do pięćdziesiątki. Mam pytanie do przewodniczącego i do pana ministra. Do pana przewodniczącego: Czy ma wiarę w to, że w tym Sejmie znajdzie się większość, która poprze te dobre rozwiązania? Do pana ministra: Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze emeryturę stażową? Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, na te wszystkie pytania postara się odpowiedzieć sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed, a na te, na które nie da odpowiedzi dziś, pewnie prześle odpowiedzi na piśmie w późniejszym terminie. Panie Marszałku! Panie Przewodniczący wraz z Całym Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej! Wysoki Sejmie! Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym rodakom, którzy podpisali się pod projektem. To prawie 240 tys. obywateli, którzy wyrazili swój pogląd.

Nie ma w tej chwili jeszcze stanowiska rządu. Ono jest opracowywane w naszym ministerstwie, ale generalnie chcemy na ten temat dyskutować, bo sprawa jest ważna.

Pan poseł Tomaszewski zapytał mnie o emerytury pomostowe.

o których tutaj była mowa w tych przykładach, skorzystałyby z wcześniejszych rozwiązań, które dotyczyły pracy w warunkach szczególnych czy o szczególnym charakterze. Zmiana ustawy, wprowadzenie emerytur pomostowych w znaczny sposób ograniczyło możliwość przechodzenia. W 2012 r. ta sama koalicja podwyższyła wiek emerytalny, odrzuciła wniosek o referendum. Też nie zapytaliśmy wtedy, bo nie było takiej szansy, nie daliście jej państwo, żebyśmy zapytali obywateli, jak system emerytalny powinien w Polsce wyglądać. Myślę, że jest dzisiaj taki moment na bazie tego projektu, żeby się zastanowić, czy jeśli chodzi o system, który od 1998 r. w Polsce funkcjonuje, czyli tzw. zdefiniowanej składki, czyli im więcej odkładamy, dłużej pracujemy, tym mamy wyższe świadczenie, czy jeszcze do tego komponent stażowy jest potrzebny. I w tym projekcie to jest pokazane.

Pracujesz krótko, nie masz stażu i od tego masz obliczaną emeryturę. Ich przybywa więcej, bo jest większa liczba osób, która nabywa prawa emerytalne. Stąd było kilkanaście tysięcy, a teraz jest ich kilkaset tysięcy.

A więc mamy zdefiniowaną składkę, ale jest ten komponent stażowy, czy jego przywracamy. Pan prezydent faktycznie zaproponował trochę inne wysokości stażu, ale dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych.

To jest kwestia, jak myślę, do dyskusji. Jak wpłynie projekt prezydencki, myślę, że również wspólnie, razem będzie to rozpatrywane.

I też pokazują dzisiejsze badania, dzisiejsze dane, które też tutaj mam, wyliczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wzrasta nam liczba osób, które po przejściu na emeryturę podejmują dalszą pracę.

Rozwiązanie, które przyjęliśmy w tym roku w Polskim Ładzie, tzw. podatek zerowy dla seniorów, też ma ten cel, czyli osoba, która nabyła prawa do emerytury, ale nie przejdzie na emeryturę, będzie od nowego roku zwolniona z podatku.

Oczywiście tutaj były różne pytania.

To też pokazuje, że zależało nam na tym, aby najniższe świadczenia wzrastały, jak też oczywiście waloryzacja kwotowo-procentowa.

Jeśli chodzi o koszty, bo to wielokrotnie przebijało w tej dyskusji, oczywiście mamy przygotowane, tak jak też tutaj pan minister Marcin Zieleniecki już przedstawiał, dla tak jakby dwóch grup, czyli 100% osób korzysta z tych rozwiązań i na poziomie 50%.

Padło też pytanie o emerytury KRUS-owskie.

Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj precyzyjnie nie da się określić, jakiej grupy to dotyczy i jakie też będzie pojedyncze świadczenie, bo to wynika z indywidualnego wyliczenia dla poszczególnej osoby, która by przechodziła na emeryturę.

W trybie sprostowania poprosił o głos pan poseł Tadeusz Tomaszewski z klubu parlamentarnego Lewica. Bardzo proszę, panie pośle.

Tylko tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Marcina Zielenieckiego o zabranie głosu.

Bardzo dziękuję, na to liczyłem, szczerze mówiąc. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałem podziękować za merytoryczną dyskusję nad, przypomnę, obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającym emerytury stażowe.

Najczęściej chyba przewijał się wątek przesłanki uzależniającej prawo do emerytury stażowej od wypracowania kapitału czy wkładu emerytalnego, pozwalającego na ustalenie emerytury w kwocie najniższego świadczenia emerytalnego. Dość często też pojawiał się wątek dotyczący właśnie tych niskich świadczeń, tego, czy są w tym projekcie zabezpieczenia dla osób, których świadczenie może być niskie. A więc właśnie ta przesłanka, przesłanka uzależniająca możliwość przejścia na emeryturę stażową od posiadania prawa do emerytury w kwocie najniższego świadczenia, właśnie pełni taką rolę osłonową. Ona ma zapobiegać temu, aby te świadczenia stażowe nie były świadczeniami głodowymi, jak to się niekiedy mówi. Tylko osoby, które osiągnęły długi staż, ale jednocześnie opłacały składki od wynagrodzeń osiąganych w takiej wysokości, w której przejście na emeryturę pozwala po prostu na ustalenie tego świadczenia w kwocie minimalnego świadczenia, nabędą prawo do emerytury. Oczywiście te świadczenia będą ustalane - tutaj macie państwo rację - według formuły zdefiniowanej składki. Wiemy, jak ta formuła działa, wiemy, że wysokość świadczenia w tym systemie zależy od wartości wkładu emerytalnego, czyli wysokości składek wniesionych w okresie aktywności zawodowej, ale ten proponowany staż, w przypadku kobiet - 35 lat, w przypadku mężczyzn - 40 lat, jest gwarancją tego, że ten wkład będzie odpowiednio dużej wartości. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o drugi element tej formuły zdefiniowanej składki, bo przecież emeryturę obliczamy, dzieląc ten wkład emerytalny przez średnie dalsze trwanie życia osób w wieku osoby przechodzącej na emeryturę wyrażone w miesiącach.

Tutaj zgadzam się z państwem, że osoby, które spełnią te wymagania stażowe, będą musiały podjąć indywidualną, świadomą decyzję co do tego, czy w tym konkretnym momencie decydować się przejść na emeryturę, czy też poczekać.

Każda z tych decyzji jest decyzją indywidualną.

Od pracownika zależy, czy chce pracować dłużej i uzyskać świadczenie emerytalne w wyższej wysokości, czy też, kierując się innymi względami, zdecyduje się przejść na emeryturę wtedy, kiedy spełni warunki stażowe.

Nie mamy do czynienia z dyskryminacją osób, które studiowały.

Nie proponujemy w nim tylko tego, aby osoby, które były ubezpieczone z tytułu pozostawania w stosunku pracy, miały uprawnienie do emerytury stażowej. To jest projekt adresowany do różnych kategorii ubezpieczonych, w tym osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Było pytanie dotyczące liczby osób, które skorzystają czy będą mogły skorzystać z rozwiązań zawartych w obywatelskim projekcie ustawy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w opinii dotyczącej tego projektu szacuje liczbę takich osób na 470 tys.

Państwo pamiętają treść art. 39 Kodeks pracy. Wiemy, że Kodeks pracy zapewnia szczególną ochronę trwałości stosunku pracy osobom, które są w wieku niższym o 4 lata od wieku emerytalnego. W tym zakresie ten projekt niczego nie zmienia.

Myślę, że te przykłady, które podawałem, prezentując projekt ustawy, są dość wymowne.

Historia każdego z ubezpieczonych jest inna, różna jest sytuacja materialna, sytuacja rodzinna, różny jest punkt startu, różna jest wysokość wynagrodzeń, ale możemy dzięki temu sobie wyobrazić, jakie kategorie osób mogą czy będą mogły skorzystać z dobrodziejstwa emerytury stażowej. Mianowicie uważam, że ten wątek, który się pojawił w dyskusji, o edukacyjnym, wychowawczym charakterze emerytury stażowej jest bardzo ważny, dlatego że model zatrudnienia, który przedstawiłem: wczesny start, nieprzerwana praca przez wiele dziesiątek lat, bardzo często praca na jednym stanowisku pracy bez względu na warunki pracy, jeżeli chodzi o młode pokolenia - państwo też tutaj kilkakrotnie ten wątek przywoływaliście, mówiąc o repartycyjnym systemie ubezpieczenia społecznego - wcale nie jest, że tak powiem, chętnie przyjmowany.

Na koniec chcę podziękować przede wszystkim panu ministrowi za słowa, za deklarację dotyczącą przystąpienia do prac nad projektem ustawy, przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych za życzliwość i przychylność dla tego projektu.

Dziękuję serdecznie. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań.

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Pan poseł Tomasz Zieliński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tuż przed ogłoszeniem kolejnej edycji programu Polski Ład warto kilka słów powiedzieć o wielkości środków pozyskanych przez samorządy z terenu Zamojszczyzny w ramach pierwszego naboru w zakresie Programu Inwestycji Strategicznych. Dzisiejsza Zamojszczyzna to 55 samorządów, w tym 50 gmin wiejskich i miejskich, cztery starostwa powiatowe oraz jedno miasto na prawach powiatu. Jest to teren, na którym samorządy muszą systematycznie odrabiać zapóźnienia gospodarcze i społeczne, szczególnie w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowej, wodociągów, kanalizacji, modernizacji szkół i placówek oświatowych, bibliotek, domów kultury oraz szeregu budynków użyteczności publicznej, takich jak świetlice wiejskie czy remizy strażackie. Wielkość budżetów szczególnie małych wiejskich gmin uniemożliwia przeprowadzenie samodzielnie takich inwestycji, tak bardzo potrzebnych mieszkańcom, których celem jest ogólnie rozumiana poprawa życia lokalnej społeczności. Ogłoszenie w lipcu tego roku pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego był odpowiedzią na potrzeby samorządów Zamojszczyzny, tym bardziej że w skali kraju przeznaczono na bezzwrotne dotacje 23 mld zł. Wnioski można było składać zgodnie z ustalonymi kryteriami w ramach czterech priorytetów, zaś wkład własny samorządu wynosił w zależności od wartości zadania inwestycyjnego od 5% do 20%.

W poszczególnych powiatach dotacje wyniosły: w powiecie biłgorajskim - ponad 107 mln, hrubieszowskim - 66 mln, tomaszowskim - 86 mln, zamojskim - 97 mln, zaś miasto Zamość otrzymało 23 mln zł. Należy podkreślić, że dotacje, wbrew obawom polityków opozycji, otrzymały wszystkie samorządy i nikt podczas oceny wniosków nie brał pod uwagę poglądów politycznych ich włodarzy. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych na Zamojszczyźnie zrealizowanych zostanie 96 projektów z różnych dziedzin. Rzeczywiście dominują inwestycje związane z budową i modernizacją dróg gminnych i powiatowych, budową wodociągów i kanalizacji, modernizacji oczyszczalni ścieków, budową przedszkoli, boisk sportowych oraz wiele, wiele innych. Podczas akcji przekazywania symbolicznych czeków samorządowcom oraz podczas spotkań ogromna większość z nich podkreślała wyjątkowość tego programu. Po pierwsze, ilość otrzymanych środków jest bardzo duża, w wielu przypadkach sięga połowy aktualnego budżetu gminy. Po drugie, niewielki wkład własny umożliwia gminie, nawet będącej w trudnej sytuacji finansowej, realizację planowanej inwestycji. Po ogłoszeniu wyniku wspomnianego wyżej naboru w ciągu tygodnia samorządy otrzymały kolejne bardzo dobre informacje. Zgodnie z założeniami rząd premiera Mateusza Morawieckiego postanowił wesprzeć projekty wodno-kanalizacyjne dodatkową kwotą 4 mld zł.

W ramach tego programu gminy z terenu Zamojszczyzny otrzymały ponad 135 mln zł bezzwrotnej dotacji z podziałem na inwestycje związane z wodociągami, z zaopatrzeniem w wodę - ponad 40 mln zł, oraz inwestycje kanalizacyjne - ponad 95 mln zł. Program Inwestycji Strategicznych uruchomiony w ramach programu Polski Ład jest ogromną szansą dla mieszkańców całego kraju, ale w szczególności dla terenów Polski wschodniej, gdzie występują bardzo duże braki w zakresie infrastruktury. Jako mieszkaniec Lubelszczyzny głęboko wierzę, że kolejne edycje tego programu definitywnie zlikwidują dysproporcje rozwojowe występujące pomiędzy poszczególnymi obszarami naszego państwa. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub parlamentarny Lewica.

Moje oświadczenie dotyczy zaniedbań ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad związanych z przebudową i remontem drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno - Żydowo - Czeluścin. Kilka lat wcześniej generalna dyrekcja dróg krajowych przeprowadziła remont pierwszego odcinka drogi, Września - Czeluścin.

Wiele tych uzgodnień niestety traci już swoją ważność ze względu na upływ czasu.

Po drugie, ten odcinek drogi łączy dwa ośrodki, jest to droga również w kierunku na Wrocław. Z tej drogi korzystają też mieszkańcy tamtej części Polski, przemieszczając się, krótko mówiąc, nad morze. Dlatego też od kilku lat czynię starania, wspólnie z przedstawicielami samorządów, aby remont tej drogi został przeprowadzony wcześniej. Jest jakaś nadzieja, bo jak informują media, został przeprowadzony przetarg na wykonanie dokumentacji i uzgodnień administracyjnych w zakresie przebudowy tego odcinka drogi. Niemniej jednak zapowiedź mówiąca o tym, że dopiero w 2023 r. ma być prowadzona ta inwestycja, mieszkańców i samorządowców nie satysfakcjonuje. Dlatego też po raz kolejny 3 grudnia pozwoliłem sobie złożyć interpelację do ministra infrastruktury.

Bardzo na to liczę i wnoszę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o poinformowanie o sposobie załatwienia tej interwencji w ramach odpowiedzi na interpelację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Bartłomiej Dorywalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Strajk w obronie krzyży we Włoszczowie. W okresie PRL krzyże pojawiły się w szkołach, gdy powstawała „Solidarność”, w 1980 i 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego władze powróciły jednak do ateizacji społeczeństwa. Ze szkół zaczęto usuwać symbole wiary i tak było we Włoszczowie. W piątek 30 listopada 1984 r. młodzież postanowiła bardzo uroczyście poświęcić krzyże w miejscowym kościele.

W dłoniach nieśli drewniane krzyżyki, takie jakie zwyczajowo wiesza się nad drzwiami w domach. W tym czasie w szkole zorganizowano dyskotekę. Uczniowie ją zignorowali, wybierając wieczorne nabożeństwo. Podczas mszy ówczesny ksiądz proboszcz Kazimierz Biernacki poświęcił krzyże i tłumaczył młodym ludziom, jaką odpowiedzialność biorą na siebie, niosąc krzyż Chrystusowy. W sobotę krzyże zawisły w klasach. Młodzi ludzie modlili się i śpiewali pieśni kościelne, dawali nauczycielom krzyże do pocałowania i dopiero wieszali nad drzwiami. Ponowne zdjęcie krzyży ze ścian doprowadziło do protestu, który przybrał formę strajku. W dniu 3 grudnia 1984 r. ówczesny dyrektor szkoły Julian Lis podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu zajęć szkolnych i wezwał młodzież do opuszczenia budynku szkoły. Młodzież nie podporządkowała się temu zarządzeniu i ok. 200 osób, w tym dwaj księża, Marek Łabuda i Andrzej Wilczyński, pozostało w szkole, domagając się ponownego zawieszenia w salach lekcyjnych krzyży usuniętych na polecenie dyrekcji. Drogi dojazdowe do Włoszczowy zostały obstawione przez patrole ZOMO. Funkcjonariusze legitymowali osoby wjeżdżające, niejednokrotnie blokując możliwość jakichkolwiek kontaktów ze stroną strajkującą. Część nauczycieli, zwolenników dyrektora Lisa, odwiedzała domy uczniów i namawiała rodziców, żeby zabrali swoje dzieci ze szkoły. Lokalna społeczność solidaryzowała się ze strajkującymi, do szkoły zanoszono wyżywienie oraz odzież. Sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz bardziej tragiczna. Niepewność, ciągłe oczekiwanie na wiadomości ze strony uczniów, spowodowała, że rodzice wystosowali petycję do ministra oświaty. Niestety nic ona nie dała. W obawie o uczniów, a także o swoją przyszłość nauczyciele prosili, aby doprowadzić do zakończenia strajku. Niektórzy rodzice nawet siłą zabierali dzieci do domu. Ostatecznie w szkole zostało ok. 80 osób. Tego dnia do Włoszczowy przybył bp Mieczysław Jaworski i dziękował młodzieży za dojrzałą postawę. Od szkoły do pobliskiego kościoła ruszyła procesja z krzyżami, po drodze dołączali do niej mieszkańcy Włoszczowy. Na represje ze strony szkoły nie trzeba było długo czekać. Na zwołanej po świętach radzie pedagogicznej podjęto decyzję o wyrzuceniu Renaty Gałkiewicz ze szkoły. Anna Synowska i Mariola Lewicka zdały maturę dopiero kilkanaście lat później. Z pracy próbowano zwolnić nauczyciela Kazimierza Ostrowskiego, jednak po odwołaniu od wypowiedzenia decyzję cofnięto. Władze szkolne nie wywiązały się z wcześniejszych zapewnień o braku stosowania represji wobec strajkujących, wręcz przeciwnie, byli oni szykanowani. Z kolei uczestniczący w strajku duchowni stanęli przed sądem i zostali zmuszeni do wyjazdu za granicę, na misje do Afryki. Od wydarzeń z tamtych lat minęło już 37 lat. Wielu z uczestników strajku już nie żyje. Ciężko jest odpowiedzieć za nich, czy dzisiaj, znając konsekwencje tych czynów, zdecydowaliby się na taki akt jak wtedy, w grudniu 1984 r. Ci, którzy pozostali, zapewniają, że tak. Pamięć o tych wydarzeniach wśród włoszczowian jest wiecznie żywa, czego wyrazem były uroczyste obchody, jakie miały miejsce w dniu 3 grudnia br. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie w województwie kujawsko-pomorskim przekazał następujący komunikat: Informujemy, że planowana wypłata świadczenia wychowawczego 500+ w dniu 14 grudnia 2021 r. będzie zrealizowana w późniejszym terminie, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z urzędu wojewódzkiego. Panie i Panowie Ministrowie! To jedna z najmniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Panie i panowie ministrowie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla niektórych liczy się każdy grosz. W związku z tym mam pytanie: Kiedy beneficjenci programu 500+ z gminy Świekatowo otrzymają należne środki, by godnie przygotować święta Bożego Narodzenia? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Dzisiaj dzięki wygranemu głosowaniu podczas posiedzenia połączonych komisji edukacji i Komisji Obrony Narodowej opozycji udało się zablokować prace nad fatalnym projektem ustawy o zmianie Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. To mały sukces opozycji, ale wielkie zwycięstwo wszystkich, którzy protestowali przeciwko tym zmianom, przede wszystkim rodziców, nauczycieli i uczniów. Szanowni Państwo! Dlaczego wbrew deklaracjom Ministerstwa Edukacji i Nauki o odbiurokratyzowaniu pracy szkół i placówek projekt zmian w Prawie oświatowym procedowany w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zawiera rozwiązania wymuszające gromadzenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wdrożenia zajęć dodatkowych, uzupełniających, projektów edukacyjnych wzbogacających ofertę edukacyjną szkół i placówek publicznych? Ujęte w ramy prawne procedury administracyjne utrudniające prace nad budowaniem dobrej szkoły świadczą o braku zaufania aktualnie rządzących do dyrektorów szkół i placówek, do nauczycieli i rodziców uczniów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Lorek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stan wojenny na ziemi piotrkowskiej. Zakłady przemysłowe ziemi piotrkowskiej bardzo wcześnie włączyły się w ogólnopolski ruch niepodległościowy, którego finałem było utworzenie na podstawie tzw. porozumień sierpniowych „Solidarności” 8 sierpnia rozpoczął się strajk w Zakładzie Transportu i Sprzętu Technologicznego przy KWB Bełchatów. Protestowano w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Fale strajków przetaczały się przez region od września do listopada 1980 r. Zazwyczaj kończyły się podpisaniem porozumień, które zapewniały, iż postulaty płacowo-socjalne robotników będą realizowane. Stopniowo też tworzyły się w różnych zakładach pracy zalążki komórek niezależnych związków zawodowych. W połowie stycznia miały już ok. 44 tys. członków. Przez cały okres „Solidarności” prowadzono różnego rodzaju działalność protestacyjną. Największe zgromadzenie odbyło się 30 lipca w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w manifestacji, która zakończyła się przed budynkiem urzędu wojewódzkiego, wzięło udział 4 tys. ludzi. W zakładach utrzymywano gotowość strajkową, atmosfera nabrzmiewała. W nocy z 12 na 13 grudnia milicja i Służba Bezpieczeństwa rozpoczęły aresztowania. Zabrzmiała groźna fraza: stan wojenny.

Do takich osób należał Adam Trybus, dawny cichociemny, człowiek wtedy już ciężko chory, represjonowany w okresie stalinowskim.

Był to protest przeciwko jego wprowadzeniu. Zarówno rodziny internowanych, jak i oni sami otrzymali pomoc od pozostających na wolności działaczy „Solidarności” oraz od Kościoła katolickiego.

Działalność niepodległościową przeniesiono do podziemia. Wydawano wiele tytułów prasy, były także periodyki, które ukazywały się nieregularnie, ponieważ ich redakcje były permanentnie inwigilowane i zamykane. W Piotrkowie Trybunalskim powstało Duszpasterstwo Ludzi Pracy, na zaproszenie którego po mszach św. za ojczyznę odbywały się spotkania, na których bywali m.in. Jan Olszewski, Jerzy Kropiwnicki czy Kornel Morawiecki. Motywy jego wprowadzenia do dziś są badane przez historyków i nadal budzą wielkie emocje. Dziękuję bardzo. Pan poseł Aleksander Mrówczyński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Samorządowiec, radny Rady Powiatu Starogardzkiego, radny rady miasta, społecznik. Człowiek serdeczny, skromny, pełen empatii, bardzo oddany małej i tej dużej ojczyźnie, oddany Bogu.

Przez cały czas pracy w Sejmie VIII kadencji przy każdej możliwej okazji przekonywał o konieczności budowy obwodnicy.

Przygotowaliśmy wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury w maju 2017 r. w jego mieście, w Starogardzie Gdańskim, i w Chojnicach. Pragnę dodać, że w naszych miastach nigdy wcześniej nie było posiedzenia komisji sejmowej. W czasie tych 2 dni, bo było to dwudniowe wyjazdowe posiedzenie, dyskutowaliśmy o wykluczeniu komunikacyjnym, o planach związanych z drogą krajową nr 22, o jego obwodnicy, obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

Wieniec na grobie złożył m.in. wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.

Niestety z powodu choroby i złego samopoczucia nie mogłem uczestniczyć w rocznicowych obchodach, czego bardzo żałuję. W moim imieniu głos zabrał wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk. W uroczystościach wzięła udział rodzina oraz m.in. pan poseł Kazimierz Smoliński, działacze Prawa i Sprawiedliwości ze Starogardu Gdańskiego i z Tczewa. Janku, spoczywaj w pokoju. Bardzo mi ciebie brakuje.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Kryj, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku lat 80. XX w. największym pracodawcą w Ostrowcu Świętokrzyskim, a jednocześnie najsilniejszym zakładem pracy w strukturze świętokrzyskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” była Huta im. Marcelego Nowotki. W tzw. starym i nowym zakładzie huty pracowało wówczas 16 tys. osób, spośród których zdecydowana większość należała do związku.

Jego wybuch należy wiązać z internowaniem przywódców ostrowieckiej „Solidarności”, jakie miało miejsce nocą z 12 na 13 grudnia. Łącznie na terenie miasta zatrzymano ponad 20 osób, wśród których byli m.in. Wiesław Standzikowski, Henryk Gruszka, Robert Minkina, Adam Mitura, Józef Gurczyński i Henryk Nawojski. Internowania rozpoczęły się o północy i trwały do godz. 3 nad ranem. Pierwszymi spośród osób, które zostały poinformowane o zatrzymaniu związkowców, byli ich koledzy dyżurujący w Delegaturze Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na osiedlu Ogrody: Marceli Czarnecki, Tadeusz Kiełkiewicz, Mieczysław Kadewski, Józef Fudala. To do nich ok. godz. 1 dotarli bliscy internowanych, którzy opowiedzieli o brutalności działań milicjantów. Po ich wysłuchaniu dyżurujący w siedzibie delegatury rozeszli się po mieście, aby informować o zachodzących wydarzeniach innych działaczy związku. Niezależnie od nich akcję ostrzegawczą zorganizowała Wiesława Standzikowska, żona internowanego szefa hutniczej „Solidarności”, która powiadomiła o tym Zygmunta Jakubowskiego i Wiesława Kwiatkowskiego. W ten sposób powiadomieni zostali również Stefan Kowalski i Waldemar Gomuła. Dzięki akcji ostrzegawczej kilku czołowych działaczy „Solidarności” hutniczej uniknęło internowania i większość z nich znalazła się na terenie swoich zakładów pracy, gdzie włączyli się w organizację strajku. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób.

Hutnicy zawiązali wówczas komitet strajkowy, który następnie przekształcił się w komitet ocalenia związku. Powołali straż robotniczą i ogłosili postulaty, wśród których znalazło się m.in. żądanie uwolnienia internowanych kolegów. Epilogiem tego strajku były procesy wytoczone przywódcom i szczególnie aktywnym uczestnikom strajku. Należeli do nich Marceli Czarnecki, Andrzej Dudek, Jerzy Jabłoński, Tadeusz Stasiowski, Jerzy Borowiec, Henryk Piątek, Marian Susfał, Jan Szaran, Andrzej Wójcik, Janusz Ziajski i Józef Fudala. Kolejnymi osobami skazanymi na kary więzienia za działalność w strukturach podziemnej „Solidarności” byli Leszek Olszewski, Krzysztof Partyka, Jarosław Salita, Ryszard Sobala, Zbigniew Walczyk i Andrzej Żółciński. Osób prześladowanych, m.in. zwolnionych z pracy było znacznie więcej. W dniu 10 grudnia staraniem działaczy Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989” Jerzego Jabłońskiego, Wiesława Kwiatkowskiego, Mieczysław Dudka, Krzysztofa Mikosa, Stanisława Oleszka, Tadeusza Relikowskiego, Wojciecha Krasuskiego, Marka Kolczugi i Jana Kaptura w Ostrowieckim Browarze Kultury została otwarta wystawa „40-lecie wprowadzenia stanu wojennego” Wieczorem 13 grudnia w kościółku hutniczym odprawiona została msza święta, a następnie przeszedł marsz pamięci ofiar stanu wojennego. Jego uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową na rondzie „Solidarności” Chwała bohaterskim ostrowieckim hutnikom, którzy sprzeciwili się wprowadzenia stanu wojennego. Chwała bohaterom walki o wolną Polskę. Dziękuję bardzo. Pan poseł Maciej Kopiec, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Alert RCB to wiadomości SMS, które wysyłane są tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie i zdrowie ludzi. Tak opisany jest przez rząd na oficjalnej stronie internetowej. Wczoraj mieszkańcy Rybnika otrzymali alert o treści: Uwaga! Dnia 13 i 14 grudnia prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. To kuriozalne, że rząd ostrzega przed nieudolnością rządu, która to nieudolność zagraża zdrowiu i życiu obywateli. Katowice i Kraków wprowadziły dziś bezpłatną komunikację miejską po to, by ograniczyć emisję, co powoduje, że po raz kolejny koszty nieudolności rządu będą ponosiły samorządy.

Jeśli nic się nie zmieni, do końca jego trwania wydamy zaledwie 9 mld. Zmarnujecie państwo 90% zaplanowanych środków. To jest prawdziwa miara waszej efektywności i troski o zdrowie ludzi. Kilka dni temu, 9 grudnia zapadł wyrok w prawie Oliwera Palarza z Rybnika, który wykazał przed sądem częściową utratę zdrowia oraz ograniczenie wolności ze względu na panujący smog. Z wyroku wynika więc jasno, że państwo narusza dobra osobiste obywateli. Ponadto art. 38 konstytucji mówi jasno o tym, że państwo polskie zapewnia wszystkim obywatelom prawną ochronę życia. Tymczasem dziecko idące do szkoły oddycha powietrzem porównywalnym do palenia papierosów. Polski Alarm Smogowy w grudniu ub.r. obliczył, że w województwie śląskim trzeba będzie wymienić 140 tys. kotłów. Głównym powodem, dla którego Polacy nie zmieniają źródła ogrzewania i energii, są ceny. To nie jest tak, że oni to robią na złość. Ich po prostu na to nie stać. W budżecie Polski są tylko jedne pieniądze i to wyłącznie od PiS zależy, jak są wydawane. Fakty. Centralny Port Komunikacyjny - budżet 35 mld zł. To 350 tys. ekologicznych źródeł ciepła połączonych z OZE. To 180 tys. źródeł ciepła. To 25 tys. źródeł ciepła. To 20 tys. źródeł ciepła. W 30 s znalazłem źródła finansowania dla ponad pół miliona nowoczesnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych. Polski Alarm Smogowy w zeszłym roku obliczył, przypominam, że w samym województwie śląskim należy wymienić 140 tys. kotłów. To tak dla wskazania skali. Ale rząd zamiast zająć się czystym powietrzem załatwia spółce Solorz - Obajtek monopol na ogrzewanie atomem, żeby przypadkiem nikt nie zrobił tego taniej i lepiej. Jednym z filarów Funduszu Odbudowy jest transformacja energetyczna i zielone źródła energii. Państwo jeździcie po Polsce i rozdajecie bony na pieniądze z tego funduszu, tymczasem to czeki bez pokrycia. Tych pieniędzy nie będzie przez łamanie praworządności, przez ksenofobię, przez wasz kierunek na polexit. Wiecie już, że wasz upór w demontażu praworządności odebrał Polsce 770 mld zł. Premier Morawiecki jest już tak zrozpaczony, że wysyła SMS-y do polityków europejskich, podpisując się: ostatni Europejczyk w tym rządzie. Jak nisko trzeba upaść? Takie są konsekwencje konszachtów z Orbánem i Le Pen i wygłaszania bzdur. Veto albo śmierć. Będzie śmierć wywołana chorobami spowodowanymi oddychaniem powietrzem, które zabija, i to wy jesteście za to odpowiedzialni. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Zapraszam, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Są w historii sztuki postaci cokolwiek kontrowersyjne, np. Daniele da Volterra, przyjaciel i uczeń Michała Anioła, który w XVI w. na polecenie papieża Pawła IV domalował elementy garderoby na słynnym fresku „Sąd ostateczny”, albo np. papież Pius IX, który w połowie XIX w. zasłynął tym, że podobno własnoręcznie dłutem odrąbywał elementy przyrodzenia wszystkim rzeźbom znajdującym się w państwie kościelnym. Do tego niesławnego panteonu dołączyła ostatnio dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach, pani Maria Czarnecka. Oto podczas 11. Triennale Grafiki Polskiej w tymże muzeum zauważyła, że jedna z prac jest zatytułowana w sposób, który uwzględnia hasło: lex Szyszko. Była to praca pana Michała Krawca, jednego z polskich grafików, kolaż przedstawiający maszyny do wycinania drzew na tle stalowych, poprzemysłowych budynków. Tego nie ma tutaj być, tego nie może tu być, przez takie postawy pan prof. Szyszko nie żyje - miała powiedzieć dyrektorka i nakazać pracownikom Muzeum Śląskiego natychmiastowe wydrapanie ze ściany tego właśnie elementu nazwy. Nie zezwolę na rozpoczęcie konferencji prasowej otwierającej triennale, jeżeli ta nazwa, ten napis natychmiast nie zniknie. Przypomnijmy, że chodziło o tytuł grafiki jednego z uczestników triennale. Ze zdumieniem ostatnio usłyszałem, że pan marszałek województwa śląskiego kompletnie tą sytuacją zainteresowany nie jest. Mówi: nie było mnie tam, nie mam nic wspólnego z tą wystawą, nie mam bladego pojęcia, dlaczego pani dyrektor zachowała się właśnie w taki sposób. Poprzednią dyrektorkę Muzeum Śląskiego odwołał. Co istotne, po sądowej batalii okazało się, że odwołał ją z poważnym naruszeniem prawa. Zarzucał jej zresztą niekompetencję. Jak bardzo była niekompetentna, świadczy jej obecna praca. Poprzednia dyrektorka Muzeum Śląskiego jest dziś szefem Galerii Narodowej w Pradze - czeskiej Pradze, wybranym oczywiście w konkursie. Bracia Czesi bardzo są dumni z jej pracy.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 10 grudnia obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka. To święto ustanowione w rocznicę przyjęcia w 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To dokument niezwykle ważny dla wszystkich, myślę, ludzi na świecie. Ogłoszono w nim niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej, niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy też innego statusu. W tym dniu szczególnie pamiętamy o orędownikach praw człowieka, którzy dążą do zapewnienia ochrony praw własnych oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawionych pracy czy niesłusznie więzionych. Z okazji święta pamiętamy o ich odwadze i osiągnięciach. Ale to też okazja do refleksji, na ile nasz stosunek do innych ludzi wyraża nasze człowieczeństwo. Dziś jest to pytanie niezwykle aktualne, dlatego zachęcam, aby sięgnąć do deklaracji i odkryć ją dla siebie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Waldemar Andzel. No to mnie martwi ta absencja. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Składam oświadczenie w sprawie zmiany przepisu dotyczących dodatków COVID-owych dla pracowników medycznych. Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące rozliczania dodatków COVID-owych przewidują, że są one wypłacane za każdą godzinę opieki nad pacjentem z COVID-19 lub podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dodatki stanowią 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej należnego za każdą godzinę pracy, ale maksymalna miesięczna kwota nie może być wyższa niż 15 tys. zł. Muszą być też spełnione wymagane kryteria. Kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie: a) wykonuje zawód medyczny; b) uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2; c) pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, tzw. II poziom zabezpieczenia COVID-owego. Oświadczam, że wysoce niesprawiedliwe jest pominięcie tysięcy pracowników, którzy nie spełniają wymogu z pkt c. Wymóg mówiący o bezpośrednim kontakcie z pacjentem wykluczył z dodatków diagnostów laboratoryjnych, którzy takiego kontaktu nie mają, choć codziennie w swojej pracy każdy z nich ma kontakt z materiałem zakaźnym osób chorujących na COVID-19. Tysiące pracowników ochrony zdrowia codziennie i z poświęceniem biorą czynny udział w procesie leczenia chorób, również narażając swoje życie i zdrowie. Ich praca wygląda tak samo jak pracowników będących pracownikami tzw. oddziałów COVID-owych: wielogodzinne noszenie kombinezonów, używanie szkodliwych środków do dezynfekcji itp. Pracownicy, którzy zostali wykluczeni według nowych zasad rozliczenia dodatków COVID-owych dla medyków, to: pracownicy pracowni diagnostycznych - podstawą leczenia COVID-19 jest diagnostyka obrazowa układu oddechowego: badanie tomografii komputerowej płuc, zdjęcia RTG i wiele innych - pracownicy pracowni endoskopii i pracownicy bloków operacyjnych. Wymienieni pracownicy zmagają się z czwartą falą. Wykonują ponad 100 tys. testów na dobę. Do tej pory wykonali 20 mln testów w kierunku COVID-19. Powyższe statystyki pokazują, że nie ma wątpliwości co do zasadności włączenia tej grupy medyków i tej grupy zawodowej do katalogu uprawnionych, którzy powinni otrzymać dodatek COVID-owy. Oświadczam, że grupa pracowników pracowni diagnostycznych, pracowni endoskopii i pracowników bloków operacyjnych została wykluczona z otrzymywania dodatku COVID-owego, mimo że codziennie w takim samym stopniu jest narażona na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Świadczenia za miesiąc październik nie zostały wypłacone powyższym pracownikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dla mnie jako posła z Pomorza najważniejsze są oczywiście inwestycje w województwie pomorskim, więc co roku zabiegam o te najważniejsze, które są zgłaszane przez mieszkańców.

Obydwa węzły ze względu na swoją niewymiarowość mają bardzo złą widoczność, co utrudnia kierowcom włączanie się do ruchu. Ponadto obydwa węzły nie są przystosowane do ruchu rowerowego i pieszego.

Zarówno mieszkańcy, jak i miasto Gdańsk od lat zabiegają o budowę tych węzłów. Niestety koszt ich rozbudowy przekracza możliwości finansowe miasta Gdańska. Apeluję więc do rządu PiS o akceptację tych poprawek i poparcie przeznaczenia pieniędzy na rozpoczęcie rozbudowy tych dwóch ważnych węzłów. Na posiedzeniu komisji finansów posłowie PiS, nawet ci z Pomorza, którzy tak bardzo w czasie kampanii wyborczej obiecywali pomagać mieszkańcom, niestety nie poparli tych dwóch poprawek. Brak słów. Dziękuję. Panie pośle, zapraszam. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 40 lat temu 13 grudnia 1981 r. w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Oczywiście było ich znacznie więcej, niemalże wszyscy zamordowani przez tzw. nieznanych sprawców byli rzeczywistymi ofiarami SB, MO lub ZOMO. Uważam, że 40. rocznica tego tragicznego dnia w polskiej historii jest doskonałą okazją, aby wszystkich odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego nazywać przestępcami lub sprawcami. Skończmy z retoryką nazywania bandytów architektami, twórcami czy autorami stanu wojennego. A doskonale wiemy, że towarzysze Kiszczak i Jaruzelski nie są jedynymi sprawcami. Pan Andrzej Kołodziej, działacz „Solidarności” i sygnatariusz porozumień sierpniowych, stwierdził, że wprowadzenie stanu wojennego było zdradą elit, w tym elit „Solidarności” Pięknym gestem upamiętniającym ofiary stanu wojennego było zapalenie w wielu miejscach na świecie świateł wolności. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.